Wysoka Izbo! Idzie jesień strajków. Ulicami Warszawy właśnie przeszedł wielki protest szeregowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, a to jest dopiero początek. Kuratorzy sądowi, inspekcje, kolejne grupy szeregowych pracowników budżetówki domagają się godnych płac. Za chwilę wybuchnie strajk w ZUS-ie i staną pod znakiem zapytania wypłaty 500+ i emerytur. Tutaj trzeba działać, szanowna strono rządząca, a nie chować głowę w piasek. Wysoka Izbo! Pracownicy budżetówki od lat padają ofiarą ideologii tzw. taniego państwa. Zwracam się tutaj do prawej strony sceny politycznej, bo kiedyś - i słusznie - krytykowaliście państwo, kiedy Tusk kazał zaciskać im pasa, ale teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości robi dokładnie to samo. Nie słuchacie tych ludzi, a to są ludzie, którzy ciężko i ofiarnie pracują dla polskiego państwa i zasługują na godne płace. Dlatego w imieniu klubu Lewicy składam wniosek o przerwę (Dzwonek) i uzupełnienie porządku obrad. Żądamy pilnego rozpatrzenia naszego projektu ustawy, który podnosi płace w budżetówce natychmiast, o przynajmniej 12%. O tym, co się znajdzie w porządku obrad, już zdecydowaliśmy, natomiast padł wniosek o przerwę. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Nie działa aparatura?

Sejm wniosek odrzucił. Z wnioskiem formalnym pani poseł Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Dla wielu z nas, przyjaciół, bliskich, to tragedia wiecznie żywa, to tragedia, o której nie możemy zapomnieć. Niestety, cały czas służy do politycznych rozgrywek. 36 dni temu obecny tutaj pan Antoni Macierewicz podobno ukończył raport. Panie Pośle! Mam prawo zobaczyć ten raport, a pan wybiera rodziny, którym pan go pokazuje. Jest pan szefem podkomisji. To pan nadzoruje Ministerstwo Obrony Narodowej. Rzeczpospolita, obywatelki i obywatele, a także rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej i przyjaciele mają prawo dowiedzieć się, co robiliście za publiczne pieniądze, jakie są ustalenia [[Oklaski]] i kto te ustalenia poczynił.

O co? O co wniosek formalny pani składa, pani poseł?

Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! Raport został przegłosowany przez całą komisję 10 kwietnia. Zostały one zaproszone na poniedziałek 2 dni temu.

Jeżeli można. Jeśli do pań nie dotarło to zaproszenie.

Wszyscy państwo będziecie mieli go do dyspozycji. Pani poseł, złożyła pani wniosek o przerwę.

Ale złożyła pani wniosek o przerwę, pani poseł.

Widzę, co pani złożyła na piśmie.

W takim razie ja składam wniosek o przerwę. W miniony piątek w Warszawie protestowali pracownicy sądów i prokuratur. Domagały się podwyżek, poszanowania, zwiększenia liczby etatów, godnych warunków pracy oraz podjęcia konkretnych działań w celu zaprzestania mobbingu w sądach. Do protestujących, którzy przyjechali do stolicy w ramach urlopu, nie wyszedł nikt z kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Protestowali przy zamkniętej twierdzy resortu. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości pojawili się przedstawiciele związków pracowników sądów i prokuratur, jednak minister Michał Woś nie zamierzał z nimi w Sejmie rozmawiać. Przedstawił tylko ogólne informacje na temat tego, jak w sądach jest świetnie, a potem opuścił salę, tłumacząc się naradą u premiera. To oznaka lekceważenia. Dlatego składam wniosek o przerwę w obradach, by minister, poseł Michał Woś.

Związkowcy zostali w Warszawie. Za kilka minut rozpocznie się posiedzenie komisji, więc panie ministrze, wysłuchajcie postulatów związkowców, pracowników sądów i prokuratur. Z wnioskiem przeciwnym pan minister Michał Woś. Wysoka Izbo! Chciałbym i z wnioskiem przeciwnym, i w trybie sprostowania, bo padły nieprawdziwe słowa.

Dialog.

Ponieważ padł wniosek formalny o odroczenie posiedzenia, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił.

Mam nadzieję, że ta ustawa już nigdy nie wróci do Sejmu, bo była zaiste szalona. Teraz druga szalona rzecz, która tutaj się odbyła dosyć po cichu przy sprzeciwie jedynie Grzegorza Brauna i Konfederacji.

To jest ustawa, która odwraca do góry nogami cały system podatkowy, to jest ustawa, po której miliony Polaków będą musiały zmieniać tryb swojego zatrudnienia. To jest ustawa, która milionom Polaków, którym wy chcecie dokopać, narzuci wyższe opodatkowanie.

O głos poprosił minister - członek Rady Ministrów pan Michał Wójcik. Proszę bardzo, panie ministrze.

Przepraszam, zapomniałem nazwiska. Otóż, szanowni państwo, państwo powinniście kierować swoje pretensje do Donalda Tuska. A dlaczego? Bo z tej mównicy wszyscy powinni wiedzieć o tym, ile w roku 2010. Donald Tusk dał pracownikom sądów i prokuratur. Zero złotych. Zero złotych. Zero złotych. Zero złotych. Proszę nie zakrzykiwać.

do tak trudnej sytuacji doprowadził rząd Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Taka jest prawda. A kuratorzy nam dziękują, tylko wy nie chcecie o tym mówić.

Proszę bardzo. Panie Ministrze! Ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że Donald Tusk postępował nie w porządku wobec budżetówki. Problem polega na tym, że weszliście w jego buty. A te podwyżki, o których pan mówi. Panie Ministrze! Proszę odpowiedzieć na pytanie.

Czcigodna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Działając na podstawie art. 43 ust. 6 regulaminu Sejmu, niniejszym przedstawiam sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy. Bardzo proszę państwa posłów niezainteresowanych tym punktem porządku dziennego o opuszczenie sali i umożliwienie panu posłowi sprawozdawcy przedstawienia sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Kwestia dotyczy druku nr 1368. Na skutek podejmowanych prac zarówno w podkomisji stałej do spraw zmian w nowelizacjach odnośnie do prawa karnego, jak i następnie już w komisji głównej w dniu 22 lipca 2021 r. udało się przedstawić finalny produkt legislacyjny, a tym samym przedstawiam wniosek o uchwalenie rzeczonego projektu ustawy w kształcie zaproponowanym przez komisję. Szanowni Państwo! Pomimo dokonania szeregu korekt, retuszy w pierwotnym projekcie główny rdzeń, kościec założeń wnioskodawców został utrzymany. Projekt przewiduje zaostrzenie konsekwencji i dodatkowe dolegliwości dla sprawców czynów korupcyjnych. Osoby skazane za przestępstwo korupcyjne enumeratywnie wyszczególnione w założeniach będą mogły zostać pozbawione praw publicznych, jak również będą orzekane w stosunku do nich środki karne w postaci zakazu wykonywania funkcji czy zawodów. W przypadku wystąpienia recydywy taki zakaz będzie orzekany dożywotnio. Szanowni państwo, tym samym będzie realizowana funkcja zarówno prewencyjna, jak i retrybutywna prawa karnego. Szanowni państwo, w pierwotnym założeniu te zapisy były troszeczkę bezzębne, mianowicie nie było penalizacji zachowań polegających na złamaniu tego zakazu, czyli zakazu wykonywania funkcji czy zawodów. Na skutek zmian będzie tutaj penalizacja, zostanie zmodyfikowany art. 244 Kodeksu karnego. Szanowni Państwo! Rozbudowany zostanie także zakaz możliwości piastowania funkcji przez posłów i senatorów, jak również parlamentarzystów. Można powiedzieć, że to będzie taki zakaz chałturzenia. Dodatkowo wprowadzone zostaną nowe przepisy odnośnie do zapewnienia większej przejrzystości i transparentności życia publicznego. Partie polityczne będą zmuszone przedstawiać źródła finansowania, jak również wydatki, które są czynione przez nie na poczet swoich działań. Trzeba podkreślić, że ci najbardziej hojni dobroczyńcy partyjni będą też musieli być uwidaczniani, wpłaty tutaj będą na poziomie 10 tys. zł. Dodatkowo przewiduje się, wyposaża Państwową Komisją Wyborczą w narzędzia do karania podmiotów w partii w sytuacji, w której nie będzie dokonywany ten obowiązek notyfikacji. Szanowni Państwo! Podsumowując, ten projekt ustawy to szansa na sanację sytuacji w obszarze, w którym będą dokonywane ingerencje legislacyjne. Trzeba podkreślić, że dodatkowo zwiększy to zabezpieczenie antykorupcyjne, jak również zwiększy przejrzystość życia publicznego.

Dziękuję bardzo. Witam państwa. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam honor przedstawić stanowisko naszego środowiska. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie popiera rzeczony projekt aktu normatywnego. Poseł sprawozdawca dość szeroko zrecenzował proponowane założenia i zmiany prawne, zatem nie ma potrzeby ich przytaczania i dublowania. Przedstawione argumenty nas przekonują. Projekt przewiduje nowy arsenał środków karnych, który powinien odstraszać potencjalnych sprawców. Ludzie władzy, którzy są sprzedajni, muszą się liczyć z tym, że będą rugowani, usuwani z życia publicznego. Dodatkowo zwiększa się przejrzystość życia publicznego poprzez, tak jak już wcześniej sygnalizowałem, konieczność ujawniania źródeł finansowania, jak również wydatków. Ogranicza się, szanowni państwo, do subminimum możliwość wykonywania pracy przez parlamentarzystów i samorządowców. Te przepisy będą wręcz skłaniały do przechodzenia na zawodowstwo. Tym samym osoby, które pełnią te funkcje, będą musiały skupić się, skoncentrować się na swojej działalności podstawowej. Szanowni Państwo! Prawo i Sprawiedliwość popiera zmiany i jest na tak. Chciałbym jednocześnie wnioskować, i złożyć poprawkę na podstawie art. 45, o rozszerzenie katalogu zadań Państwowej Komisji Wyborczej i zwiększenie roli opiniującej Państwowej Komisji Wyborczej przy wydawaniu rozporządzeń dotyczących określenia wzoru rejestru wpłat.

Taka kumulacja. Ciekawi jesteśmy, co w tej sprawie ma do powiedzenia poseł z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, pan poseł Tadeusz Zwiefka. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Każda zmiana legislacyjna, która ma na celu zaostrzenie przepisów w walce z korupcją, a także niegodnymi zachowaniami w życiu publicznym i zwiększenie transparentności tego życia publicznego, znajdzie poparcie w szeregach Koalicji Obywatelskiej.

Odnoszę wrażenie, że zatrzymaliśmy się gdzieś w połowie drogi. Mianowicie został zrobiony krok w prawidłowym kierunku, tylko że w połowie drogi zatrzymaliśmy się i nie chcemy zrobić kolejnego kroku, który doprowadziłby nas do finału. Czego one dotyczą? One dotyczą kilku kwestii.

Co powoduje, że nie jesteśmy do końca zadowoleni? Otóż projektodawcy przewidują, że ten przepis ma wejść w życie dopiero od przyszłej kadencji. My uważamy, że on powinien wejść w życie z momentem wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia przyszłego roku. Bo co?

Nie jest to ani moralne, ani uczciwe. Kolejna kwestia dotyczy transparentności życia publicznego.

Tylko ona potrzebuje, panie marszałku i Wysoka Izbo, odpowiedniego przepisu prawnego.

Pojawił się zarzut, że nie możemy tego uczynić, ponieważ taki wniosek został już złożony w przypadku ustawy z poprzedniej kadencji, a prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Otóż nie jest to wniosek tożsamy, proszę państwa, ponieważ tam chodziło także o dzieci. Trzecia kwestia dotyczy rozszerzenia zakresu niemożliwości łączenia funkcji, mandatu posła i senatora.

To jest moim zdaniem absolutnie niezbędne do tego, aby ta transparentność została w pełni zapewniona. Po raz kolejny zatem, panie marszałku, pozwolę sobie na pańskie ręce złożyć poprawki, które mam nadzieję, tym razem zostaną uwzględnione i naprawią ten projekt idący w dobrym kierunku, ale jak powiedziałem, niepełny, nieco tchórzliwy. Bądźmy bardziej odważni, bądźmy transparentni, tak jak oczekują tego nasi wyborcy. Mam nadzieję, że zostaną uwzględnione. Zapraszam panią posłankę Annę Marię Żukowską z klubu parlamentarnego Lewica. Bardzo proszę. Ustawa antykorupcyjna - jak to pięknie brzmi, prawie tak pięknie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, którego szefem jest Andrzej Stróżny, człowiek, który według komisji śledczej w sprawie śmierci Barbary Blidy powiedział nieprawdę, który już raz został pozbawiony certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. I tak jak powołanie tegoż CBA nie zlikwidowało w Polsce korupcji, tak uchwalenie tej ustawy też tego nie spowoduje. Do jej uchwalenia dochodzi nie z powodu jakichś wewnętrznych przekonań Prawa i Sprawiedliwości, bo chce tego partia, która, przypomnijmy, na własnym kongresie musiała przepychać uchwałę przeciwko nepotyzmowi. Tak, to o państwu, o panu, o pańskiej partii, panie Suski, mówię i o działaczach Prawa i Sprawiedliwości. A nepotyzm, tak jak kumoterstwo, to jest forma korupcji. Bowiem korupcją jest wszystko to, co jest wynikiem monopolu władzy partii rządzącej i uznaniowych decyzji, którym towarzyszy brak rozliczalności, a wy, panie i panowie z Prawa i Sprawiedliwości, właśnie dokładnie to robicie. Przed państwem mały przegląd afer korupcyjnych Prawa i Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości - Najwyższa Izba Kontroli po wyrywkowym sprawdzeniu zakwestionowała wydatki wynoszące w sumie 33 mln zł. Polska Fundacja Narodowa - fundacja zasłynęła kampanią „Sprawiedliwe sądy”, która miała wspierać zmiany w sądownictwie przeprowadzone przez partię rządzącą, bo była finansowana z pieniędzy spółek Skarbu Państwa. Sąd uznał, że kampania była niezgodna ze statutem fundacji. No i dalej: afera podkarpacka.

Z doniesień medialnych wiemy, że ówczesny szef CBA Ernest Bejda miał złożyć na ręce Mariusza Kamińskiego dymisję, która nie została jednak przyjęta.

Przepłacone przyłbice od żony tegoż instruktora narciarstwa. Ale to nie wszystko, bo odchodzący z rządu Jarosław Gowin ujawnił, że posłowie Porozumienia otrzymywali atrakcyjne oferty polityczne, byle zostali w klubie PiS. Zatem jesteście ekspertami nie tylko w zwykłych machlojach i przewalaniu pieniędzy, jesteście wybitnymi praktykami korupcji politycznej. Przeforsowanie na poprzednim posiedzeniu Sejmu lex TVN jest tego najświeższym i koronnym przykładem. W PiS-ie są wręcz konkretne korupcyjne cenniki.

Ma etat doradcy w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W tej naturze leży bezczelne, brutalne, niczym nieskrępowane rozpasanie. Wam już nawet nie jest ani odrobinę wstyd. Pani marszałek Witek, której akurat w tej chwili nie ma, wprawdzie z miną, jakby zjadła cytrynę, ale zarządziła reasumpcję głosowania, bo posłom Kukizowi i Sachajce, których też nie ma - a widzę pana posła Sachajkę - zajęło półtorej godziny dowiedzenie się, że się pomylili, bo wcześniej sami na to nie wpadli. Mentalność PiS-u jest jak woda, wejdzie w każdą szparę i po jakimś czasie spowoduje gnicie. Meandruje jak płytka, brudna rzeka, płynie, a na brzegach tworzy rozległe bagna. W tych bagnach klientelizmu siedzą po uszy działacze, rodziny, krewni, znajomi i kupieni przez PiS politycy. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Krzysztofa Paszyka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję. Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Zdaniem klubu Koalicji Polskiej wszelkie próby eliminowania z życia publicznego zjawisk korupcyjnych zasługują na poparcie. Takie poparcie ze strony klubu Koalicji Polskiej, naszych parlamentarzystów zarówno tu, w Sejmie, jak i w Senacie też będzie.

To nie służy dobrze temu, aby to było dobre prawo. Jeszcze gdyby to był targ polityczny w tle z argumentami, to pół biedy. Natomiast dobrze wiemy, że za nami kryzys w partii rządzącej związany z utratą większości na tej sali, i dlatego trwają prace nad tą ustawą.

Wsłuchałem się w to bardzo uważnie. Myślę, że państwo nie jesteście całkiem szczerzy wobec zarówno tej ustawy, jak i pomysłodawców tej ustawy. Bo gdybyście byli szczerzy i faktycznie chcieli eliminować wszelkie zjawiska patologiczne z życia publicznego, to ta ustawa wchodziłaby w życie niezwłocznie, a jej vacatio legis odsunięte do kolejnej kadencji parlamentu pokazuje nie całkiem szczerość, nie w pełni szczerość intencji.

Jeśli jesteście szczerzy w tym, co mówicie, to powinniście tę poprawkę poprzeć i powiedzieć: Tak, nie mamy nic do ukrycia, też zgadzamy się na to, aby eliminować korupcję z życia publicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Bardzo proszę pana posła Michała Gramatykę, Polska 2050. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Gdyby dzisiaj obowiązywały przepisy tej ustawy, pan poseł Lech Kołakowski nie mógłby np. pracować w państwowym banku, bo prawo nie zezwoliłoby mu na to. Nie wiadomo, co tam robi ani ile zarabia, wiadomo natomiast, że jest gwarantem utrzymania politycznej większości w Sejmie. Gdyby dziś to prawo obowiązywało, w radzie nadzorczej Kolei Śląskich nie mogliby zasiadać prezydenci Katowic i Opola. Uprzedzając pytania, tak, Koleje Śląskie to spółka rządzonego przez PiS województwa śląskiego, nie mają kapitałowo nic wspólnego z miastem Katowice, nie jeżdżą także do Opola. Jeżdżą za to do Kluczborka w województwie opolskim, ale tamtejszy burmistrz nie cieszy się względami pana premiera Morawieckiego. Jak Polska długa i szeroka takich przykładów są dziesiątki i zgodnie uznajemy je za patologiczne. Dlatego te rozwiązania są słuszne.

W odpowiedzi od pana posła Sachajki usłyszałem, że do końca trwającej kadencji panaceum na te patologiczne sytuacje mają być wyborcy. Jeżeli im się nie spodoba burmistrz, który sobie dorabia na boku, to go po prostu po raz kolejny nie wybiorą. Składamy więc te poprawki po raz kolejny. Jeżeli waszym celem jest walka z nepotyzmem, jeżeli waszym celem jest walka z korupcją, jeżeli ta ustawa naprawdę ma być antykorupcyjna, to każdy z was bez chwili wahania powinien za tymi poprawkami zagłosować.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia pragnę podziękować wszystkim członkom komisji, którzy zaangażowali się w pracę nad omawianym projektem, z jej przewodniczącym Piotrem Sakiem na czele. Dziękuję również Ministerstwu Sprawiedliwości z obecnym tutaj ministrem Marcinem Warchołem za dużo cennych uwag. Korupcja zwykle postrzegana jest jako działanie w sferze politycznej. Niestety niedoceniany jest jej zgubny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Wiedząc o zgubnym wpływie korupcji, proponujemy surowe rozwiązania, które będą pełniły funkcję prewencyjną i będą skutecznie zabezpieczały naszą ojczyznę przed niszczącym zjawiskiem korupcji. W projekcie zakłada się kilka fundamentalnych zmian. Po pierwsze, poszerzono katalog przestępstw, które będą skutkowały bardzo surowymi sankcjami, gdyż zmieniamy nie tylko Kodeks karny, ale również ustawę o sporcie i o refundacji leków. Dotkliwe sankcje, o których przed chwilą mówiłem, to obligatoryjna utrata pracy, a za dwukrotne skazanie za korupcję -dożywotni zakaz pracy w instytucjach publicznych. Instytucje publiczne powinny cieszyć się szczególnym zaufaniem. Po drugie, wprowadzono zakaz ubiegania się przez skazanych o zamówienia publiczne, czyli odcinamy ich od pieniędzy publicznych. Po trzecie, umożliwiamy sądowi pozbawienie skazanego za przestępstwa korupcyjne praw publicznych. W ten sposób wykluczamy możliwość ubiegania się o mandat wójta, burmistrza, prezydenta, posła i senatora. Po czwarte, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz posłowie i senatorowie nie będą mogli być zatrudniani w spółkach należących do Skarbu Państwa ani jednostek samorządowych. Po piąte, wprowadzamy większą transparentność w funkcjonowaniu partii politycznych poprzez obowiązek prowadzenia i aktualizacji rejestru wpłat, który będzie umieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej. Po szóste, partie polityczne będą miały obowiązek prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru zawieranych i zmienianych umów, które również będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Po siódme, wprowadza się transparentność w finansach publicznych samorządów poprzez obowiązek publikowania rejestru umów wraz z ich zmianami na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Wymienione rozwiązania zapobiegają tak szkodliwej korupcji i są to jedynie niektóre propozycje, jakie znajdują się w tej ustawie. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Oczywiście przepraszam za to, że nie dodałem części: demokracja bezpośrednia. Poprawię się. Bardzo proszę, pani poseł Agnieszka Ścigaj, Polskie Sprawy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projektodawcy! Panie Ministrze! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Koła Poselskiego Polskie Sprawy wobec projektowanej poselskiej ustawy o zmianie Kodeksu karnego i innych ustaw. Trochę jest tak, że czuję się nieswojo, stojąc tutaj i mówiąc o sprawach, które powinny być absolutnie oczywiste. Ktoś, kto był skazany za korupcję i wszystkie inne przestępstwa, które są z tym powiązane, nie był uczciwy, nie był przejrzysty, nie był transparentny. Po prostu tego nie powinno być w życiu publicznym.

Kilka moich uwag dotyczy natomiast tego, co mówił pan poseł sprawozdawca, że chcemy zmusić polskich parlamentarzystów m.in. do tego, żeby nie pracowali zawodowo, nie łączyli funkcji, tylko siedzieli i pracowali. Ja się z tym nie mogę zgodzić. Uważam, że nie ma w tym nic złego, że parlamentarzysta pracuje np. w ośrodku pomocy społecznej albo jest nauczycielem czy pielęgniarką w miejskim ośrodku zdrowia. Nic w tym złego nie ma. To miałoby rację bytu, kiedy byłaby zmiana ordynacji wyborczej i poseł musiałby pracować ze swoimi wyborcami, a nie tylko przy uchu swojego prezesa partii, bo tu się nie musi narobić, nic się nie narobi.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do zadawania pytań.

Bardzo proszę.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odkąd PiS objął władzę niestety poziom korupcji w Polsce stale rośnie. Ustawa mająca przeciwdziałać korupcji i nepotyzmowi jest oczywiście bezwzględnie potrzebna, ale z waszych ust brzmi to jak kpina, bo wy stale korupcję zwiększacie. Czym jeśli nie korupcją jest np. ułaskawienie skazanych za podżeganie do korupcji Kamińskiego i Wąsika? Każda wasza afera ma podłoże korupcyjne. Dwie wieże Kaczyńskiego, respiratory i maseczki Szumowskiego, wybory kopertowe Sasina, PCK Zalewskiej, pałace Obajtka - albo korupcyjne, albo złodziejskie. Mało tego, ta ustawa jest również owocem korupcji politycznej, której oddał się systemowy antysystemowiec. Dlatego chcę zapytać, jak zamierzacie dociągnąć do końca kadencji bez korumpowania posłów, bo z większością u was jest dosyć słabo.

Panie Ministrze!

Po pierwsze, przepisy dotyczące korupcji w stosunku do posłów i senatorów mają wejść w życie dopiero od kolejnej kadencji. Co to za przepisy antykorupcyjne, które będą obowiązywać za kilka lat? Tak naprawdę mówicie Polakom, że dzisiaj ci państwo mogą kraść bez opamiętania, a dopiero następna władza będzie podlegała tym przepisom. Przecież to hucpa. Kwoty poniżej 10 tys. zł nie będą ewidencjonowane w zakresie wpłat na partie polityczne. Jakie to są przepisy antykorupcyjne, które otwierają taką autostradę do tego, żeby ta korupcja kwitła? Dzisiejsza władza będzie z tego korzystała bez żadnych ograniczeń (Dzwonek), musicie to wiedzieć. Dzisiaj chodzi wyłącznie o to, żeby przy tej władzy trwać i niestety Kukiz’15 stał się częścią tego obozu władzy.

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Piotr Adamowicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Panie i Panowie Posłowie! Projekt ustawy przewiduje m.in. zakaz zawierania przez parlamentarzystów umów cywilnoprawnych z podmiotami, których Skarb Państwa posiada co najmniej 10%. Dlatego też chcę zapytać, czy projektodawcy zajmowali się taką oto sytuacją - i bez urazy panie pośle Pawle: jest mianowicie artysta, piosenkarz, lider zespołu, parlamentarzysta. Jego koncert jest organizowany przez prywatną agencję muzyczną, ale sponsoruje go np. Orlen pana Obajtka. Inna kwestia. Emisja spotów i utworów w tzw. mediach publicznych, czyli Skarb Państwa. Przez ZAIKS czy w innej formie - to jest inna zupełnie kwestia.

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Michał Szczerba, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Mam wrażenie, że mamy jakiś strasznie napompowany projekt, który ma być wielkim przełomem. Nie słyszałem głosu pana posła Kukiza, kiedy poseł Kołakowski był zatrudniany w Banku Gospodarstwa Krajowego. Za ile? Nie wiemy, panie pośle, ponieważ jak pytamy z posłem Jońskim, to bank odpowiada: To tajemnica bankowa. Poseł Mejza, poseł niezrzeszony głosujący z kołem reasumpcja, szanowni państwo, od kwietnia nie złożył oświadczenia majątkowego. Co dostał? Wypowiedział się pan w tej sprawie? Ja nie wiem. Kolejna sprawa. Czy kiedykolwiek, rozmawiając z prezydentem Dudą, zapytał się pan, co się dzieje z ustawą skierowaną do Trybunału Konstytucyjnego? Nic pan w tej sprawie nie zrobił. Trzy razy sprawdzam i trzy razy nawaliliście. Dziękuję serdecznie. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że pan poseł Mejza złożył oświadczenie majątkowe wczoraj albo przedwczoraj. Proszę bardzo, pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kolejny raz mamy do czynienia z projektem, który za pomocą jednego dokumentu nowelizuje szereg ustaw, począwszy od prawa do posiadania psa czy kota przez zasady określające zatrudnienie posłów oraz senatorów aż po kwestie związane z finansowaniem partii politycznych. Pytanie pierwsze. Dlaczego wprowadzono limit 10% udziału Skarbu Państwa w spółkach, w których nie może pracować poseł czy senator? W obecnym systemie przenikania form własności spółek limit ten powinien być ograniczony do zera. Kolejne pytanie. Jak rozumieć pojęcie stosunku pracy posłów i senatorów na rzecz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa? Pozostawia to olbrzymią furtkę pozwalającą na zarobkowanie w innej formie niż świadczenie pracy na rzecz omawianych spółek.

Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dlaczego? Jaki jest powód?

Czy możemy spodziewać się kolejnego projektu, który przesunie wejście w życie tych przepisów na kolejną kadencję? Mam nadzieję, że jak opozycja będzie rządziła, to tego nie zrobi.

Kilka przykładów z tej sali. Była już mowa o jednym z posłów, który za powrót do Zjednoczonej Prawicy otrzymał funkcję w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego pensja w momencie objęcia tej funkcji - nie wiem, czy on w ogóle w tym banku kiedykolwiek był - była pięciokrotnie wyższa od uposażenia poselskiego. Drugie pytanie. jest pytanie, czy on czasami nie księguje milionów zł z PiS-u lub spółek Skarbu Państwa w zamian za to, że głosuje z PiS-em ręka w rękę? Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Kiedy przyglądam się temu projektowi ustawy, mam wrażenie, że mógłbym zadać bardzo wiele pytań. Odpowiedź na każde z tych pytań udowodniłaby, jak dalece proponowane rozwiązania są niewystarczające. Ale zadam trzy. Jak chcecie państwo zapobiec korupcji, jeśli w Polsce oświadczenia majątkowego nie musi składać żona premiera, a np. dyrektor przedszkola musi? Jak chcecie zapobiec korupcji, jeśli na sali sejmowej zasiada parlamentarzysta, który bezkarnie odmawia składania oświadczenia majątkowego? I wreszcie jak chcecie zapobiec korupcji, jeśli na sali sejmowej zasiada parlamentarzysta, który najpierw odchodzi z klubu, potem do niego wraca, po czym otrzymuje lukratywną posadę, a potem zarabia, jak słyszałem, gdzieś ok. 40 tys. zł i będzie mógł to robić nadal przynajmniej przez 2 lata? Jak chcecie zlikwidować w Polsce korupcję, skoro akceptujecie takie rozwiązania? Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ale dlaczego nie obejmuje parlamentarzystów i parlamentarzystek obecnej kadencji? A może macie coś do ukrycia? Po tych wszystkich aferach i niejasnościach zaczynam mieć dużo co do tego wątpliwości, ale też zaczynam się bardzo mocno nad tym zastanawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Małgorzata Pępek, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Myślę, że wnioskodawca musi się zastanowić nad odpowiedzią na pytanie, dlaczego to wchodzi nie od zaraz, ale za 2 lata, gdyż już 12 osób zadało to pytanie. Słusznie. Wysoka Izbo! W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że wszystkie zmiany w ramach przepisów antykorupcyjnych powinny być szeroko omawiane z udziałem przedstawicieli administracji centralnej i samorządów. Tymczasem tak ważna ustawa procedowana jest jako projekt poselski, bez żadnych konsultacji, co już należy uznać za standard i złe praktyki legislacyjne. Ponadto wątpliwości budzi dyspozycja proponowanej normy prawnej. Formułuje się przepis ze słowami „sąd może” i nie wskazuje się przy tym dodatkowych dyrektyw, jakimi powinien się sąd kierować, orzekając taki środek karny. Brak takich przesłanek spowoduje, że w skali kraju sądy wytworzą niejednolite praktyki orzecznicze na tym gruncie. Czy wobec powyższego (Dzwonek) nie zachodzi ryzyko orzekania środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych tylko na podstawie uznania sądu? Dlaczego ustawa wchodzi w życie w następnej kadencji? Dziękuję serdecznie. Pan poseł Grzegorz Lorek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Ustawa jest bardzo ważna. Wreszcie mamy krok milowy - możemy walczyć z korupcją. Wreszcie to nastąpiło. Przez 30 lat nie mogło się to wydarzyć. Mamy wreszcie tę ustawę. Ja bym powiedział więcej: kto nie zagłosuje za tą ustawą, to jest za korupcją, to znaczy, że taki model państwa mu się podoba. I w tym zakresie ta ustawa ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli macie państwo uwagi, to zajmijmy się sprawami merytorycznymi. Tak, zadaliście 13 razy to pytanie, pewnie jeszcze wiele razy je zadacie. Ale zacznijcie myśleć nad konsekwencjami tych przepisów, bo o tym w ogóle nie chcecie mówić. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! W końcu mamy ustawę, która wprost odpowiada na zapotrzebowanie społeczne, ogranicza korupcję wśród polityków i osób sprawujących władzę. Chcę podziękować panu posłowi Zwiefce, pani poseł marszałek Dolniak, bo w podkomisji pracowaliście państwo merytorycznie nad tą ustawą. A więc tutaj ta sprawa nie powinna nas różnić. Natomiast mam apel do pana Michała Szczerby, który tutaj tak grzmi i używa wielkich słów o walce z korupcją. Proszę zachęcić swojego kolegę partyjnego pana marszałka Tomasza Grodzkiego, aby poddał w końcu wniosek o uchylenie immunitetu pod głosowanie. Chcecie walczyć z korupcją, to niech pan marszałek Grodzki podda się ocenie sądu, bo wpłynął akt oskarżenia związany z prawdopodobieństwem, oskarżeniami wielu osób. o przyjmowanie korzyści majątkowych. To jest naprawdę pierwszy poważny krok, aby poważnie walczyć z korupcją, i jestem przekonany (Dzwonek), że będziemy tę ustawę jeszcze nowelizować i zaostrzać. Dziękuję serdecznie. Rzadko to robię, ale powiem, że jest wiele uroku w tym, jak parlamentarzyści PiS-u dziękują panu Kukizowi za to, że wreszcie wprowadził ustawę antykorupcyjną.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To, co powiedział pan marszałek - paradoks. Ale gratuluję. Jestem jak najbardziej za. Transparentność - jak najbardziej za. Ale nie dotyczy to obecnej władzy, nie dotyczy to obecnych posłów, senatorów. Dlaczego? Dlatego że gdyby dotyczyło, to po pierwsze, PiS by stracił większość parlamentarną, a ci państwo, panowie straciliby swoje intratne posady. Moje pytanie brzmi: Dlaczego to ma nie dotyczyć tej władzy, tylko ma być dopiero od nowej kadencji?

Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Joński, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Celem tego projektu ustawy jest walka z nepotyzmem i korupcją.

Nic. Co więcej, teraz się pojawia projekt ustawy, który ma działać za 2 lata. Dzisiaj model państwa jest taki, że dokładnie działa bezkarność.

Wszystkie te sprawy są umarzane, bo obowiązuje ustawa o bezkarności, a wy mówicie o tym, że wprowadzimy ustawę, która będzie walczyła z korupcją i nepotyzmem. I na koniec chcę powiedzieć taką jedną rzecz. Otóż wydaje się, że jest odpowiedź, dlaczego ta ustawa ma działać dopiero za 2 lata. Właśnie dlatego, żeby te wszystkie afery związane oczywiście z zakupami, z Ostrołęką, z handlarzem bronią zostały umorzone, żeby to wszystko zostało umorzone. Dopiero za 2 lata mamy walczyć z korupcją. Na tym polega ten projekt. Dziękuję serdecznie. Proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przyjmuję, że każdy, kto tutaj zasiada, chciałby działać uczciwie i przejrzyście. Nikomu nie odbieram prawa do tego i nikogo nie krytykuję za to, że jego intencje są inne.

To też jest oczekiwanie społeczne, bo każdy, kto jest wybrany przez społeczeństwo, oczekuje, żeby taka była władza. Bardzo się cieszę, bo udział parlamentarzystów, wójtów, burmistrzów i prezydentów w spółkach Skarbu Państwa czy samorządowych powinien być ograniczony.

Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Wysoka Izbo! W projektowanych przez was przepisach pojawia się środek karny, który polega na tym, że osoba skazana za przestępstwo musi być przez sąd ukarana również zakazem zajmowania stanowisk, wykonywania pracy, świadczenia usług na rzecz organów i instytucji publicznych. Mam pytanie o to „musi” Dlaczego ten środek karny jest obligatoryjny? Czy to nie ogranicza swobody podejmowania decyzji przez sąd? Czy to nie ogranicza niezawisłości sędziowskiej wyrażonej w art. 8 Kodeksu postępowania karnego? Jeszcze jedno pytanie: Dlaczego ten środek karny spośród katalogu przestępstw zakwalifikowanych do stosowania tego środka karnego wyleciał na jednym z etapów prac? Przecież to jest ten artykuł, w przypadku którego będą odpowiadać np. architekci kopertowych wyborów, o których dzisiaj rozmawialiśmy (Dzwonek) nieco wcześniej. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Dlaczego, panie pośle, w ustawie nie znalazło się miejsce poświęcone takim funduszom jak Polska Fundacja Narodowa czy Fundusz Sprawiedliwości, które w czystej postaci są wykorzystywane do tego, aby nagradzać różne środowiska?

Bo tu są rozwiązania, które pozwolą omijać waszą ustawę.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Wysoka Izbo! To ustawa antykorupcyjna, nawet jeżeli jest niedoskonała, nawet jeżeli czegoś jej brakuje, nawet jeżeli można ją poprawić. Dlaczego tak państwo z niej szydzicie? Dlaczego nie chcecie jej zaakceptować? Przecież w sytuacji, w której dziecko uczy się chodzić, w której dziecko uczy się jeździć na rowerku, nie mówicie: nie, daj sobie spokój, lepiej żebyś przez całe życie pełzał. Kiedy uczy się jeździć na rowerku, najpierw ma kółeczka. Po co? Żeby nauczyć się trzymać równowagę. Ustawa antykorupcyjna jest pierwszym etapem. Będą na pewno kolejne. Dajcie tej ustawie szansę. To jest niesamowita sytuacja, w której ta ustawa może być przyjęta przez wszystkie środowiska polityczne. Byliście państwo u władzy wielokrotnie. Nie zrobiliście nic. Szacunek, Paweł. Dziękuję serdecznie. Panie pośle, zostało zgłoszonych 12 poprawek przez cztery kluby. Więc myślę, że ma pan złą ocenę, bo po prostu kluby składają poprawki. Zobaczymy, co z nimi będzie.

Ale umówmy się, że nie wypuszczę pana z Sejmu. Dobrze, ale to mam tutaj.

Odpowie pan czy nie? Jak pan myśli? Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za wywołanie. Nie zmienia się reguł gry w jej trakcie.

W tej chwili konstytucję odkładacie na bok, jakieś inne porządki prawne są dla was ważniejsze niż nasza polska konstytucja. Właśnie tam jest mowa o prawach nabytych i dlatego w imię ochrony praw nabytych propozycja ta powinna być realizowana od przyszłej kadencji. W odniesieniu do pozostałych pytań, które tutaj padły, jeśli chodzi o możliwość fakultatywnego pozbawienia praw publicznych czy obligatoryjne orzekanie przez sąd zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, to nie może pełnić funkcji publicznych ten, kto w jakikolwiek sposób został uwikłany w działania korupcyjne. Tak więc te rozwiązania są nowatorskie w naszym systemie prawnym.

Dziękuję serdecznie. O głos prosił sprawozdawca komisji pan poseł Piotr Sak. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny, ale i Złośliwy Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć na państwa pytania w zależności od posiadanej wiedzy, ewentualnie improwizować. Bardzo dziękuję za wszelkie pytania, chociaż patrząc na niektóre z nich, odniosłem takie wrażenie, że te pytania i wystąpienia pomyliły się niektórym posłom czy posłankom z konkursem na jakąś najbardziej dramatyczną rolę damską czy męską. Odnosząc się do pytania posła Miszalskiego. Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Suchonia, to oczywiście nie ma idealnego panaceum, remedium, nie ma wunderwaffe na ludzkie żądze, niemniej jednak wydaje się, że ten projekt ma charakter ewidentnie odstraszający, prewencyjny, a jeżeli już dojdzie do czynu zabronionego, to będzie za to sroga odpłata ze strony państwa. Wydaje mi się, że w tym zakresie jest to klarowne.

Niezależnie od możliwości podejmowania różnych prac przez posłów, parlamentarzystów, senatorów czy samorządowców wykonywanie mandatu może mieć charakter, można powiedzieć, zawodowy i społeczny. Odnośnie do pytania pana posła Szczerby myślę, że pana ciekawość, panie pośle, zostanie niebawem zaspokojona.

Chciałbym zauważyć, że jednak dokumentujemy w oświadczeniach majątkowych stan na koniec roku, więc zakładam, że ta pana ciekawość zostanie zaspokojona pewno koło maja 2022 r. Tylko cierpliwi zwyciężają. Spokojnie.

Było tu już to przedstawiane. Mamy świadomość, że jest ustawa o jawności życia publicznego.

Mogłoby to rodzić takie konsekwencje, że ta ustawa mogłaby także zostać skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.

Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Jońskiego i generalnie wydobywając te wszystkie akcenty. Dzisiaj macie pretensje o to, że cokolwiek w tym temacie drgnęło. Rozumiem, że można kontestować, można być malkontentem, ale naprawdę pokażcie, co wy robiliście w tym obszarze. Kalibruję wzrok na tę stronę, więc myślę, że pan poseł się domyśli. Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi jeszcze o pytanie pana posła Gramatyki odnośnie do art. 231 § 2.

Oczywiście może być skutek w postaci jakiejś szkody dla interesu publicznego czy osobistego. Niemniej jednak uznaliśmy, że nie ma to.

Niedużo trzeba, bo to jest zawsze duże ryzyko.

Mam nadzieję, że te wyjaśnienia, które państwu przedstawiłem, będą satysfakcjonujące. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie pośle, mam jeszcze prośbę, jakby był pan tak uprzejmy. Chciałbym zauważyć, panie marszałku, że jednak pan nie zadał pytania z mównicy, a myślę, że najlepszym argumentem były argumenty pana ministra Warchoła. Proszę pana, chciałem panu powiedzieć, że ja jestem wicemarszałkiem Sejmu, który zadał panu pytanie z mównicy, bo to jest moja mównica. Więc jeżeli byłby pan tak uprzejmy i spróbował na to odpowiedzieć, to byłbym wdzięczny. Jeżeli nie, też będę wdzięczny, bo przecież pana szanuję.

Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku! Jarosław Sachajko. Chciałem wszystkim podziękować, wszystkim, którzy pracowali nad tą ustawą, za to, że jednak udało się tę ustawę przyjąć w dobrym kształcie. Przepraszam, nie pamiętam nazwiska pana posła z Lewicy, który jako pierwszy zadawał pytanie. Mówił on o stosunku pracy. W ogóle obawiam się, że wielu posłów nie przeczytało tej ustawy, bo tutaj nie ma mowy o stosunku pracy. Czyli tu mamy pełny wachlarz pracy.

Ja tylko przypomnę, że mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. To właśnie posłowie są tą ustawodawczą, to posłowie powinni pracować, a rząd jest władzą wykonawczą. Czyli rząd powinien wykonywać to, co posłowie przygotowują. Przygotowujcie projekty ustaw i składajcie je. Sprawdziłem, pani jest posłanką trzecią kadencję, więc miała pani okazję w swojej kadencji, w pierwszej swojej kadencji również złożyć taką bardzo ważną ustawę. Mówiła pani również, dlaczego tu jest: sąd może. Jakby pani przeczytała to o zakazie pracy, mamy obligatoryjność.

Znowu była mowa o tym, że ustawa wchodzi w życie od kolejnej kadencji. Za chwilę ona wejdzie w życie, więc nie od następnej kadencji. Są dwa przepisy, które dopiero wchodzą od następnej kadencji, ale to pan minister dosyć klarownie wyjaśnił, dlaczego od następnej kadencji.

Pan poseł Dariusz Joński mówił o tym, że będzie bezkarność tej kadencji.

Wchodzi to od tej kadencji.

Można było to dołożyć.

Dlatego jest to bardzo ważne, żeby sąd musiał w tej chwili wydać zakaz pracy.

Dziękuję bardzo, myślę. Jeszcze było pytanie pana posła Paszyka, dlaczego nie zajmujemy się finansowaniem kampanii wyborczej. Dokładnie to samo pytanie mogę panu zadać, dlaczego pan nie przyszedł i nie zwrócił uwagi na to, żeby włączyć tę kwestię do prac komisji. Dziękuję serdecznie.

Dziękuję serdecznie panu posłowi. W trybie? Nikt pani nie atakował, wydaje mi się. Proszę bardzo. 30 sekund. Wysoka Izbo! Niech pan nie ucieka, bo to, co pan mówi, nie zgadza się, nie pokrywa się to z prawdą, bo klub Koalicji Obywatelskiej złożył projekt ustawy o zniesieniu bezkarności urzędników już w lipcu 2020 r., czyli już ponad rok temu, i nie odbyło się nawet pierwsze czytanie.

No dobrze, ale wie pani, to jest Sejm, pani posłanko. Proszę bardzo, panie pośle, w trybie sprostowania - 30 sekund i kończymy. Pani Poseł!

Powiedziałem, że pani jest posłanką trzecią kadencję i zwróciłem pani uwagę, że pani jako posłanka mogła złożyć podobną ustawę już wiele, wiele lat temu, a pani tego nie zrobiła i oskarża mnie pani o kłamstwo. Wstyd. No dobrze. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, na podstawie art. 95 ust. 2 regulaminu Sejmu kieruję ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu przedstawienia sprawozdania. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1399 i 1480) Proszę pana posła Jerzego Bieleckiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Projekt wprowadza zmiany głównie w trzech ustawach regulujących tzw. sprawy obywatelskie, w ramach których określono wprowadzenie odpowiednio rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych oraz Rejestru Stanu Cywilnego. Nie ma marszałka?

Projekt zakłada przyjęcie podstaw prawnych do stosowania usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu obywatela. Usługi te przyczynią się do przyspieszenia załatwienia spraw, zmniejszą obciążenie urzędników obowiązkami, przyspieszą czas realizacji usług, jak też zredukują ilość dokumentów dostarczanych i gromadzonych w formie papierowej. Pozwolą obywatelom zaoszczędzić na opłatach skarbowych. Usługi zostaną zaimplementowane w witrynie gov.pl, stanowiącej podstawowe źródło wiedzy dla obywateli w zakresie załatwianych konkretnych spraw urzędowych przy użyciu profilu zaufanego lub profilu osobistego. Proponowane zmiany zawierają pakiet usług elektronicznych w obszarze spraw obywatelskich, których wspólnym mianownikiem jest transakcyjność i zautomatyzowanie procesów i usług dla obywateli z wykorzystaniem rejestrów wprowadzonych przez ministra cyfryzacji oraz wykorzystaniem pieczęci elektronicznej. Ze wspomnianych rejestrów obywatele będą mogli pobierać dokumenty zawierające informacje o podmiotach, którym udostępniono ich dane osobowe. W zakresie ustawy o dowodach osobistych wnioskodawcom zostanie zapewniona możliwość udostępnienia własnych danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych oraz przedkładania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających sprawdzenie przesłanek ustawowych do przyznania dostępu.

Przy elektronicznym zgłaszaniu urodzenia dziecka zostanie zapewniona możliwość otrzymania odpisu skróconego aktu urodzenia, zaświadczenia o zameldowaniu dziecka oraz powiadomienia o nadaniu nr PESEL.

Zaświadczenia pobierane z rejestru w formie elektronicznej będą opatrywane pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji i weryfikowane przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu wraz z 13 poprawkami o charakterze legislacyjnym wnosi o uchwalenie przez Wysoki Sejm przedstawionego projektu ustawy.

Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam ogromny zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nie ulega wątpliwości fakt, że jako społeczeństwo zyskujemy coraz to nowe narzędzia znajdujące się w wachlarzu szeroko pojętego rozwoju cyfrowego. Rzeczą pożądaną jest, aby w miarę możliwości i biorąc pod uwagę swoje uwarunkowania, administracja publiczna sięgała po wspomniane narzędzia i stała się dzięki temu dostępniejsza dla ludzi. Procedowany projekt ustawy ma na celu umożliwić obywatelom załatwienie podstawowych spraw urzędowych w formie zdalnej za pomocą prostych, intuicyjnych i dedykowanych konkretnym czynnościom usług elektronicznych. Jak zapewnia rząd, będzie szybciej i wygodniej, a także możliwie prościej, z myślą o osobach, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w Internecie. Istotne są też również w kontekście procedowanej ustawy doświadczenia, które administracja państwowa nabywa podczas pandemii COVID-19, gdy zdecydowanie zwiększyła się skala wydawanych zdalnie dokumentów. Najprościej rzecz ujmując, wśród najważniejszych korzyści proponowanych rozwiązań możemy wymienić ułatwienie załatwiania spraw urzędowych obywatelom, przyspieszenie i ułatwienie realizacji spraw przez urzędy oraz obniżenie kosztów finansowania niektórych zadań zleconych z obszaru spraw obywatelskich. Natomiast samymi przykładami proponowanych rozwiązań są m.in. usługa pobrania z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących osoby oraz jej dzieci przy użyciu transakcyjnej usługi elektronicznej, usługa umożliwiająca pobranie informacji o odbiorcach danych z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL, możliwość opatrywania pieczęcią ministra odpisów aktu urodzenia wydawanych z urzędu na skutek elektronicznego zgłoszenia urodzenia dziecka, usługa pobrania zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym, o danych przetwarzanych w rejestrze stanu cywilnego opatrywanych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, zapewnienie możliwości wnioskowania o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz rejestru PESEL w trybie ograniczonej teletransmisji danych przy użyciu dedykowanej usługi oraz przedkładania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek ustawowych do przyznania dostępu, usługa transakcyjnego zameldowania się w lokalu i wymeldowania się z lokalu, realizowana w systemie bez udziału urzędnika, zgłoszenie wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu oraz powrotu. Zaproponowane zmiany są zatem pakietem usług elektronicznych w zakresie spraw obywatelskich, których wspólną cechą jest transakcyjność, zautomatyzowanie procesów i usług przy wykorzystaniu rejestrów państwowych i pieczęci elektronicznej. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym również zgłosić poprawkę do procedowanej ustawy polegającą na zastąpieniu w art. 7 w pkt 1 wyrazów „art. 1 pkt 4” wyrazami „art. 1 pkt 5”

Tym samym zakładana zmiana ma na celu skorelowanie terminu wejścia w życie ustawy z terminem, w którym faktycznie zostanie uruchomiona usługa. Podkreślenia wymaga również to, że takie było pierwotne założenie projektodawcy, a do niespójności przepisów w tym zakresie doszło wskutek dokonywania zmian w toku procesu legislacyjnego przedmiotowej ustawy. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że zakładana poprawka zapewni sądom podstawy prawne do korzystania z pełnej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów Osobistych wraz z wejściem w życie ustawy. Przepis ten nie obliguje sądów do korzystania z tego trybu od dnia wejścia w życie przepisów, a jedynie im daje im taką możliwość. Stworzenie podstaw prawnych umożliwi natomiast wystąpienie przez ministra sprawiedliwości z wnioskiem o zapewnienie im takiego dostępu. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Informuję, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierał rządowy projekt (Dzwonek) ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw w dalszych pracach legislacyjnych. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Grzegorza Napieralskiego, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska chciałbym zaopiniować projekt ustawy. Projekt wprowadza zmiany w trzech ustawach regulujących funkcjonowanie rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych oraz rejestru stanu cywilnego. Proponowane zmiany dotyczą głównie możliwości wprowadzenia transakcyjności, zautomatyzowania procesów i usług dla obywateli świadczonych na podstawie rejestrów administrowanych przez ministra cyfryzacji oraz wykorzystania pieczęci elektronicznej. Wśród istniejących usług publicznych, które mają zostać udostępnione w wersji cyfrowej i transakcyjnej, są m.in. zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego, zaświadczenia z rejestru PESEL czy usługa zameldowania. Ponadto ta ustawa implementuje także nową usługę, która pozwala obywatelowi dowiedzieć się, jakie podmioty występowały o dane jego dotyczące z takich rejestrów jak rejestr PESEL. Konieczność tej implementacji wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. I co najważniejsze, szanowni państwo, nowe udostępnione usługi będą nieodpłatne dla obywateli. Dotychczas otrzymanie zaświadczenia w urzędzie wiązało się z opłatą w wysokości kilkudziesięciu złotych, teraz będzie to za darmo. Transakcyjność usługi oznacza, że dzieje się ona automatycznie na podstawie wniosku i baz danych, tj. rejestrów publicznych, ponadto nie wymaga udziału urzędnika, tak jak np. zrobienie przelewu przez stronę internetową banku nie wymaga udziału pracownika banku. Jest to ważny trend w udostępnianiu usług publicznych, pozwalający skrócić czas oczekiwania na załatwienie sprawy - w większości przypadków możliwe będzie otrzymanie zaświadczenia, nazwijmy to: od ręki - a także obniżyć koszty funkcjonowania administracji. Zgłoszone podczas pierwszego czytania poprawki miały legislacyjny i techniczny charakter i zostały jednogłośnie przyjęte przez komisje. Natomiast, panie ministrze, chciałbym dzisiaj w tym wystąpieniu zwrócić uwagę na trzy aspekty związane z tym projektem.

Poziom tego ryzyka będzie zależny od konkretnego sposobu implementacji usługi w systemie teleinformatycznym.

Natomiast ustawa idzie w bardzo dobrym kierunku. Dziękuję, panie marszałku. Pan poseł Robert Kwiatkowski, klub parlamentarny Lewica. Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jedyne uwagi, które pojawiły się w trakcie posiedzenia tej komisji, to uwagi o charakterze legislacyjnym bądź technicznym - bo też w istocie projekt tej ustawy ma taki właśnie techniczny charakter. Język podobnie jak materia są dość skomplikowane, a przecież chodzi o sprawy proste i ważne z punktu widzenia przeciętnego obywatela.

A więc można zakładać, że ta nowelizacja jest ważna, jest potrzebna i dotykać będzie spraw ważnych i istotnych dla być może milionów ludzi. Na pewno w ciągu wielu lat funkcjonowania bez zmian, na co, panie ministrze, mam nadzieję, ta ustawa dotykać będzie spraw urzędowych i mniej urzędowych milionów Polaków. Klub parlamentarny Lewica, który mam zaszczyt reprezentować, odnosząc się do tego przedłożenia rządowego, będzie popierał, tak jak uczyniliśmy to w trakcie posiedzenia komisji, to przedłożenie i projekt dyskutowanej ustawy. Pozwolę sobie jednak, podobnie jak poprzednik, sformułować dwie uwagi pod adresem pana ministra. Jedna wynika bezpośrednio z wystąpienia przedstawiciela klubu parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy.

Dlaczego to jest istotne? Dlatego że, jak mi się wydaje, potrzebna by tu była porządna kampania informacyjna, w ramach której innymi słowami niż te, z którymi się można zapoznać w uzasadnieniu tego projektu, tłumaczono i opisywano by istotę proponowanych zmian i poprawek, bo przepisy tej ustawy, a raczej nowe funkcjonalności, które się nią wprowadza w relacjach organ administracji państwowej - obywatel, pozostaną martwe dla bardzo wielu ludzi, jeśli ci ludzie, obywatele nie będą świadomi tego, że takie udogodnienia i takie ułatwienia, a one są poważne, są prawdziwe, już weszły w życie.

Bardzo dziękuję. Pan poseł Dariusz Kurzawa, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Zapraszam, panie pośle. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić uwagi mojego klubu, klubu Koalicja Polska, odnośnie do nowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1399 i 1480. Proponowane zmiany należą do tzw. spraw obywatelskich i obejmują pakiet usług elektronicznych, które mają na celu transakcyjność i automatyzację procesów oraz usług dla obywateli z wykorzystaniem rejestrów administrowanych przez ministra cyfryzacji oraz wykorzystanie pieczęci elektronicznej. Zmiany we wspomnianych ustawach spowodują ułatwienia związane z dostępem do dokumentacji. Chodzi o meldunek, bazę PESEL, informacje o pobieranych danych o dziecku, korzystanie z danych zawartych w księdze wieczystej czy też informacje o hipotece.

Ale lepiej późno niż wcale. Pojawiły się także tutaj podczas wystąpień przedstawicieli innych klubów sprawy związane choćby z dochodami gmin, bo rzeczywiście, jak spojrzymy na ilość składanych wniosków, także opłaty z tym związane, to idzie to w setki tysięcy wniosków, a co za tym też idzie - pieniądze i dochody małych gmin, np. takich jak Jeziora Wielkie, z których ja pochodzę, gdzie jest niespełna 5 tys. mieszkańców.

Jest też pytanie o zasadność takiego wyłączenia. Mam nadzieję, że pan minister rozwieje także te nasze wątpliwości. Chciałbym przedstawić stanowisko w imieniu klubu Koalicja Polska. Jest ono jak najbardziej pozytywne. Musimy iść do przodu i wprowadzać takie zmiany w administracji, które będą ułatwiały życie wszystkim Polakom. Wobec tego mój klub będzie głosował za proponowanymi zmianami, za wprowadzeniem tych zmian do ustawy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Krystian Kamiński, koło Konfederacja.

Wysoka Izbo! Sama informatyzacja poszczególnych urzędów jest niekontrowersyjna. Jednak w uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, że skutki ustawy obejmą obok polskich obywateli również 430 tys. cudzoziemców. Udostępnienie składania dokumentów przez Internet przez obcokrajowców to bardzo daleko idące udogodnienie. Powstaje pytanie, jak w związku z tym realnie weryfikować te osoby. Dlaczego rząd podejmuje takie działania? Otóż ten rząd realizuje politykę masowej imigracji, która skończy się budową społeczeństwa multikulturowego, jak na Zachodzie. Przypomnijmy, że w styczniu br. na stałe w Polsce mieszkało 2106 tys. obcokrajowców.

Kolejne dziesiątki tysięcy wniosków, jeśli nie setki tysięcy, czekają na rozpoznanie. Rząd PiS to nieustanny wzrost masowej imigracji, w szczególności z Ukrainy. Dziennik Gazeta Prawna” donosi o kolejnym projekcie mającym przyspieszyć procedurę wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy. Nie wystarczy wam ulga dla imigranta. Nie wystarczy wam emerytura dla Ukraińca. Co następne? Obywatelstwo przez Internet? Bo w tym kierunku to niestety idzie. Co to w ogóle za kryterium, że chociażby tzw. ulga na powrót ma przysługiwać komuś, kto mieszkał przez 3 lata na terenie Unii Europejskiej albo USA, albo Wielkiej Brytanii, albo Meksyku, Chile, Izraela, Nowej Zelandii, Japonii lub Kanady? Jaki powrót? Czemu zwolnienie przez 4 lata z 50-procentowego podatku PIT ma dostać Nigeryjczyk, który studiował na terenie Unii Europejskiej, albo Filipińczyk mieszkający kilka lat temu w Japonii? Konfederacja apelowała już o wykorzystanie procedury, o której mowa w art. 90b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i wyznaczenie limitu maksymalnej liczby zezwoleń na pracę. W tej chwili żądamy moratorium migracyjnego do czasu przedstawienia wiarygodnej polityki kontrolowanej imigracji przez rząd, a nie kolejnych udogodnień dla cudzoziemców. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Panie Ministrze! To jest dobre prawo. Ta ustawa automatyzuje proces przekazywania danych w kolejnych obszarach, eliminuje w nich udział człowieka, i to jest bardzo dobre. Ustawa rozpowszechnia użycie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, i to także jest godne zauważenia, podkreślenia i pochwały. Pobocznym skutkiem ustawy będzie, o czym wspominał pan poseł Napieralski, pozbawienie niektórych urzędów miast i gmin dochodów z tytułu opłat skarbowych pobieranych za tradycyjne nieelektroniczne przekazanie tego typu danych. To będzie znaczące szczególnie w przypadku mniejszych urzędów. Oto organ, który nie ma wystarczającego zaufania do przedłożonych dokumentów elektronicznych, może zażądać ich przedłożenia na piśmie. Nie za bardzo wiadomo, po co. Wszak przynajmniej od czasów bulli „Pietati proximum” papieża Grzegorza IX wiadomo, że dokument tradycyjny jest znacznie łatwiejszy do sfałszowania niż dokument elektroniczny. Ten przepis pojawia się też w dalszej części druku w odniesieniu do kolejnych sytuacji. W naszej ocenie jest on po prostu zbędny. Ale Polska 2050 jest organizacją, która patrzy w przyszłość w dalekim horyzoncie, i każda forma cyfryzacji życia publicznego może liczyć na nasze poparcie. Nie wiem, czy pan wie, ale jednym z ostatnich bastionów, które honorują wyłącznie analogowe dokumenty, jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj obywatel, który prezentuje elektroniczny dowód osobisty, nie ma kompletnie szans w starciu z dzielną Strażą Marszałkowską, bo ona po prostu takich dokumentów nie honoruje, a nie honoruje, bo nie może. Zarządzenie marszałek Sejmu w tej sprawie ma już 13 lat. Proszę mi wierzyć, że bardzo się zmienił, szczególnie w dziedzinie cyfryzacji. Obywatel nie może wysłać do Kancelarii Sejmu pisma elektronicznego. To znaczy: może je wysłać, ale nie dostanie elektronicznej odpowiedzi, a czasem się zdarza, że w ogóle nie dostanie odpowiedzi. To jest naprawdę dobry moment, żeby również Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wykonał kilka kroków w chmurach na drodze do powszechnej cyfryzacji. Dziękuję serdecznie, czcigodny panie pośle. W trybie natychmiastowym przekażę pana uwagi pani marszałek Witek. Na pewno wdroży to w trybie pilnym. Proszę państwa, sześć pytań będzie zadawanych. Pan poseł Grzegorz Lorek z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zada pytanie pierwsze. Proszę bardzo. Minuta na zadawanie pytań. Nie ma pana posła. Pani poseł Małgorzata Pępek, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Mam dzisiaj szczęście do pani, pani poseł. Będę tu częściej przychodził. Wysoka Izbo! Cyfryzacja w administracji ma pomagać obywatelom i upraszczać proces uzyskiwania dokumentów. Jeszcze do niedawna osoby chcące wyrobić dowód osobisty mogły to zrobić elektronicznie, gdy miały profil zaufany.

Tym samym istnieje ogromna baza danych biometrycznych obywateli.

Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Spóźniony pan poseł Grzegorz Lorek zabierze głos. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

O co mi chodzi?

Dziękuję. Pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Na temat kolejnych nowelizacji związanych ze sprawami dowodów osobistych oraz ewidencją ludności można w ostatnich latach napisać książkę.

Czy przepis pozwala na uznaniowe wpisywanie takich informacji do rejestru przez urząd? Jeżeli nie i rejestr ten jest uporządkowany i jednoznaczny, to dlaczego rodzic jest zobowiązany do składania oświadczenia, że dziecko znajduje się pod jego opieką? Jeżeli urząd prowadzi usystematyzowany rejestr i warunkiem udzielenia informacji jest wypełniona rubryka w tym rejestrze, to dlaczego projektodawca (Dzwonek) wymaga dodatkowych oświadczeń?

Panie Ministrze!

W szczególnych przypadkach może to posłużyć, powiedziałbym, celom zupełnie sprzecznym z tymi, które przyświecają tej ustawie.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Artur Łącki, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze!

Stawiam pytanie, jak państwo chcecie zrekompensować i czy w ogóle chcecie zrekompensować - ja bym był za tym, żebyście zrekompensowali - te przychody gmin.

Dziękuję serdecznie. Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego to pakiet usług elektronicznych dla ludności jak najbardziej właściwy, pożądany i oczekiwany. Jednak te wszystkie usługi spoczywają na samorządach. Moje pytanie do pana ministra: Czy przewidzieliście państwo rekompensatę kosztów, które poniosą samorządy na skutek utrzymania, obsługi systemu? Ale ta ustawa to także uszczerbek w dochodach samorządów. Moje pytanie: Czy przewidzieliście zwrot czy rekompensatę utraconych kosztów?

Dziękuję serdecznie. Zapraszam sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa pana ministra Janusza Cieszyńskiego. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za te pytania. W szczególności chcę podziękować nawet nie tyle za pytania, co za pozytywne nastawienie i wręcz entuzjazm dla tego projektu, nie zawsze spotykany przy przedłożeniach rządowych. Dobrze.

Otóż, szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę na to, że istotą tego projektu jest zamiana e-usług, które funkcjonują dzisiaj, polegających na tym, że składamy coś na formularzu rządowym, trafia to do samorządu i na tej podstawie samorząd generuje jakiś dokument, na usługę o charakterze - pan poseł Kwiatkowski do tego się odnosił - transakcyjnym. Co to oznacza?

Tak, to są pieniądze, które już zostały nam przyznane.

A myślę, że patrząc na kwestie związane z bezpieczeństwem, powinniśmy przede wszystkim patrzeć, czy wprowadzenie mechanizmu zdalnego czy cyfrowego w jakiś istotny sposób zmienia poziom bezpieczeństwa danej usługi. W mojej ocenie, jeżeli wymagamy od kogoś złożenia oświadczenia, to jeżeli chodzi o to, czy składa on je w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego, czy składa je na odległość, to myślę, że poziom bezpieczeństwa jest bardzo, bardzo podobny i w związku z tym tutaj dalsze zmiany nie są konieczne.

Chciałbym, żeby on był jak najwyższy.

W związku z tym w naszej ocenie lepiej jest robić pewne rzeczy w sposób kompletny, aby wszystkie sprawy z danej kategorii mogły być załatwiane w ten sposób.

To jest relatywnie prosta kwestia, relatywnie prosta konfiguracja, tak że liczymy na to, że w tym terminie się zmieścimy.

Pan poseł Kwiatkowski mówił, że brakuje informacji na ten temat. Popracujemy nad tym.

Zachęcam do oglądania.

To, co tutaj prezentujemy, to funkcjonalność, która z punktu widzenia obywatela już funkcjonuje.

Dotyczy to sytuacji, w której kopia cyfrowa załączona do wniosku jest w jakiś sposób zdaniem osoby rozpatrującej nieczytelna bądź są wątpliwości co do jej autentyczności. Myślę, że jest to racjonalne rozwiązanie. Pan poseł dopytywał też o to, kiedy mObywatel będzie mógł funkcjonować w Sejmie.

Pani poseł Pępek pytała o to, dlaczego ponownie trzeba będzie się ustawiać w kolejce po dowód osobisty. Szanowni państwo, to wynika z przepisów europejskich, które wymagają od nas wprowadzenia drugiej cechy biometrycznej.

To, że będziemy mieli bezpieczniejsze dowody, jest warte tego, żeby tę jedną dodatkową wizytę w urzędzie odbyć. Pan poseł Lorek pytał, czy nie możemy przyspieszyć cyfryzacji aktów stanu cywilnego. Wczoraj zespół programowania prac rządu wpisał bardzo ważną z tego punktu widzenia ustawę dotyczącą cyfryzacji całego procesu związanego z wystawianiem aktów zgonu i z organizacją pochówku. Myślę, że będzie to bardzo ciekawy i oczekiwany przez wiele osób projekt.

Natomiast częścią Polskiego Ładu w ramach komponentu CyberPoland 2025 jest zwolnienie z wszelkiego rodzaju opłat skarbowych w przypadku czynności, które będą realizowane w postaci e-usługi, i rzeczywiście myślę, że to będzie dobry moment na to, żeby porozmawiać o pewnym modelu finansowym.

Natomiast jeżeli chodzi o zwolnienie z opłat, to w naturalny sposób to dotyczy bardziej tych czynności urzędowych niż tych w sądach, ponieważ w sądach, jak wiemy, te opłaty mają też trochę inny charakter i one tam często są uzależnione od rodzaju sprawy itd. Mam wrażenie, że to są wszystkie pytania, które padły w tej debacie. Bardzo za nie dziękuję. I dziękuję za te deklaracje wsparcia dla naszego projektu. Dziękuję, panie ministrze. Pan poseł Grzegorz Napieralski w trybie.

Pan mówi o tych rekompensatach i faktycznie tak jest, bo ta usługa będzie tak samo jak w banku, ona się będzie odbywała bez ludzi, tak jak dokonujemy przelewu przez aplikację czy za pomocą strony internetowej. Natomiast nam chodziło dokładnie o to, że jednak gminy planowały sobie, bo daną usługę wcześniej wykonywała albo pani, albo pan.

Znaczy, ja bym jednak (Dzwonek) szukał rozwiązania, panie ministrze, żeby gdzieś to.

A więc warto by było, myślę, nad tym pracować.

Dziękuję za zaproszenie do oglądania seriali w Telewizji Polskiej, ale chciałem się panu ministrowi zrewanżować apelem o doprowadzenie do sytuacji, w której aplikacja mObywatel, czyli te elektroniczne, wirtualne dowody osobiste, będzie akceptowana choćby przez państwowe banki, bo żaden bank, z tego, co mi wiadomo, nie honoruje np. w trakcie podpisywania umów kredytowych czy jakichkolwiek umów aplikacji mObywatel i dowodów tożsamości w tym trybie, nazwijmy to, ujawnianych. Wydaje się, że to jest trochę poważniejszy problem niż seriale, przy całym szacunku i sympatii dla jakichkolwiek seriali jakiejkolwiek stacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Czy pan minister chciałby coś. Wszystko jest okej. Dziękuję serdecznie. Tryb tych dyskusji jest właściwie znany.

Proszę państwa. Do tej godziny, do której pani poseł będzie na sali. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1510) Proszę pana posła Jarosława Krajewskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu grupy posłów wnioskodawców przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, druk nr 1510. To jest projekt ustawy, który zdecydowanie ułatwia przedsiębiorcom prowadzącym skład podatkowy funkcjonowanie, likwiduje bariery akcyzowe i jest jak najbardziej pożądany i oczekiwany przez tych przedsiębiorców, którzy w ramach działalności związanej ze składami podatkowymi prowadzą na co dzień działalność związaną z wyrobami akcyzowymi. Ale ad rem. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym umieszczenie wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym umożliwia wszczęcie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Jedną z przesłanek zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy jest cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Celem projektowanej ustawy jest umożliwienie kontynuacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym. Sytuacja taka może wystąpić w przypadku zbycia prawa własności nieruchomości, na której znajduje się skład podatkowy, na rzecz nabywcy, który w tym samym miejscu będzie prowadzić skład podatkowy. Obecnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają kontynuację działalności w formie składu podatkowego przez inny podmiot niebędący następcą prawnym podmiotu dotychczas prowadzącego skład podatkowy. W składach podatkowych typu produkcyjnego, w związku z koniecznością zakończenia działalności i rozliczenia się z podatku akcyzowego w wyniku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, trzeba przerwać cały proces produkcji. Podmiot, który chciałby przejąć ten skład podatkowy wraz z wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, obecnie nie ma takiej możliwości prawnej. Wyjątek od tej zasady dotyczy wyłącznie następców prawnych, tj. podmiotów, które wstępują w prawa i obowiązki dotychczasowego podatnika w przypadku połączenia, przejęcia, przekształcenia lub podziału. W innych przypadkach zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga cofnięcia zezwolenia akcyzowego dotychczasowemu podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy i wydania nowego zezwolenia akcyzowego nowemu podmiotowi. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego wiąże się z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wszystkich wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym w dniu cofnięcia zezwolenia, co oznacza dla takiego przedsiębiorcy konieczność zapłaty akcyzy od tych wyrobów. Obecnie obowiązujące regulacje mogą zatem stanowić barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej i celem wnioskodawców jest likwidacja tych barier. Projektowana nowelizacja pozwoli na przejęcie składu podatkowego w innych przypadkach niż sukcesja podatkowa, bez konieczności likwidacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym i zapłaty akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Jeżeli mówimy o tych proponowanych rozwiązaniach, one likwidują trudności w zakresie przejęcia składu podatkowego, eliminując szereg bardzo pracochłonnych i kosztochłonnych działań po stronie firm poszerzających swoje składy podatkowe lub kontynuujących działalność w miejsce poprzednika w reżimie składu podatkowego w sposób nieprzerwany, harmonijny. Możemy określić to jako takie płynne przejęcie i kontynuację działalności. Skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne proponowanych zmian będą pozytywne zarówno z punktu widzenia podatników, ułatwiając ich funkcjonowanie, jak i Skarbu Państwa zasilanego daninami publicznymi będącymi efektem działań dobrze prosperujących przedsiębiorstw. Przygotowanie się do tych nowych regulacji, zarówno po stronie administracji skarbowej, jak i po stronie przedsiębiorców, nie wymaga dodatkowego, zbędnego czasu i dłuższego vacatio legis, w związku z czym uzasadnione wydaje się wejście w życie projektowanej ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje, co chciałbym podkreślić, wzrostu wydatków po stronie budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projektowana regulacja potencjalnie powinna wpłynąć pozytywnie na działalność tych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić skład podatkowy. Dla pozostałych przedsiębiorców należących do tych grup ta regulacja przedstawiona w projekcie ustawy będzie neutralna. W związku z powyższym wnoszę i proszę o to Wysoką Izbę, żeby przyjąć przedstawiony projekt ustawy, który, jeszcze raz podkreślę, będzie bardzo pozytywny dla tych przedsiębiorców, którzy dzisiaj prowadzą składy podatkowe. Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. I zapraszam pana posła Marka Suskiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Proszę o zabranie głosu. Jest pan poseł. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt prezentować stanowisko klubu odnośnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Tutaj pan poseł, który jest wnioskodawcą, dość dokładnie powiedział, co jest celem projektu. Ja mogę tylko powiedzieć, że jest to. projekt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmiotów prowadzących działalność w formie składu podatkowego. I jednocześnie zmiana ewentualnie nazwy podmiotu czy zmiana prowadzącego ten skład podatkowy, który wobec dzisiejszych obowiązujących przepisów co do zasady nie zezwala na taką kontynuację działalności, powodowałaby konieczność płacenia podatku akcyzowego, mimo że ten podatek akcyzowy według naszych przepisów i przepisów Unii Europejskiej jest płacony w momencie wprowadzenia towaru do konsumpcji, a nie w przypadku chociażby zmiany prowadzącego czy zmiany właściciela gruntu itd. A zatem ten przepis ma na celu ułatwienie dla przedsiębiorców, również dla urzędników - i skarbowych, i tych, którzy prowadzą interpretację przepisów - żeby na podstawie tej ustawy ten podatek był nadal płacony w sytuacji, kiedy jest wprowadzany do konsumpcji. Stąd też klub Prawa i Sprawiedliwości uważa te przepisy za godne poparcia i oczekiwane, tak jak mówię, przez wielu przedsiębiorców. Ten projekt ponadto jest projektem, który nie wchodzi w zakres przepisów Unii Europejskiej. Mamy tutaj też ekspertyzy Biura Studiów i Analiz, zlecone opinie, które mówią o tym, że jest on zgodny z przepisami Unii Europejskiej, w związku z czym może być też wprowadzony bez konsultacji czy jakiejś nostryfikacji w Unii Europejskiej. Stąd też popieramy ten projekt jako projekt wspierający polską przedsiębiorczość. Powiem też o oczekiwaniu, żeby w Polsce nie wzrastały podatki, że ten projekt też takich podatków uniknie. Te wszystkie osoby, które prowadzą składy podatkowe, akcyzowe, nie będą musiały takiego podatku prowadzić. A te składy podatkowe prowadzą przedsiębiorcy, którzy trudnią się obrotem towarów akcyzowych bądź ich produkcją albo magazynowaniem, więc w tym przypadku budżet państwa niczego nie straci, a przedsiębiorcy będą mogli bez przeszkód prowadzić działalność. Dlatego popieramy ten projekt i prosimy Wysoką Izbę o wsparcie nas w tych działaniach korzystnych dla polskiej gospodarki. Dziękuję bardzo panu posłowi. Pan poseł Paweł Poncyljusz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Podziwiam posłów Prawa i Sprawiedliwości, że są tak oświeceni, że z własnej woli wnieśli projekt ustawy o podatku akcyzowym. Podziwiam również władze Sejmu, że o podatku akcyzowym rozmawiają posłowie komisji energii, klimatu i Skarbu Państwa. A to oznacza, panie pośle, znamy się z wszystkimi posłami wnioskodawcami albo z wieloma, że tak naprawdę nie chodzi o żadnych przedsiębiorców, nie wiem, winiarzy z Podkarpacia, Małopolski, Dolnego Śląska czy Lubuskiego, którzy prowadzą takie składy podatkowe i od wielu lat sygnalizowali Ministerstwu Finansów, że problem z zamykaniem pewnej branży generuje konsekwencje natychmiastowego zapłacenia akcyzy. To jest kolejny lex Obajtek. Dlaczego? Bo jest planowane konsolidowanie Lotosu z Orlenem i w ramach decyzji Komisji Europejskiej trzeba będzie zbyć część aktywów Lotosu. I tylko z tego powodu państwo przypomnieliście sobie o przedsiębiorcach, o których piszecie, małych i średnich, ale nie piszecie o tym największym przedsiębiorcy, który prawdopodobnie wam napisał tę ustawę, czyli o Orlenie, który potrzebuje tej ustawy, ponieważ dobrze wie, że jeżeli przejmie Lotos i będzie musiał odsprzedać część tych aktywów, to Lotos musiałby zapłacić ciężkie pieniądze, akcyzę, za to, że zamyka takie składy podatkowe, bo naliczanie tej akcyzy odbywa się absolutnie tego dnia.

Może jeszcze jakieś firmy od parówek albo od czegoś i okaże się, że faktycznie przedsiębiorcom coś lepszego wysmażymy jako Sejm. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jedyna ustawa, którą pod prezesa Obajtka i te wszystkie mocarstwowe pomysły PiS-u integrowania wszystkiego wokół Orlenu będziemy mieli i mieliśmy. Mieliśmy już ustawę o rynku mocy, bo trzeba było zamieść problem kontraktu mocowego dla elektrowni Ostrołęka, który nie jest w stanie się zdarzyć w czasie, w którym deklarowała Ostrołęka. Będziemy mieli za chwilę ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu. Chodzi o to zmniejszenie, podniesienie limitu, kiedy jest konieczność odkupu akcji od mniejszościowych udziałowców, bo to będzie też dotyczyło Lotosu. A prawdopodobnie potem będziemy mieli zmianę Prawa geologicznego i górniczego, bo będzie trzeba coś zrobić z tymi koncesjami, które PGNiG ma od lat 60., prawie 200 szt., i które nie przechodzą w sposób automatyczny na Orlen, jeżeli będzie chciał przejąć PGNiG.

Sama zmiana jest dobra dla przedsiębiorców i tu akurat zgadzam się z panami. Tylko wy nie mówicie o tym, po co to robicie. Wy to robicie tylko dlatego, że będzie problem, że Lotos miałby zapłacić jakiś podatek. Gdyby to nie było przedmiotem tej zmiany, to byście nigdy się nie pochylili nad tymi przedsiębiorcami, o których tak piszecie w uzasadnieniu, że ci drobni, mali przedsiębiorcy będą mieli lżej. Może będą mieli winiarze z Podkarpacia czy Dolnego Śląska, ale to nie oni są głównymi beneficjentami. I wiecie dobrze, że można było tę sprawę załatwić dużo wcześniej.

I poza banałami, ogólnymi pohukiwaniami na opozycję nigdy nie pokazano efektu, w którym połączenie Lotosu, Orlenu i PGNiG da większą moc do transformacji energetycznej, do budowania bloków gazowych, do budowania instalacji na odnawialne źródła energii, farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych. To jest tylko taka trochę zabawa w biznes, którą przeprowadza Prawo i Sprawiedliwość i jego menedżerowie (Dzwonek) i nie wiem, czy tak naprawdę przy większej organizacji moce na transformację energetyczną, bo o to podobno chodzi w Orlenie, będą takie, jak się zakłada.

W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie nasze stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zawarte w druku nr 1510. Omawiany dziś przez nas projekt wprowadza zmiany w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Przyjmowana jest regulacja umożliwiająca kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot. Według wnioskodawców nie będzie konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Z uzasadnienia ustawy wynika, że taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku zbycia własności nieruchomości, na której znajduje się skład podatkowy, na rzecz nabywcy, który w tym miejscu będzie prowadził swój skład. I tak jak powiedział mój przedmówca, być może dzisiaj przedłożenie tego projektu ustawy jest elementem rozwiązania problemu Lotosu i Orlenu oraz kosztów, które musiałyby być zapłacone w momencie zbycia tej części nieruchomości i znajdującego się tam paliwa, a więc zapłacenia akcyzy. Zaproponowane rozwiązanie jest od dawna oczekiwane przez wiele małych podmiotów gospodarczych prowadzących właśnie taką działalność. Zwracali oni uwagę na brak możliwości kontynuacji działalności przez następcę prawnego podmiotu, który wcześniej nie prowadził składów podatkowych poprzez zakup nieruchomości. Obecnie podmiot przejmujący istniejący skład podatkowy wraz z wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie ma takiej możliwości, oczywiście z wyjątkiem następców prawnych. Czym są składy podatkowe i jak otrzymuje się zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego? Produkujesz, magazynujesz wyroby akcyzowe, np. napoje alkoholowe, paliwo lub papierosy, i nie chcesz płacić akcyzy. Wyroby sprowadzasz z zagranicy bez podatku akcyzowego, ktoś zlecił ci usługowe wykonywanie tej czynności. Aby to zrobić, musisz mieć zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu składu podatkowego. Zatem skład podatkowy jest miejscem, w którym mogą być produkowane, przetwarzane oraz magazynowane wyroby akcyzowe bez konieczności zapłaty akcyzy do momentu wprowadzenia danych wyrobów z systemu zawieszenia poboru opłat akcyzy. W efekcie przemieszczanie wyrobów akcyzowych z użyciem składu podatkowego powoduje odroczenie płatności podatku akcyzowego ciążącego na wspomnianych wyrobach i przenosi ten obowiązek na okres, w którym wyroby opuszczają skład w celu ich wprowadzenia do swobodnego obrotu. Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, wnioskujący o to podmiot gospodarczy musi spełnić wiele wymagań: złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu, przedstawić dokumenty odnośnie do tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona ta działalność, przedłożyć plan składu, złożyć zabezpieczenie akcyzowe. Jest to proces długotrwały i rozumiem dzisiaj przedsiębiorców, którzy przejmując taką nieruchomość, chcą, aby ta procedura została skrócona, a druga strona nie musiała płacić tak dużej kwoty, jeśli tam w wyniku produkcji zostały, powiedzmy, te materiały bądź jeśli są one na składzie. Zaproponowane regulacje ustawowe pozwolą we wszystkich przypadkach, w których nie mamy do czynienia z sukcesją podatkową uniwersalną, na przejęcie składu podatkowego przez inny podmiot bez konieczności likwidacji działalności prowadzonej w przejmowanym składzie i zapłaty akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Zatem to rozwiązanie zapewni ciągłość działalności w składzie produkcyjnym, w tym stosowania procedury akcyzy w przypadku składu podatkowego typu produkcyjnego, a być może czasami zatrzymanie ludzi, którzy tam pracowali, a musieliby być zwalniani. Przedsiębiorcy zwracają uwagę właśnie na trudności dotyczące głównie działalności prowadzonej w składzie podatkowym typu produkcyjnego, w którym w związku z zakończeniem działalności gospodarczej i rozliczaniem się z podatku akcyzowego w wyniku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy przedsiębiorcy muszą przerwać cały proces produkcyjny. Obecnie przepisy co do zasady nie zezwalają na kontynuację działalności w składzie podatkowym przez inny podmiot niż dotychczasowy, prowadzący skład podatkowy. I tą ustawą panowie posłowie, którzy złożyli ten projekt, to zmieniają. Zgodnie z dziś obowiązującą ustawą z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na prowadzenie składu podatkowego następuje zakończenie procedury poboru akcyzy. Oznacza to, że przedsiębiorca tam funkcjonujący jest zmuszony zapłacić czasami bardzo wielkie kwoty. To ma się zmienić.

Bardzo proszę, pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Dyskutujemy dziś o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Projektodawcy przekonują, że na zmianie przepisów skorzysta wielu przedsiębiorców, i to jest ważne. Szkoda, że nie wymienia się tu obszarów, sektorów, których to najbardziej dotyczy. Mówiąc o przedsiębiorcach, mam na myśli podmioty, które produkują, składują bądź przetwarzają wyroby określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 47 ustawy o podatku akcyzowym produkcja takich towarów musi odbywać się w składzie podatkowym. Dopóki towary nie zostaną wyprowadzone ze składu podatkowego, dopóty nie ma konieczności zapłaty podatku. Według projektodawców proponowane rozwiązania mają wychodzić naprzeciw podatnikom i być dla nich korzystne. Ponadto wprowadzenie nowych przepisów ma sprawić, że nie będzie występować sytuacja alokowania czasu koniecznego na przygotowanie się do nowych regulacji ani po stronie administracji skarbowej, ani po stronie przedsiębiorców. Projektodawcy uznają, że proponowane zmiany będą pozytywne zarówno z punktu widzenia podatników, ułatwiając ich funkcjonowanie, jak i szerzej, dla Skarbu Państwa zasilanego daninami publicznymi będącymi efektem działań przedsiębiorstw.

Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym ujętego w druku nr 1510. Wysoka Izbo! Celem projektu jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które umożliwią kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, ale bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym. Obecnie obowiązujące przepisy co do zasady nie zezwalają na kontynuację tej działalności w składzie podatkowym przez inny podmiot niż dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bowiem zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, co oczywiście oznacza, że ta akcyza musi zostać uregulowana. Te regulacje rzeczywiście pozwolą we wszystkich przypadkach, w których nie mamy do czynienia z sukcesją uniwersalną, na przejęcie tego składu w praktyce przez inny podmiot bez konieczności likwidacji tej działalności, czyli bez konieczności de facto zapłaty tej akcyzy w całości, co oczywiście może być uciążliwe. Powstaje pytanie.

Nie należy natomiast zapominać, że są wielkie pytania o to, czy ta fuzja jest korzystna dla naszej gospodarki, dla naszego państwa, czy wprost przeciwnie - szkodzi naszemu państwu i szkodzi gospodarce. Myślę, że z tym pytaniem musimy zaczekać na odpowiedź. Natomiast na pewno przydałaby się w tym obszarze głębsza, bardziej merytoryczna dyskusja, do czego zachęcam, a równocześnie zgłaszam wniosek o przekazanie do właściwej komisji tego projektu ustawy celem dalszego procedowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Jeśli ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania, to bardzo proszę to zrobić. Zamykam listę. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. 1 minuta na zadanie pytania. Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Komisjo!

Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości pójdzie za tropem i wskazaniem swojego lidera pana prezesa Kaczyńskiego (Dzwonek) i dojdzie do obniżenia stawki akcyzy na paliwa, dzięki czemu Polacy będą mogli płacić mniej na stacjach benzynowych? Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Wysoka Izbo! Sam zamysł zmiany ustawy o podatku akcyzowym należy uznać za dobry, a proponowane rozwiązania za celowe i potrzebne.

W grę mogą tutaj wchodzić ogromne kwoty, których pobór został czasowo zawieszony. Czy takie rozwiązanie nie stworzy zdaniem rządu mechanizmu, który zostanie wykorzystany w sposób niezgodny z prawem, co mogłoby prowadzić do uszczuplenia należnego podatku akcyzowego? Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Wiesław Szczepański, Lewica. Czy mógłby pan powiedzieć, ile dzisiaj przedsiębiorstw czy podmiotów gospodarczych prowadzi skład podatkowy w rozróżnieniu na branżę paliwową, papierosy, alkohole? Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska.

Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Ceny paliw na stacjach benzynowych wzrosły o 29%.

Jak mówili moi przedmówcy, prezes Kaczyński powiedział, że można obniżyć podatki, aby te ceny były niższe, bo ok. 59% ceny tych artykułów to są podatki, w tym podatek akcyzowy.

To jest po prostu skandaliczne. A obywatele czekają, aż wreszcie to obniżycie i będziecie słowni w tym, co robicie.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Chciałabym się dowiedzieć, ile w Polsce mamy zarejestrowanych składów podatkowych. Szczególnie chciałbym się dowiedzieć, jak dużą grupę przedsiębiorstw obejmuje dzisiaj omawiany projekt ustawy. Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Celem projektu jest wprowadzenie regulacji umożliwiających kontynuowanie działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot w składzie podatkowym. Projekt jest jak najbardziej dobry dla przedsiębiorców, ale dotyczy ogromnych kwot podatku akcyzowego. I czy to nie jest projekt napisany przez pana prezesa Obajtka na jego potrzeby w związku z połączeniem Orlenu i Lotosu?

Wysoka Izbo! Zacznę od odpowiedzi na pytania pana posła Suchonia i pani poseł Skowrońskiej odnośnie do obniżki akcyzy na paliwo. Już teraz wysokość akcyzy w Polsce jest na poziomie nieznacznie wyższym od poziomu minimum unijnego, tak że nie ma tutaj szerokiego pola do dokonania obniżki, która skutkowałaby zmniejszeniem cen paliwa na stacjach. Tym bardziej że chcielibyśmy gorąco podkreślić, że ceny paliwa w Polsce już teraz są na poziomie jednych z najniższych cen w Unii Europejskiej.

To wszystko podmioty, które szczególnie teraz, w dobie pandemii, sytuacji COVID-owej, mogą być zainteresowane tym, żeby dokonywać pewnych zmian w swojej strukturze właścicielskiej, łączyć się z innymi podmiotami, tak żeby w lepszy sposób przetrwać pewne zmiany na rynku, jakie aktualnie zachodzą. Wprowadzane teraz, proponowane przez państwa posłów zmiany zdecydowanie ten proces ułatwią. Skończą się sytuacje, w których w przypadku łączenia firm w sposób inny niż sukcesja uniwersalna dochodzi do zapłaty akcyzy od produktów, które nie zostały sprzedane, nie zostały wyprowadzone ze składu akcyzowego.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo!

Zwracam uwagę na to, że tutaj nie wydzielamy składów podatkowych i nie rozróżniamy pojedynczych przedsiębiorców - tak żeby wskazać, że jakakolwiek grupa przedsiębiorców zostałaby pominięta.

Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zawarty w druku nr 1510, do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Marszałek Sejmu proponuje, aby Sejm na podstawie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu wyznaczył termin przedstawienia sprawozdania umożliwiający rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1530) Proszę minister rodziny i polityki społecznej panią Marlenę Maląg o zabranie głosu.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci została wprowadzona do polskiego systemu prawnego i wprowadziła nowe świadczenie „Rodzina 500+”, potocznie nazywane 500+. Program „Rodzina 500+” jest jednym z flagowych programów rządu stanowiący fundament wsparcia polskich rodzin. Ale jest przede wszystkim dowodem troski naszego rządu o rodzinę, o inwestycje w rodzinę.

W ramach programu „Rodzina 500+” rodzice otrzymują świadczenie na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Jest to jeden z czynników, który wspiera rodziny w podejmowaniu decyzji o tym, że rodzą się kolejne dzieci. Od początku realizacji tego programu do polskich rodzin jako inwestycję w rodzinę przekazaliśmy ponad 156 mld zł. Obecnie ten program jest obsługiwany przez jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast proces optymalizacji, usprawniania realizacji zadania, który przerobiliśmy w tym roku w związku z programem rządowym „Dobry start” i innych programów w czasie pandemii koronawirusa, spowodował, że możemy ten program usprawnić, jeżeli chodzi o jego realizację.

Tak jak państwu przed chwilą powiedziałam, koszty obsługi tego programu przez samorządy w roku 2020 wyniosły ponad 326 mln zł.

Wprowadzamy w ramach optymalizacji możliwość składania wniosków tylko drogą elektroniczną, a więc poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez system Emp@tia ministerstwa rodziny, poprzez bankowość elektroniczną.

W zeszłym roku o tej samej porze było 300 tys. wniosków mniej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł porozumienia z Pocztą Polską, z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zorganizował mobilne punkty i rodzice dzieci, którzy mogą ubiegać się o świadczenie i „Dobry start”, a więc to jest ta sama grupa rodziców, która będzie mogła ubiegać się o świadczenie 500+ drogą elektroniczną, nie mają problemu z dostępem do usług. Dlatego też to usprawnienie spowoduje, że w budżecie państwa z jednej strony będziemy mieli oszczędności, ale te oszczędności już planujemy, aby dalej były przekazywane na nowe programy, które będą dedykowane dla polskich rodzin. W piątek będziemy tutaj razem z panią minister prezentować państwu nową ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym, która te pieniądze przekaże już na kolejne wsparcie dla polskich rodzin. W ustawie, którą państwu przedstawiamy, również wprowadzamy zmiany w ramach koordynacji świadczeń, czyli wypłaty świadczenia, jeżeli jest potrzebna koordynacja międzynarodowa, jeżeli rodzice migrują. Wielokrotnie państwo też jako parlamentarzyści zwracaliście się do nas o usprawnienie tego procesu, bo rodzice czekają długo na wypłatę tego świadczenia. Wprowadzamy też w ramach obowiązujących przepisów automatyzację wypłaty świadczeń koordynowanych, aby przede wszystkim wspierać jak najskuteczniej, jak najszybciej polskie rodziny, bo na tym nam bardzo zależy, bo na budowaniu silnej polskiej rodziny chcemy opierać przede wszystkim budowę silnego polskiego państwa. Będziemy wprowadzali, tak jak powiedziałam, od 1 stycznia automatyzację tego procesu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Te wnioski, które są obsługiwane przez samorządy do zakończenia obecnego okresu, będą realizowały jeszcze samorządy. Podobnie też jak w przypadku koordynacji, wojewodowie zamkną okres świadczeniowy i rozpocznie Zakład Ubezpieczeń Społeczny od nowego okresu świadczeniowego. Wnioski rodzice będą składali elektronicznie w okresach rozliczeniowych. Tak jak państwu tutaj przytoczyłam, przerobiony w tym roku program „Dobry start” na zasadzie automatyzacji, optymalizacji tych procesów usprawnienia przede wszystkim został przez rodziców dobrze przyjęty, mamy konkretne efekty szybkiego działania. Możemy też przytoczyć pozytywne działania. To jest tak naprawdę wyzwanie współczesnego czasu, a COVID jeszcze nam pokazał, że sprawne, funkcjonujące państwo, a więc wprowadzanie narzędzi szybkiego wsparcia poprzez elektroniczne składanie wniosków. Pamiętacie państwo, wprowadzaliśmy dodatek solidarnościowy dla osób, które traciły pracę, też była to tylko droga elektroniczna, szybko, sprawnie obsłużony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także bon turystyczny, który był wsparciem zarówno dla polskich rodzin, jak i dla branży turystycznej. Dlatego też, szanowni państwo, przede wszystkim kierując się postępem czasu i sprawnością, państwo powinno realizować sprawnie swoje zadania, podjęliśmy taką decyzję jako rząd, aby przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy o zmianie świadczenia „Rodzina 500+” w zakresie realizacji obsługi. Program jest nadal powszechny i bez kryterium dochodowego 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia. Dlatego prosiłabym wysoką radę o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1530. Wysoka Izbo! Rząd Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzając w 2016 r. świadczenie wychowawcze 500+, przyczynił się do poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należyty priorytet, gdyż polityka prorodzinna jest inwestycją w przyszłość naszego państwa. Wsparcie to przekłada się na poprawę zarówno sytuacji finansowej, jak i jakości życia rodzin. Co ważne, o czym wspomniała pani minister, nowelizacja ustawy w żaden sposób nie ograniczy ani nie zmieni kręgu osób uprawnionych w przypadku wysokości przyznawanych świadczeń. Procedowany dziś projekt ustawy dotyczy m.in. powierzenia obsługi programu „Rodzina 500+” Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, co wpłynie na zmniejszenie kosztów obsługi programu i pozwoli zaoszczędzić w przeciągu dekady ponad 3 mld zł. Przyjęcie proponowanych rozwiązań spowoduje istotne odciążenie samorządów, co pozwoli na efektywniejsze realizowanie innych zadań ustawowych, w szczególności w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Kolejną wprowadzoną zmianą jest możliwość złożenia wniosku tylko za pośrednictwem Internetu.

Do tej pory niemal 4,2 mln dzieci zostało zgłoszonych do skorzystania ze świadczenia programu 300+. Zmiana formy wynika przede wszystkim z obserwacji, które wskazują na znaczący coroczny wzrost dotyczący wykorzystania elektronicznych kanałów składania wniosków. W razie braku możliwości - to jest bardzo ważne - złożenia wniosku drogą elektroniczną, analogicznie do przypadku programu „Dobry start”, rodzice będą mogli skorzystać z pomocy pracownika ZUS. Procedowana ustawa przewiduje również zmianę sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego. Dotychczasowe świadczenie, które było wypłacane w sposób wybrany i wskazany przez organ właściwy, np. poprzez przelew środków na konto bankowe wskazane we wniosku, wypłatę świadczenia w kasie urzędu czy przekazanie kwoty świadczenia przekazem pocztowym, zostanie zastąpione, jako że nowelizacja ustawy wprowadza wypłatę świadczeń wyłącznie w formie bezgotówkowej. Zmiana ta ma na celu uzyskanie oszczędności po stronie kosztów związanych z dystrybucją świadczenia i uproszczenie procesu, gdyż zaledwie w przypadku niespełna 2% osób wypłata świadczenia odbywa się w innej formie niż przelew na rachunek bankowy.

Podsumowując, celem zmian jest wyłącznie optymalizacja procesu obsługi świadczenia poprzez wykorzystanie coraz bardziej powszechnych narzędzi, jakimi są systemy informatyczne, oraz położenie nacisku na bezgotówkowe formy wypłaty świadczenia wychowawczego, a także dążenie do zmniejszenia kosztów związanych z przyznawaniem i przekazywaniem uprawnionym środków pieniężnych poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Koalicja Obywatelska zaprezentować stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1530. Informacja, że ZUS ma od 2022 r. wypłacać środki z programu „Rodzina 500+”, doprowadziła urzędników na skraj wytrzymałości i w sierpniu br. skłoniła aż sześć związków zawodowych w tej instytucji do wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą, a to jest prosta droga do strajku. Jak mówią: Frustracje narastały przez lata, ale jeszcze nigdy urzędnikom ZUS nie dołożono tak wielu obowiązków w tak krótkim czasie. Tarcze nas pogrążyły, nie otrzymaliśmy etatów w związku z obsługą programu „Dobry start”, zajmujemy się realizacją bonów mieszkaniowych, dojdzie teraz 500+, a w perspektywie jest jeszcze program „Kapitał opiekuńczy”, czyli 12 tys. zł na każde nowo narodzone drugie dziecko i na kolejne dzieci. Ostatnie miesiące swojej pracy podsumowują tak: 35 stopni w pokoju, brak klimatyzacji, brak wody do picia, płaca minimalna, obowiązkowe nadgodziny i gigantyczna presja ze strony państwa i obywateli. A na to wszystko prezes ZUS odpowiada w mediach - i to oburza urzędników najbardziej - że instytucja jest tak scyfryzowana, iż większość działań przeprowadza się tam za pomocą zaledwie jednego kliknięcia. Automaty robią może 30% roboty, reszta jest przerabiana przez nas, ludzi - mówią. System informatyczny jest niewydolny i nieprzystosowany do ilości spraw, które musi przerobić. Z każdym kolejnym dorzucanym przez rząd programem jest coraz bardziej przeciążony i zawiesza się na całe dni, całkowicie uniemożliwiając urzędnikom pracę. Pracownicy ZUS mówią: żeby przesłać płatnikowi pismo przez aplikację, muszę wylogować się z dwóch innych, inaczej nie pójdzie. Gdy system pada w poniedziałek, to dopiero w środę centrala wydaje zalecenie, żeby zaczynać od spraw pilnych, a tych niepilnych nie robić. 35 spraw emerytów i rencistów do zrealizowania w ciągu tygodnia z powodu awarii systemu, a od poniedziałku do środy można zrobić najwyżej pięć wniosków. Przecież w ogóle nie przystajemy do naszych czasów. Nie jesteśmy przystosowani do zadań, które mamy na dziś. Jeśli nam dołożą 500+, to będę musiała przynieść swój komputer z domu. Biurka poklejone taśmą, bo drzazgi w palce wchodzą. Rolety kupiliśmy sami, bo nic już na monitorach nie było widać. Wysokość monitora wyregulowałam sama dwoma ryzami papieru. Notatniki i długopisy mam też swoje, z domu. Czy będzie komu kolejne dodatkowe zadania wykonywać, jeśli dojdzie do strajku, a liczba zwalniających się pracowników zwiększy się jeszcze bardziej niż teraz? A przecież w związku ze zmianą i wdrożeniem nowych rozwiązań polegających na tym, iż wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną, deklarują państwo pomoc w okresie składania wniosków, a więc komputery w jednostkach ZUS, asystę pracownika ZUS przy składaniu wniosku drogą elektroniczną, otwarcie dodatkowych punktów składania wniosków w innych placówkach czy urzędach, np. na poczcie, czy w KRUS. Takich miejsc ma być na terenie kraju ponad 8 tys. Kto będzie realizował te zadania związane z pomocą w wypełnianiu wniosków drogą elektroniczną? Na kogo spadną te obowiązki? Znowu, jak w przypadku pracowników ZUS, zostaną one przerzucone na kolejnych urzędników kosztem wykonywania i realizacji innych podstawowych obowiązków? Zatrudniono i przeszkolono pod względem obsługi programów prawie 12 tys. pracowników samorządowych, którym w związku z proponowanymi przez rząd zmianami grożą masowe zwolnienia. Rząd uważa, iż ta zmiana pozwoli na odciążenie samorządu terytorialnego od realizacji zadań o charakterze cyklicznym i akcyjnym, czyli corocznego procesu związanego z przyjmowaniem i rozpatrywaniem milionów wniosków. To wytłumaczenie jest co najmniej dziwne z uwagi na fakt, że może okazać się, iż nie będzie miał kto realizować tych zadań ustawowych. Czyli tak: zwalniamy pracowników samorządowych, a dokładamy dodatkowe obowiązki lub zatrudniamy pracowników w instytucjach państwowych. To bardzo wygodne zmieniać przepisy, a odpowiedzialność za losy ludzi, którzy nie są już do obsługi waszego szlagierowego programu potrzebni, zrzucić na samorządy. Bo to na gminy spadnie obowiązek dokonania zmian organizacyjno-kadrowych, gdyż to one są de facto pracodawcami pracowników samorządowych. A przecież środki przekazywane na wykonywanie tego zadania (Dzwonek) stanowią ważny element budżetów gmin. To stała kwota, która ma wpływ na dochody samorządu. W związku z powyższym klub Koalicji Obywatelskiej odnosi się krytycznie do pomysłu przeniesienia systemu wypłat do ZUS. Uważamy, że jest on źle przygotowany, skierowany przeciwko jednostkom samorządu terytorialnego, nie uwzględnia sytuacji pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będziemy głosowali przeciwko temu projektowi. Bardzo proszę, pani poseł Magdalena Biejat, klub Lewica. Wysoka Izbo! Pani Minister! Muszę powiedzieć, że tyle razy usłyszałam słowo „optymalizacja” dzisiaj w pani wystąpieniu, że poczułam się jak na zebraniu szefów jakiejś wielkiej korporacji. Jest to zaskakujące jak na rząd, który mieni się prosocjalnym. Cóż, dużo było o tym: reorganizacja zadań, restrukturyzacja, przeniesienie obowiązków. Naprawdę brzmi to znajomo. Brzmi to właśnie jak typowe zwolnienia pod kątem optymalizacji, pod pretekstem optymalizacji w dużych firmach. I tutaj też będziemy mieć do czynienia ze zwolnieniami, bo w jednostkach samorządu terytorialnego do obsługi 500+ jest dzisiaj zatrudnionych ponad 11 tys. osób. To są dane z ministerstwa. Pracownicy socjalni szacują na podstawie danych, które spływają do nich na podstawie wniosków z informacji publicznej, że prawdopodobnie od 6 do 7 tys. z tych osób straci pracę. I to, szanowni państwo, też są polskie rodziny. W bardzo wielu miejscach te rodziny, te osoby, które pracują, pracują w małych gminach, w których rynek pracy jest trudny. Są one często jedynymi żywicielami rodziny. Ludzie pobrali kredyty, mają dzieci i stają przed sytuacją, w której pracodawca mówi im dzisiaj: zacznijcie szukać nowej pracy, bo na pewno ją stracicie. Kiedy pisałam interpelację do pani minister i pytałam o to, czy ministerstwo w ogóle myślało o tych ludziach, którzy zostaną zwolnieni, w odpowiedzi dowiedziałam się, że nie, ponieważ jest to problem samorządów, a nie ministerstwa. Najwyraźniej skreślenie w tabelce w Excelu 7 tys. miejsc pracy nie stanowi dla rządu żadnego problemu. Mówiła pani minister również dużo o ZUS-ie i o „Dobrym starcie”, o tym, jak to świetnie poszło. Bo ja tak.

Zapominacie wspomnieć, że te oszczędności - tak - będą, ale odbędą się kosztem pracowników, kosztem pracowników w samorządach, kosztem pracowników w ZUS-ie. Robicie to w dniu, w przededniu wielkich strajków budżetówki, w momencie kiedy pracownicy budżetówki już zaczynają w niektórych miejscach strajkować. Strajkują pracownicy sądów. Strajkują pracownicy ochrony zdrowia. Zapowiadają strajk pracownicy ZUS-u, którzy już weszli w spór zbiorowy, protestując przeciwko fatalnym warunkom pracy, które są właśnie takie. Protestują przeciwko temu, że stają się twarzą coraz mniej wydolnej instytucji, bo ona nie może być wydolna w momencie, kiedy oszczędza się na pracownikach, którzy muszą dostarczać usługi publiczne, za które są odpowiedzialni.

Jednocześnie dokonujecie tej cyfryzacji i przenosicie obsługę programu dalej od tych osób, które takiego wsparcia będą potrzebować.

Fatalne wykonanie kosztem pracowników (Dzwonek), kosztem zwykłych ludzi, kosztem także dużej części polskich rodzin. Bardzo proszę, pani poseł Bożena Żelazowska, Koalicja Polska.

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Otóż pozwólcie państwo, że w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści przedstawię stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z druku nr 1530. W programie Polskiego Stronnictwa Ludowego od wielu lat, a dzisiaj w polityce programowej Koalicji Polskiej polityka prorodzinna, polityka demograficzna zajmuje bardzo ważne miejsce. Wiele rozwiązań, które są dzisiaj przez rząd kontynuowane, zostało wprowadzonych, kiedy ministrem pracy i polityki społecznej był Władysław Kosiniak-Kamysz. Wówczas wprowadzono takie programy jak kosiniakowe, które funkcjonuje również dzisiaj, program dotyczący żłobków, jak też liczne programy finansowe dla seniorów. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego głosował również za wprowadzeniem programu 500+. Mamy świadomość, drodzy państwo, że polityka prorodzinna jest najlepszą inwestycją, bo inwestycją w polską rodzinę, która jest fundamentem silnego państwa. Chcemy, aby polskim rodzinom żyło się dobrze i bezpiecznie. Proponowane w tej ustawie rozwiązania powinny służyć właśnie rodzinie. Jednak zapisy tej ustawy nie są dobre i nie wszyscy będą mogli w pełni z nich skorzystać. Ustawa zakłada szereg rozwiązań teleinformatycznych usprawniających załatwienie spraw.

Główną zmianą będzie powierzenie obsługi programu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Już dzisiaj wiemy, że jest to bardzo złe rozwiązanie i dla rodzin, ale też dla pracowników ZUS-u, którzy protestują, ponieważ i tak są bardzo mocno obciążeni pracą za niewspółmierne wynagrodzenie. Pracownicy ZUS-u nie od dziś piszą do nas, posłów, petycje w tej sprawie. Te środki powinny być tak jak dotychczas dysponowane przez samorządy, które znają sytuację rodzin i mogą zweryfikować, czy kwota będzie wykorzystana w pełni na dziecko. Z perspektywy odległego ZUS-u nie będzie to możliwe. Zabranie możliwości realizacji świadczenia 500+ i wychowawczego wójtom, burmistrzom, prezydentom miast jest też pozbawieniem samorządów znacznej części środków finansowych, a pracownicy tych samorządów po prostu stracą pracę. Kontrowersyjny również w tej ustawie jest zapis zmieniający formułę składania wniosków jedynie przez Internet, a wypłata świadczeń może nastąpić tylko w formie bezgotówkowej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe. Odejście od wypłaty w formie gotówkowej nie pozwoli wszystkim rodzicom czy opiekunom otrzymać należnego wsparcia, bo zwyczajnie, drodzy państwo, wciąż około 15–20% obywateli takiego konta nie posiada. Wątpliwości budzi również efektywność badania przez ZUS przesłanek dotyczących przysługiwania świadczenia, w szczególności wspólnego zamieszkania z dzieckiem i pozostawania dziecka pod opieką matki albo ojca. Gminy są zdecydowanie bliżej rodziny i opiekunów niż ZUS. Ponadto to właśnie gminy przyznają części beneficjentów 500+ także świadczenia rodzinne, więc znają sytuację przynajmniej niektórych rodzin. ZUS takich informacji nie posiada i nigdy się nie pokusi o sprawdzenie. A ucierpią na tym dzieci. Kolejna grupa osób, w wypadku której potrzebne jest prowadzenie poszerzonego postępowania wyjaśniającego, to cudzoziemcy. Pytanie, jak z prowadzeniem takich postępowań wyjaśniających poradzi sobie ZUS. Klub parlamentarny Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe zgłosi w tym zakresie stosowne poprawki. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Krystian Kamiński, Konfederacja.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Głównym celem omawianej regulacji jest przeniesienie obsługi świadczenia 500+ z poziomu samorządu terytorialnego, czyli gmin, do jakże lubianego przez wszystkich, docenianego i całkowicie pozbawionego wad biurokratycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odważna decyzja, muszę przyznać. Zaledwie jeden akapit jest poświęcony samorządom. Zawarte jest w nim twierdzenie, że pozwoli to na istotne odciążenie samorządu terytorialnego, i dalej, że pozwoli im na efektywniejsze realizowanie innych zadań ustawowych, w tym walkę z obecnym zagrożeniem epidemicznym. Właśnie na tym aspekcie chciałbym się skupić. Rozmawiałem z samorządowcami o tej zmianie i nie odnosili się oni do niej przychylnie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że dużą część budżetów gmin stanowiły właśnie środki, które były związane z obsługą tego programu. Zmieni to mocno poziomy budżetów praktycznie wszystkich gmin w Polsce. Zmienią się, co za tym idzie, możliwości inwestycyjne, możliwości zaciągania kredytów, poziomy wkładu własnego do inwestycji. Szczególnie małym gminom, które mogą na tej zmianie stracić najwięcej, w sensie rozwojowym. Jak wiemy, urzędy były również zmuszone zatrudnić nowych pracowników do obsługi programu 500+. I co teraz mają zrobić z tymi urzędnikami? Mają być zwolnieni czy po prostu zająć się czymkolwiek innym? Czy ktoś o tym myślał? Kolejno nasuwają się inne pytania. Ile w związku z tą zmianą będzie musiało być zatrudnionych nowych osób w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Jakie nowe koszty w związku z tym powstaną? Jako zdecydowany plus całej zmiany wskazują państwo, że cały system 500+ będzie praktycznie w pełni zinformatyzowany, łącznie z wypłatą tych pieniędzy. Sytuacja związana z COVID-em pokazała, że gminy jednak radzą sobie coraz lepiej, właśnie w tych kwestiach informatycznych, informatyzacji. Kontakty z mieszkańcami były ograniczone, co nie wpływało de facto na współpracę z nimi. Oczywiście, że mogłaby i dobrze państwo o tym wiedzą, ale jak sami napisaliście, ZUS jest waszym zdaniem instytucją funkcjonującą znakomicie. Sadzę, że ta opinia nie pokrywa się z tym, co większość Polaków sądzi o tej instytucji, delikatnie rzecz biorąc. Ta zmiana jest typowo centralistyczna, czyli taka, którą obecna władza preferuje w wielu aspektach życia społecznego w Polsce. Jest to kolejny krok w celu dobijania samorządów w Polsce pod względem finansowym i odbierania im kolejnych kompetencji. Dziękuję, panie pośle. I bardzo proszę, pani poseł Joanna Mucha, Polska 2050. Pani Marszałek! Pani Minister!

Pani ma obowiązek dbać o ludzi, a tą ustawą uderza pani w trzy grupy polskich obywateli i wywołuje pani naprawdę dramatyczny stres u tych ludzi. Po pierwsze, świadczeniobiorcy.

Jedna z moich przedmówczyń przed chwilą mówiła, że to jest 6 tys. czy 7 tys. osób, które być może zostaną zwolnione. Słyszę z jednostek samorządu terytorialnego, że być może jest to nawet ok. 10 tys., 12 tys. ludzi. Pani ich dzisiaj zwalnia. To jest dbałość o rodzinę? Po trzecie wreszcie, pracownicy ZUS-u. Ci pracownicy, którzy skarżą się już dzisiaj na to, jak dramatycznie są przepracowani.

Do tego dochodzą jeszcze obowiązki stwierdzenia stanu faktycznego, rzetelności pobierania tych świadczeń. Piszecie państwo: jednostki samorządu terytorialnego poprzez swoje ośrodki pomocy społecznej będą nadal to robiły. Ale już bez środków, już bez kosztów pokrytych przez państwo. Powiedzmy wprost: ta ustawa jest po to, żeby władzy było wygodniej. Ale pani minister, rządzenie nie polega na tym, żeby władzy było wygodniej. Rządzenie polega na tym, żeby ludziom było wygodniej. Wam się naprawdę coś pomyliło. 12 tys., 10 tys. osób do zwolnienia. Odprawy, trzynastki, których zapewne nie będzie. Wskaźniki, które polecą. Moi przedmówcy już o tym mówili, że te wskaźniki dotyczące jednostek samorządu terytorialnego stanowią bezpośrednie uderzenie w samorządy. Kolejny temat: system informatyczny. Będę panią pytała w trakcie zadawania pytań, czy ten system informatyczny już został zakupiony, czy dopiero państwo planujecie zakupienie, bezprzetargowo, bo COVID. W tym, żeby zorganizować przetarg? Nie rozumiem. Proszę mi pozwolić. Wypłata na konto. Teraz nagle będzie wypłata na konto. Dosłownie parę tygodni temu tutaj w tej Izbie procedowaliśmy nad ustawą autorstwa pana prezydenta Dudy, w której to ustawie była mowa o tym, że sklepy nie mogą przejść wyłącznie na obrót bezgotówkowy. Czyli jeśli to jest obowiązek po stronie ludzi, to zostaje, ale jeśli jest to obowiązek po stronie państwa, żeby państwo zapewniało obrót gotówkowy i bez gotówkowy, to nie. Bo wam się wydaje, że to wam ma być wygodniej. Naprawdę puknijcie się w głowę. Bardzo proszę, pani poseł Agnieszka Ścigaj, Polskie Sprawy. Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Polskie Sprawy chcę zaprezentować opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Po pierwsze, w wielu wystąpieniach pani minister, ale też i posłów, medialnie i tutaj na tej sali padało właściwe stwierdzenie, że program 500+ jest programem socjalnym, programem, którego głównym celem jest przeciwdziałanie ubóstwu. Trzeba było to zrobić. Rzeczywiście ubóstwo wśród dzieci, szczególnie na wsiach, było dość duże. Wynika to już jasno i wyraźnie ze wskaźników, że dzietności to nam nie poprawiło w żaden sposób.

Niestety tak się dzieje. Nie dotyczy to przeważającej liczby rodzin, ale w części rodzin jest tak, że niestety te pieniądze nie trafiają do dzieci i gdyby nie pomoc społeczna, gdyby nie pracownicy socjalni i np. ta wariantowość dotycząca tego, że w przypadku takich sytuacji można zamienić pomoc finansową na pomoc rzeczową czy zakupić usługi.

Te rodziny wypadają z systemów pomocy społecznej, dlatego że często po prostu nie chcą przyjść do tego ośrodka, skoro mają 500+ i nie muszą być tam zarejestrowane. Często dopiero po długim czasie dowiadujemy się, że może tam się dziać coś niedobrego z dziećmi.

Powiem tylko, że gminy były przygotowane do tego, żeby sprawnie i szybko zbierać informacje, ponieważ mają dostęp do różnych systemów i mogą się dowiedzieć, gdzie dziecko chodzi do szkoły, czy jest opieka naprzemienna, czy świadczenie nie będzie należnie pobrane. Natomiast państwo znowu pewnie zakupicie system bezprzetargowo, jak każdego roku, za 800 mln zł - tyle wydajecie na informatyzację ZUS.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, to już zamykam listę. I jako pierwsza - pani poseł Monika Falej, Lewica. 1 minuta na zadanie pytania. Wysoka Izbo! W ostatnich dniach coraz głośniej jest o tym, że pracownicy ZUS mają dość swoich przełożonych, tj. zarządu i prezesa. Pracownicy skarżą się na zbyt dużą liczbę obowiązków i na niewspółmierne wynagrodzenia, szczególnie właśnie w momencie kiedy dochodzą nowe zadania. Zarząd utrzymuje, że średnia płac wynosi 5,8 tys. zł, jednak pragnę zauważyć, że średnia ta została wyliczona na podstawie wynagrodzeń nie tylko przeciętnych pracowników, ale też dyrektorów i członków zarządu, prezesa etc. W rzeczywistości zgodnie z doniesieniami medialnymi szeregowi pracownicy i pracownice zarabiają mniej więcej 3 tys. zł na rękę. Jednak zarząd ZUS nie chce udzielić oficjalnej informacji swoim pracownikom na temat średniego wynagrodzenia. Dlatego pytam: Ile wynosi średnie wynagrodzenie szeregowych pracowników i pracownic ZUS zatrudnionych na merytorycznych stanowiskach (Dzwonek), w domyśle: bez kadry kierowniczej? Czy za pomysłem obarczenia pracowników i pracownic ZUS kolejnymi obowiązkami pójdą należne im podwyżki płac, tak by wynagrodzenia były współmierne do ilości wykonywanej pracy? Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Wysoka Izbo! Pani minister, ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy systemu teleinformatycznego. W uzasadnieniu projektu raz jest mowa o tym, że ten system już jest, w innym miejscu jest mowa o tym, że ten system dopiero będzie. Czy to będzie wykonawca, który już wykonuje jakieś usługi na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy to zadanie zostanie powierzone komuś w tzw. trybie z wolnej ręki, bez żadnego trybu konkurencyjnego?

Pani minister, dużo mówicie o ludziach, ale to jest chyba pierwszy rząd, który tak lekką ręką zwalnia 11 tys. ludzi. Naprawdę podziwiam dobry nastrój pani minister, która jest na tej sali. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Pani Minister! Wysoka Izbo! W tysiącach gmin trzeba było przygotować lokale, sprzęt komputerowy, przeszkolić oraz zatrudnić personel. Sam system informatyczny kosztował dziesiątki milionów złotych. Dzisiaj rząd w ramach odciążania tych samych samorządów pozostawia je z całą infrastrukturą oraz z personelem na lodzie. Kto tym ludziom, pani minister, zapewni pracę? Dlaczego dobijacie finansowo samorządy? Chciałem też zapytać o koszty, jakie poniesie ZUS w związku z przejęciem obowiązków samorządów w tym zakresie. Trzy konkretne pytania: Jakie rząd planuje rekompensaty dla gmin i dla zwalnianych pracowników? Jakie środki przewidziano dla ZUS w zakresie wynagrodzeń i podwyżki płac dla pracowników, którzy będą mieli wykonywać dodatkowe zadania? Ja bym prosił, pani minister, aby pani nad tym się głęboko zastanowiła, bo już raz pani odpowiedziała, że żadne. Bardzo proszę, pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Wiele krytycznych słów płynie ze strony samorządów, ale do zmiany negatywnie też odniosło się Rządowe Centrum Legislacji, które wyraźnie uznaje, iż może zostać tutaj naruszona zasada równości. Dotyczy to nie tylko wymogu składania wniosków w formie elektronicznej na profile PUE ZUS, ale także doręczania decyzji administracyjnych i innych pism. Brak umiejętności cyfrowych czy odpowiednich środków technicznych, a nawet transportowych może nawet pozbawić rodziny prawa do świadczeń wychowawczych, a więc nie będzie to już program, jak pani minister mówiła, powszechny. Należy podkreślić, że ośrodki pomocy społecznej są zlokalizowane w każdej, nawet najmniejszej gminie, w przeciwieństwie do oddziałów ZUS, do których trudniej dotrzeć. Chciałabym, żeby ministerstwo się odniosło do sprawy wymuszania posiadania profilu PUE ZUS. Czy nie budzi to wątpliwości konstytucyjnych według ministerstwa? Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Główne zmiany w omawianej nowelizacji ustawy to obsługa i wypłata świadczeń 500+ wyłącznie przez ZUS, a nie ośrodki pomocy społecznej, jak dotychczas, wnioski będą składane wyłącznie przez Internet, a środki będą przekazywane wyłącznie bezgotówkowo. Jak zatem będą obsługiwani beneficjenci programu, którzy niestety nie mają możliwości złożenia wniosku on line lub nie posiadają konta w banku? Samorządy poniosły spore koszty organizacyjne i wdrożeniowe związane z realizacją programu. Zatrudniono ponad 12 tys. dodatkowych osób do obsługi programu w całej Polsce, po to aby środki efektywnie trafiały do uprawnionych odbiorców. Dlaczego? Co z pracownikami w ośrodkach pomocy społecznej? Czy ministerstwo planuje udzielić pomocy pracownikom, którzy stracą pracę wskutek przeniesienia realizacji programu (Dzwonek) do ZUS? I co z pracownikami ZUS, którzy już teraz są bardzo obciążeni i obawiają się, że kolejne obowiązki zablokują system? Pani poseł Małgorzata Pępek. Bardzo proszę, pan poseł Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Pani Minister! Wysoka Izbo! Padają na tej sali bardzo istotne pytania dotyczące świadczenia 500+. Pozwolę sobie po części je także powtórzyć, żeby głośno wybrzmiały na tej sali, a wynikają one z rozmów zarówno ze stroną samorządową, jak i z ośrodkami pomocy społecznej czy samymi rodzicami. Pytanie dotyczące składania wniosków tylko elektronicznie. Czy to nie doprowadzi do wykluczenia części beneficjentów, którzy nie mają dostępu do Internetu bądź też mają problem z jego obsługą? Mam też pytanie dotyczące pracowników ośrodków pomocy społecznej. Co z nimi? Co z tymi, którzy zostali zatrudnieni do wykonywania zadań związanych z programem 500+? Prawdopodobnie w związku z tym nastąpi redukcja etatów. I dlaczego zrzucane są na samorządy koszty związane z redukcją etatów i ewentualnych odpraw? Bardzo proszę, pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Pani Minister! Wysoka Izbo! Ta ustawa miała być dla ludzi, a tymczasem wprowadziła ogromny niepokój. Boją się pracownicy, że stracą pracę, boją się osoby mniej sprawne technologicznie, że sobie z tym nie poradzą, pytają mnie, czy dostaną pieniądze, czy w ogóle ich nie dostaną. Boją się wszyscy, że krótkie vacatio legis spowoduje, że sobie nie poradzicie z technologią i że będzie tak wielki bałagan, że będą opóźnienia w wypłatach. Zatem pytam o jedną, najważniejszą kwestię, bo o najsłabszych. Ile w tej chwili jest osób, które nie mają konta i które otrzymują pieniądze, że tak powiem, do ręki? Czy mogę prosić o odpowiedź w liczbach bezwzględnych, nie procentowych, jaka to jest grupa?

Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Państwa rozwiązanie de facto utrudnia wychowywanie dzieci. Proszę spojrzeć, iść naprawdę szczególnie do tych małych, biednych gmin. W Polsce 5 mln osób, według najnowszych badań, nie korzysta z Internetu i z komputera. Przecież to gmina, której chcecie odebrać wypłacanie świadczenia 500+, jest najbliżej obywatela, każdego obywatela. To nie są argumenty, które mają pomóc rodzinom, one zwyczajnie utrudnią, nie tylko poprzez fakt niewypłacania w formie gotówki, ale również poprzez to, że tych kilka tysięcy czy może kilkanaście tysięcy wyszkolonych, znakomicie wyszkolonych pracowników w samorządach straci pracę. Pracownicy ZUS-u nie są jeszcze do tego przygotowani.

Bardzo proszę, pani poseł Anna Wojciechowska, Koalicja Obywatelska. Pani Minister! Wysoka Izbo! Już program „Dobry start”, którego obsługą od 1 lipca zajmuje się ZUS, pokazał, że system elektronicznego składania wniosków nie działa sprawnie i stwarza problemy. Pracownikom ZUS zostały przydzielone dodatkowe zadania, które wykraczały poza normę ich czasu pracy. Wnioskodawcy nadal zwracają się o pomoc do punktów obsługujących jeszcze program „Rodzina 500+” w swoich gminach. Ale i tych może wkrótce zabraknąć. Beneficjenci świadczeń pozostaną bez profesjonalnej pomocy, natomiast pracownicy zatrudnieni dotychczas do obsługi programu „Rodzina 500+” mają uzasadnione obawy, że zostaną bez pracy. Należy również zauważyć, że organy realizujące przepisy ustawy mają narzędzia do tego, by kontrolować, czy świadczenia wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem, o czym mówiły moje poprzedniczki. W związku z powyższym zwracam się do pani minister (Dzwonek) z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania: Ile osób w związku z obsługą programu 500+ jest zatrudnionych obecnie w kraju? Czy w związku z przeniesieniem zadań związanych z jego realizacją powstaną tam nowe miejsca pracy? Co stanie się z pracownikami obsługującymi do tej pory program? Bardzo proszę, pani poseł Barbara Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister!

Od kwietnia 2016 r. 500+ jest wypłacane. Czegoś takiego wcześniej nie było. Za tym programem, oprócz tego, że od razu popłynęły pieniądze do budżetów samorządów, popłynęły też bardzo duże pieniądze na jego obsługę, o czym zresztą pani minister mówiła, a tutaj padają słowa, że gminy nic nie otrzymały.

Bo to też była dodatkowa pomoc. Z dzisiejszej debaty, która jest jak zwykle krytyką, krzykiem itd., wynika (Dzwonek) jedno dobro. Państwo zwróciliście uwagę na to, że są pracownicy ZUS-u, którzy bardzo ciężko pracują. Przez lata rządów Platformy Obywatelskiej - PSL tylko mówiliście źle o ZUS-ie, a nawet padały tu słowa: należy tych darmozjadów zwolnić, pieniądze wrócą do budżetu państwa. Faktycznie pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bardzo źle zarabiają. Te podwyżki są, ale one są wciąż małe, dlatego taki apel.

Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Przez ostatnie 6 lat nie słyszałam z tej trybuny żadnego apelu o wynagrodzenia dla pracowników ZUS. Pani poseł, pani przez 6 lat o tym nie mówiła. A teraz do rzeczy. Po pierwsze, pokazaliśmy, że na 11 tys. pracowników może być zwolnionych ok. 8 tys. Chciałam zapytać panią minister: Czy pani napisze im list pożegnalny, tym zwalnianym pracownikom? Czy pani napisze list pożegnalny do samorządów, które będą traciły pieniądze? Czy pani wie, jak wygląda wdrażanie programu elektronicznego, możliwości przesyłania i ile dostaną podwyżki pracownicy ZUS-u? I czy to jest pierwszy etap (Dzwonek), bo są zapowiedzi, że ZUS będzie przekazywał również świadczenia emerytalno-rentowe dla nowych emerytów w formie elektronicznej? Kiedy i czy państwo w tym zakresie poczynili jakieś starania? I ostatnia sprawa dotycząca ratingu samorządów. Przecież państwo rządowo te samorządy pominęli. Rating samorządów - to znaczy, że żaden z samorządów, jeżeli utraci 500+ i był zadłużany, nie będzie mógł zaciągnąć żadnego kredytu, nawet w sytuacjach kiedy samorządowi potrzeba, bo będzie miał kategorię D, Co państwo wtedy zrobicie? Nie będzie możliwości emisji obligacji komunalnych, nie będzie możliwości zaciągnięcia kredytu. Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Pani Minister! Gratuluję pomysłu. Projekt dotyczy powierzenia obsługi programu 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, zmiany formy składania wniosków tylko na elektroniczne i możliwości wypłaty środków jedynie na konta bankowe. Co z ludźmi, którzy nie mają dostępu do Internetu? Co z rodzinami, które nie mają konta bankowego? Wypadną z systemu? Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Do tej pory dobrze funkcjonował system obsługi 500+. Robiły to samorządy, stworzyły miejsca pracy, zakupiły sprzęt, wyposażyły, przeszkoliły osoby. Trzeba to wszystko wywrócić do góry nogami, żeby utrudnić życie ludziom i samorządom. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Bożena Żelazowska, Koalicja Polska. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Moje pytanie do pani minister to pytanie, które zadają samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast: Dlaczego zabieracie państwo środki finansowe i zadania samorządom, które dobrze te zadania realizują, które są bliżej swoich mieszkańców, które znają potrzeby polskich rodzin, rodzin, które tam właśnie mieszkają? Co mają zrobić osoby, które są świetnie przygotowane, które pracują i obsługują te programy? Gdzie oni pójdą do pracy? To też przedstawiciele polskich rodzin. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Szczęść Boże! Dobry wieczór.

Zmieńcie, proszę, tytuł swojej ustawy i nie mówcie więcej o tym, że pomagacie dzieciom. kiedy pod pretekstem walki z pandemią niszczycie polską rodzinę, nie mówiąc oczywiście o przedsiębiorczości. Bardzo proszę, pani poseł Daria Gosek-Popiołek, Lewica. Pani Minister!

Ono padło nie tylko dzisiaj. Od tygodni sami pracownicy, związki zawodowe, posłowie i posłanki, do których, tak jak do mnie, ci pracownicy się zwracają, zadają to pytanie. A pani minister ucieka od odpowiedzi, nie daje żadnych konkretów, nie ma żadnych pomysłów. Jak rozumiem, los tych kilku tysięcy osób, które być może stracą pracę, jest wam zupełnie obojętny. Zwracam uwagę na to, że osoby te przez lata zdobywały doświadczenie, uzupełniały swoją wiedzę, doskonale znają ten program, a ponieważ są pracownikami gminnymi, bardzo często mają naprawdę bliskie relacje, są w stanie pomóc w sytuacjach, w których inne osoby potrzebują pomocy. Nagle mówi im się (Dzwonek), że muszą znaleźć pracę w sytuacji kryzysu. Pani poseł Katarzyna Kotula, Lewica. Wysoka Izbo! To dobry krok w kierunku informatyzacji i cyfryzacji, co oczywiście zawsze się chwali, niestety rzeczywistość wciąż jest brutalna. Statystyki pokazują, że ponad 4,5 mln Polek i Polaków nigdy nie korzystało z Internetu. Kiedy przyglądamy się temu bliżej, to widzimy, że najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe są gospodarstwa domowe o najniższych dochodach. Aż 945 tys. osób z niepełnosprawnościami, czyli 36%, nigdy nie korzystało z Internetu. Chciałabym w związku z tym zapytać. W okresie zasiłkowym 2019-2020 31,5% wszystkich wniosków zostało złożonych drogą tradycyjną, czyli drogą papierową. Wiemy, że z tej formy wystąpienia o świadczenie dla dzieci w dużej mierze korzystali odbiorcy wrażliwi, czyli rodziny ubogie, z mniejszych [[Dzwonek]] ośrodków miejskich lub ze wsi, a także rodziny wykluczone cyfrowo, czyli te, o których przed chwilą mówiłam. To właśnie te rodziny szczególnie narażone na skutki wykluczenia, a więc wymagające wsparcia, mogą stać się ofiarami ograniczonej dostępności i stworzonych barier.

Zaczynam mieć wrażenie, że pomimo że 500+ to dobry program, ta nowelizacja może być niestety sposobem na wylanie dziecka z kąpielą. Pani poseł Agnieszka Hanajczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Minister! Wysoka Izbo! Sztandarowy projekt 500+ jest faktem. Państwo często o tym mówicie i nikt z tym nie dyskutuje.

Ale czy państwo jesteście świadomi tego, jak wielka praca została wykonana? Przyznam szczerze, że dzisiaj byłam trochę, a może dość mocno, zażenowana, kiedy pani minister, reprezentując, niejako będąc szefową ministerstwa empatii, wrażliwości, nawet się nie zająknęła na temat ludzi, którzy będą szukać pracy, może jej nie znajdą, może będą bezrobotni. Nie zająknęła się pani minister. Zwyczajne słowo: dziękuję. A z drugiej strony, pani minister, czy pani jest świadoma, że.

Nie wierzę w to, że pani minister o tym nie wie. Pani poseł Magdalena Łośko, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nawet ZUS nie rozumie zmian w obsłudze programu 500+. Propozycje rządu mogą utrudniać wypłatę świadczeń, zmieniają coś, co dobrze funkcjonowało. Nie jest jasne, dlaczego rząd podjął decyzję o przeniesieniu obsługi 500+ do ZUS. MOPS-ów jest przecież ponad osiem razy więcej niż oddziałów ZUS-u. MOPS-y zostały specjalnie przygotowane i wyszkolone do obsługi programu. Trudno w to wszystko uwierzyć. Czemu rząd chce rozbijać powstałą strukturę, obciążać kolejnymi obowiązkami Zakład Ubezpieczeń Społecznych, odbierając zadania już wcześniej przeszkolonym pracownikom i narażając ich na możliwe zwolnienia? Mam zatem pytanie, pani minister: Czy ministerstwo planuje zaangażować zewnętrzne podmioty do obsługi programu? Nie muszę chyba wspominać, że będzie to rażąca niegospodarność i arogancja wobec ewentualnie zwolnionych osób. Dziękuję, pani poseł. Ostatnie pytanie zadaje pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! To nie jest dobry projekt. Ten projekt nie jest dobry przynajmniej z kilku powodów.

To uderza w samorząd. Proszę państwa, samorząd w tym zakresie wykonał gigantyczną pracę i teraz kilka tysięcy osób, które były zatrudnione w instytucjach samorządowych, może tę pracę stracić. W wielu miejscach, w małych miejscowościach, jeśli chodzi o pracę, znaleźć ją będzie bardzo, bardzo trudno. Samorząd miał już duże doświadczenia. Kolejny element: korzystający.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej panią minister Barbarę Sochę o odpowiedź na pytania.

Wysoka Izbo! Postaram się pokrótce odpowiedzieć na większość państwa trosk i wątpliwości związanych z tym projektem. Po pierwsze, ten projekt nie wprowadza żadnych zmian związanych z uprawnieniami rodzin i ich dostępem do świadczenia 500+.

Szanowni Państwo! Ja cierpliwie słuchałam z wielką uwagą państwa wystąpień i bardzo bym prosiła, żeby nie przerywać. Głównym celem, jak było mówione, jak pani minister przedstawiała w swoim wystąpieniu, jest wprowadzenie pewnych znaczących oszczędności związanych z obsługą tego świadczenia.

Jeśli chodzi o rodziny i wielokrotnie podnoszone wykluczenie cyfrowe i społeczne. Szanowni państwo, to nie jest pierwszy raz, kiedy zmierzamy w stronę cyfryzacji, automatyzacji usług.

W tej chwili jesteśmy w trakcie, a właściwie już można powiedzieć, że nabór wniosków w programie 300+, który był pewnego rodzaju pilotowym programem w stosunku do tej zmiany, praktycznie dobiega końca, dlatego że na 4200 tys. uprawnionych dzieci do świadczenia 300+ już mamy złożonych 4200 tys. wniosków. To jest o 250 tys. więcej wniosków, niż mieliśmy w zeszłym roku o tej samej porze, co oznacza - i można z tego wysnuć wnioski - że jest to łatwiejsze do wdrożenia i wygodniejsze dla rodziców. Co więcej, nie odbieramy żadnych sygnałów od rodziców, którzy narzekaliby na tę zmianę i mieli jakiekolwiek problemy z ubieganiem się o świadczenie 300+. Jeśli chodzi o sytuację samorządów związaną z tą zmianą.

Jeśli chodzi o sytuację związaną z pracownikami w samorządach. Szanowni państwo, pracownicy samorządowi, którzy w związku z tą zmianą rzeczywiście w iluś przypadkach może się zdarzyć, że stracą pracę, będą oczywiście mieli odprawy zgodne z Kodeksem pracy.

Co do sytuacji cudzoziemców i związanej z tą obsługą koordynacji świadczeń, nadal to zadanie jest wykonywane przez wojewodów i środki na to są utrzymywane. W tej sytuacji to się nie zmieni. Na obsługę tego świadczenia środki były przeznaczane przez rząd od samego początku. Początkowo dodatkowe 60 mln zł na przygotowania dla samorządów do wypłaty tych świadczeń.

Dzisiaj tą zmianą planujemy przenieść obsługę świadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Mianowicie fakty są takie. Z tych ponad 4 mln wniosków, o których mówiłam, czyli ogromnej większości już osób uprawnionych, 99% wniosków jest obsługiwana przez automat. Nie jest tu wymagana ingerencja żadnego pracownika. To nie jest tak, że wszyscy pracownicy ZUS w całej Polsce zajmują się obsługą programu „Dobry start”, tak samo jak nie będą zajmowali się obsługą programu 500+. Przewidywane jest między 50 a 70 etatów - tyle osób będzie się zajmowało obsługą programu „Rodzina 500+” Właśnie na tym polega automatyzacja.

2% wypłat do tej pory odbywało się w formie gotówkowej, czyli ok. 90 tys. osób pobierało świadczenie w formie gotówkowej. Z różnych powodów te osoby wolały, żeby to świadczenie było wypłacane im w formie gotówkowej. Szanowni państwo, ci pracownicy są bardzo dobrze wyszkoleni i dobrze realizują swoje zadania.

Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 1530, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Marszałek Sejmu proponuje, aby Sejm, na podstawie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu, wyznaczył termin przedłożenia sprawozdania umożliwiający rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład (druk nr 1531) Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Sebastiana Skuzę o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład. Finanse samorządu terytorialnego to temat niezwykle istotny zarówno z punktu widzenia samych jednostek samorządu terytorialnego, jak i całego systemu finansów publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma już kilkanaście lat i wymaga dyskusji. Te rozmowy może nie są łatwe, ale są konstruktywne i wspólnie doszliśmy do wniosku, że pewne zmiany są jednak potrzebne. Oczywiście nie bez znaczenia dla finansów jednostek samorządu terytorialnego są rozwiązania proponowane w systemie podatkowym w ramach programu Polski Ład. Wiadomo, że historyczna obniżka podatków proponowana w Polskim Ładzie będzie miała wpływ na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też przedstawiamy projekt ustawy, w przypadku którego punktem wyjścia jest to, aby system finansów samorządu terytorialnego zapewnił większą stabilność i przewidywalność, jeśli chodzi o dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Podział ten uwzględniałby również poziom zamożności jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku rozwiązań doraźnych proponowane jest również uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego przez modyfikację reguł fiskalnych. Obecnie funkcjonują rozwiązania zabezpieczające jednostki samorządu terytorialnego przed nadmiernym zadłużeniem. Jest to zasada zrównoważenia budżetu bieżącego oraz ograniczenia możliwości zaciągania zobowiązań. Jest to oparte na tzw. indywidualnym wskaźniku zadłużenia każdej jednostki samorządu terytorialnego. W projekcie ustawy proponuje się czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego, czyli w średnim okresie czteroletnim w pewnych latach bieżący budżet jednostki samorządu terytorialnego mógłby być niezrównoważony, niemniej jednak musiałby być zrównoważony w całym okresie czteroletnim. W 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego umożliwione miałby również bilansowanie części bieżącej budżetu wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych. Co jeszcze w zakresie zmian dotyczących działań bieżących? Jeszcze jedną zmianą w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań byłaby propozycja zmiany możliwości wyboru przez jednostki samorządu terytorialnego okresu, na podstawie którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna. Jednostki samorządu terytorialnego miałyby tutaj przejściowo możliwość wyboru. Co zaproponowano w rozwiązaniach docelowych? Pierwsza rzecz: na wniosek samych jednostek samorządu terytorialnego z limitu zadłużenia zmniejszono próg udziału środków Unii Europejskiej w finansowaniu programów. To znaczy, że obecnie jeżeli jakiś program jest finansowany powyżej 60% ze środków unijnych, nie jest on uwzględniany w indywidualnym wskaźniku zadłużenia. Na wniosek samych jednostek samorządu terytorialnego ten procent został obniżony do 50%. Jakie z kolei zmiany docelowe proponuje projekt ustawy? Po pierwsze stabilizacja i przewidywalność dochodów. Od przyszłego roku projekt przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego udziały z tytułu PIT i CIT otrzymywałyby w 1/12 przewidywanych środków na dany rok budżetowy, czyli podobnie jak w przypadku subwencji miałyby stały regularny dochód w znanej wysokości - 1/12. Następnym rozwiązaniem - jak myślę - istotnym dla jednostek samorządu terytorialnego jest kwestia oparcia mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego na bieżących wpływach z tytułu PIT i CIT. W obecnym systemie korekcyjno-wyrównawczym występuje dwuletnie przesunięcie pomiędzy rokiem, na podstawie którego oblicza się wpłaty, a rokiem, w którym te wpłaty są realizowane. Chodzi o kwestię janosikowego, że np. wypłacane byłoby ono w roku n w trakcie dekoniunktury, a naliczenie byłoby z okresu n-2, czyli koniunktury. Projekt przewiduje również rozwiązanie proinwestycyjne polegające na wprowadzeniu nowej części subwencji ogólnej, tzw. części rozwojowej. I tu muszę podkreślić, że część rozwojowa nie będzie traciła przymiotu subwencji i będzie mogła być wykorzystana na wszelkie zadania jednostek samorządu terytorialnego i będzie traktowana w budżetach jednostek samorządu terytorialnego jako dochód bieżący, czyli będzie można nią finansować również wydatki bieżące. Ona ma taką nazwę: rozwojowa, bo wprowadzone są pewne mechanizmy zachęty, żeby jednak jednostki samorządu terytorialnego inwestowały jak najwięcej tych środków. Ta część rozwojowa subwencji składałaby się z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej. Kwota podstawowa przysługiwałaby każdej jednostce samorządu terytorialnego, a jej podział następowałby proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego z określeniem minimalnych i maksymalnych kwot. Premia aktywizująca przysługiwałaby takiej jednostce samorządu terytorialnego, która w przeliczeniu na jednego mieszkańca te wydatki inwestycyjne miałaby powyżej przeciętnej. Premiera inwestycyjna z kolei przysługiwałaby takim jednostkom samorządu terytorialnego, w których wskaźnik wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca po prostu będzie rósł proporcjonalnie do wydatków majątkowych uprawnionych odpowiednio jednostek samorządu terytorialnego, czyli procent, przyrost procentowy będzie wyższy niż średnia. Z tą częścią subwencji prorozwojowej jest powiązany pewien mechanizm zabezpieczający jednostki samorządu terytorialnego przed spadkami dochodów z tytułu CIT i PIT. Mianowicie projekt ustawy przewiduje mechanizm, że w danym roku budżetowym, począwszy od roku 2023, dochody z tytułu udziału w CIT i w PIT nie będą mogły być niższe niż kwota referencyjna, którą jednostki samorządu terytorialnego same wyprognozowały w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022, jeszcze przed skutkami Polskiego Ładu, czyli można powiedzieć, że na starych zasadach. Ta kwota byłaby waloryzowana nominalnym wzrostem PKB, czyli uwzględniającym wzrost gospodarczy i inflację.

Czyli jest np. luka na poziomie 6 mld zł, subwencja prorozwojowa musi wynieść 6 mld zł. Gdyby tej luki nie było, to wtedy rząd jest zobligowany ustawą zabezpieczyć kwotę 3 mld zł subwencji inwestycyjnej również waloryzowaną wzrostem nominalnego PKB. Czyli jednostki samorządu terytorialnego zyskiwałyby zapewnienie pewnej kwoty z tytułu udziału w podatku CIT i PIT. Pojawiały się tutaj głosy, że lepszym rozwiązaniem dla jednostek samorządu terytorialnego byłoby zwiększenie udziałów w podatkach dochodowych, niemniej jednak zwracam uwagę, że to nie działałoby np. w małych i średnich gminach. Z tego względu, że zakładam, że wszyscy bądź prawie wszyscy popierają rozwiązanie klina podatkowego, czyli zwiększenia kwoty wolnej od podatku i wtedy w gminach, w których jest dużo emerytów o niskich dochodach, w których ludzie pracują na minimalnych wynagrodzeniach lub trochę wyższych, zwiększenie udziału procentowego nic by nie dało. Na zakończenie chciałbym jeszcze nawiązać do wystąpienia pani minister Barbary Sochy i jednoznacznie zapewnić, że jeżeli chodzi o kwestię dotacji na działania bieżące, czyli tutaj z tytułu 500+, to te środki nie są uwzględniane we wzorze na indywidualny wskaźnik zadłużenia w art. 242.

Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za uwagę. Pozostaję do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość do projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład (druk nr 1531) Tak by się mogło nawet wydawać. Tylko oczywiście zapewnienia o tym, że rząd przygotowuje rozwiązania osłonowe dla gmin, teraz się materializują i faktycznie można powiedzieć, że samorządy wręcz zyskują na Polskim Ładzie i to kwoty - powiedziałbym - niebotyczne.

Tutaj zresztą wielokrotnie o tym z panem ministrem rozmawialiśmy, że w momencie, w którym będzie procedowany Polski Ład, powinna być też procedowana ustawa o kompensacji utraconych przychodów przez gminy. Ale powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że ta kompensacja będzie tak hojna.

Można się o tym przekonać, analizując sposób podziału tej kwoty na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Moją gminę, w której kiedyś byłem wójtem, mogę podać jako przykład.

Ale do tego jeszcze są kwoty stabilizujące, subwencja wyrównawcza, subwencja rozwojowa i - co jest ważne - wszystkie te subwencje są dochodami bieżącymi.

Ale też warto wspomnieć, że samorządy dzięki znakomitej polityce gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości zyskały też ogromne udziały i ogromne wpływy. Bez względu na to, jak byśmy.

Sama Warszawa, która najbardziej tutaj płacze, bo wydaje pieniądze też nie wiadomo jak. Akurat w Warszawie wzrost tych dochodów wyniósł 47%. I pewnie prezydent Trzaskowski będzie mówił, że jest biedny z tego powodu jeszcze, nadal biedny.

Ja tylko wspomnę 13 mld zł z poszczególnych transzy COVID-owych czy ponad 100 mld zł teraz w rządowym funduszu inwestycji strategicznych. Takich pieniędzy samorządy nie miały i pewnie w historii daleko by sięgać, żeby tak było.

Proszę, pan poseł Jacek Protas, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawiam nasze stanowisko dotyczące projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład. Na początku chcę się zgodzić z tezą zawartą w uzasadnieniu projektu, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 r. wymaga gruntownych zmian, a właściwie trzeba ją napisać od nowa, bowiem nie uwzględnia nowej sytuacji oraz nowych zadań, jakie przez 17 lat zostały powierzone samorządom.

W międzyczasie natomiast rząd zaproponował, a większość sejmowa uchwaliła, szereg zmian ustawowych destabilizujących finanse samorządu.

Tego pan chyba nie zazdrości, panie pośle. Dodatkowo samorządy obarczane były, i są, większymi wydatkami na utrzymanie oświaty. W 2014 r. subwencja oświatowa pokrywała 66% wydatków na utrzymanie szkół i placówek, w 2019 r. już tylko 60%. Te ubytki w dochodach stoją w sprzeczności z zapisaną w art. 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą adekwatności zasilania finansowego do zakresu zadań. Tymczasem zgodnie z rządowymi danymi zmiany podatkowe w Polskim Ładzie mają skutkować spadkiem dochodów jednostek samorządu terytorialnego o dalsze 12 mld zł rocznie. Natomiast propozycje zrekompensowania tych ubytków zawarte w omawianym przez nas dzisiaj projekcie ustawy są dalece niewystarczające. Stosowne projekty dotyczące tych rekompensat były składane przez nas w Sejmie i uchwalone przez Senat. Niestety trafiły do zamrażarki pani marszałek.

Po trzecie, komplikują i tak już nieprosty system finansowania zadań realizowanych przez samorządy. Samorządy oczekują natomiast stabilizacji dochodów własnych. Dla parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, ale też dla samorządów projekt ustawy w tym kształcie jest nie do przyjęcia. Nie został też uzgodniony przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, panie pośle. Jego przyjęcie skutkowałoby dalszym drastycznym obniżeniem dochodów samorządów terytorialnych, a co za tym idzie - zahamowaniem inwestycji oraz pogorszeniem jakości usług publicznych. Szkoły, przedszkola, żłobki, pomoc społeczna, służba zdrowia, transport publiczny, jakość dróg i chodników - na to wszystko łożą przecież samorządy. Dlatego na jutrzejszym posiedzeniu połączonych komisji Koalicja Obywatelska po konsultacjach z przedstawicielami samorządów złoży poprawki, które pozwolą zrekompensować jednostkom samorządu terytorialnego dotychczasowe straty i zapewnią im stosowny do zadań poziom dochodów poprzez procentowy wzrost udziałów w podatkach PIT i CIT. Zakładając dobrą wolę rządu i większości sejmowej, liczymy na poparcie naszych merytorycznych propozycji.

Bardzo proszę, pani poseł Monika Falej, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Lewica mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład. Polski Ład miał być obietnicą stabilnej i długofalowej strategii wychodzenia z kryzysu po pandemii. A czym jest? Niespełna 4 miesiące przed nowym rokiem Polki i Polacy nie wiedzą, jakie zapłacą podatki, a polskie samorządy, jakie poniosą koszty.

Szereg rozwiązań budzi kontrowersje. Co chwila dowiadujemy się o nowym propozycjach, które szybko i bez przemyślenia dorzucane są do karuzeli obietnic, choćby w nowej wersji, gdzie pojawił się nowy podatek. Ministerstwo Aktywów Państwowych alarmuje, że nawet ono nie miało możliwości skonsultowania tego projektu, a skutki mogą być opłakane, zwłaszcza dla spółek państwowych. W Polskim Ładzie co chwila coś się zmienia, wszystko oprócz jednego - od początku wiadomo, kto będzie główną ofiarą, a żadne kolejne rozwiązania tego nie zmieniają. To samorządy. Polski Ład ewidentnie ma uderzyć w polskie samorządy i ich niezależność. Stracimy na tym wszyscy, ponieważ proponowane przez premiera Morawieckiego zmiany w podatkach to mniej pieniędzy na szkoły, żłobki, mieszkania komunalne, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, to wyższe ceny biletów i cięcia w inwestycjach infrastrukturalnych. Zmiany w podatkach PIT i CIT znacząco uszczuplają budżety lokalne i to wszyscy wiedzą. Chyba wszyscy poza twórcami Polskiego Ładu. Dziś przedstawiacie projekt próbujący naprawić konsekwencje swoich planów. Rozwiązania dziś proponowane nie zrekompensują jednak strat.

Będą cięcia nie tylko inwestycji, ale także wydatków bieżących w samorządach, to oczywiste. Przedstawiacie państwo rozwiązania, które sami zainteresowani negatywnie zaopiniowali podczas konsultacji w komisji wspólnej rządu i samorządu.

Tak się nie stanowi prawa. Wiecie doskonale, że rozwiązania dziś proponowane nie są ofertą dla samorządów, a karą. A więc albo nie potraficie liczyć, albo macie jakiś inny cel - zmienić kompletnie model finansowania samorządów, by je od siebie uzależnić i nagradzać swoich. Lewica będzie za każdymi prostymi i bezpiecznymi rozwiązaniami dla samorządu. Chcemy, aby samorządy nie straciły ani złotówki, by miały zagwarantowane pełne wyrównanie strat dla samorządów na stałe, a nie jednorazowo. Dlatego Lewica złoży do druku, ale akurat nr 1532, czyli dużej ustawy podatkowej, poprawki, które dotyczyć będą wprowadzenia mechanizmu, dzięki któremu jednostki samorządu terytorialnego wyszłyby na samej reformie podatkowej co najmniej w tym momencie na zero. Bez takiego mechanizmu ustawa podatkowa będzie siłą rzeczy oznaczała gorsze samorządowe usługi publiczne.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Urszula Nowogórska, Koalicja Polska. Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicji Polskiej - PSL, Unii Europejskich Demokratów, Konserwatystów mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu parlamentarnego w odniesieniu do projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład, zawartego w druku sejmowym nr 1531. W uzasadnieniu przedłożenia czytamy, że podstawowym celem projektu jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego optymalnych warunków prowadzenia przez nie gospodarki finansowej w związku z programem Polski Ład. Zapis brzmi dumnie, pod warunkiem że wszystkie samorządy będą miały możliwość równego rozwoju, a podział środków będzie pobudzał ich aktywność i nie będzie uznaniowy. Szanowna Pani Marszałek! Samorządność lokalna jest wielkim osiągnięciem demokratycznej transformacji Polski, budząc przez trzy dekady poczucie zaufania Polaków i podkreślając fundamentalną zasadę i rolę samorządów w ustroju terytorialnym kraju. Wola polityczna wzmocnienia wspólnot lokalnych gmin, powiatów, miast i województw była źródłem siły całego państwa i wszyscy byśmy chcieli, żeby tak dalej pozostało. Po-covid-owa codzienna rzeczywistość pokazuje ogromną niepewność, przed jaką stanęły samorządy. Przykładem takiego stanu rzeczy i nieprzemyślanych czasem decyzji o zmianach granic administracyjnych miast i gmin może być gmina Dobrzeń Wielki, której przedstawiciele na wczorajszym posiedzeniu komisji samorządu terytorialnego podkreślali i pokazywali problemy finansowe, z którymi gmina boryka się sama, ale te problemy finansowe w niedługiej przyszłości mogą dotyczyć również innych samorządów. Tę niepewność potęguje również brak zapewnienia ze strony państwa rekompensaty ubytków w dochodach bieżących jednostek samorządu, brak udziału samorządów w podatku VAT, brak systemu zwolnień z podatku VAT, brak zapewnienia udziału w PIT. W ostatnich latach dość powszechną zasadą stało się również dociążanie jednostek samorządu terytorialnego przez rząd nowymi zdaniami, z pominięciem mechanizmu rekompensaty finansowej. Samorządy pracy się nie boją. Są bardzo blisko ludzi, znają ich potrzeby, chcą realizować inwestycje, ale obawiają się, że nawet subwencja inwestycyjna określona w projekcie ustawy, która będzie dochodem majątkowym, nie uzupełni ubytków udziałów we wpływach z PIT, które są zmniejszeniem dochodów bieżących.

To spowodować może, że 1/3 jednostek samorządu terytorialnego utraci od razu płynność finansową, ich nadwyżka operacyjna netto spadnie poniżej zera. Znaczna część pozostałych samorządów będzie miała kłopoty ze sfinansowaniem wydatków bieżących związanych np. z oświatą, pomocą społeczną, utrzymaniem dróg. Nieliczni tylko utrzymają możliwość rozwoju. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne staje się wprowadzenie mechanizmu rekompensaty ubytku w dochodach bieżących przez np. zwolnienie z podatku VAT od towarów i usług nabywanych do realizacji przez samorządy projektów inwestycyjnych. To zresztą np. zostało mocno wyartykułowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, który jest największą regionalną korporacją samorządową w Polsce. Takie działania na pewno pobudziłyby inwestycyjną aktywność samorządową i bezpośrednio wpłynęłyby na utrzymanie bądź podwyższenie jakości życia mieszkańców. Poza tym wpisałoby się to w zasadę subsydiarności, decentralizacji i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w decydowaniu o wykonywaniu własnych zadań i kształtowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Wysoka Izbo! Po szczegółowej analizie projektu, która będzie miała miejsce jutro na posiedzeniu połączonych komisji, przedstawimy stosowne poprawki do tego projektu ustawy i określimy swoje stanowisko w tej sprawie.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Jest to jednak - mam wrażenie i myślę, że wszyscy mamy takie wrażenie - doraźne rozwiązanie wieloskładnikowe zamiast prostych, stabilnych, systemowych rozwiązań, których potrzebują samorządy. Słuchałem z uwagą pana posła Kowalczyka, którego wypowiedź zacytuję: Samorządy zyskują i dlatego robimy ustawę o kompensacji strat. Brawo. Brawo, gratuluję, wszyscy zyskują.

To jest coś dobrego i tego gratuluję.

Będzie to skutkować ograniczeniami działań inwestycyjnych oraz niższymi nakładami na realizację usług świadczonych mieszkańcom poszczególnych wspólnot samorządowych.

Te rekompensaty, jednorazowe subwencje, jak również nowe subwencje rozwojowe są dalece niewystarczające i nie załatają dziury budżetowej, jaka powstanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Rządowa polityka wobec samorządów i samorządowców jest w tym względzie taka, aby jak najbardziej uniesamodzielnić samorządy. Wyciągnięcie pieniędzy od przedsiębiorców, obywateli oraz wydrenowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwoli wam zapewne sfinansować Polski Ład, nasuwa się jednak pytanie, jakim kosztem i właściwie po co. W skali samorządowej efektem waszych działań będzie brak czystej wody w kranie, brak zajęć dodatkowych dla dzieci w szkołach, brak środków na remonty lokalnych dróg oraz zapewne podwyżki podatków i opłat lokalnych. I dlatego m.in. jako Konfederacja od samego początku zdecydowanie odrzucamy zaproponowane przez rząd rozwiązania i apelujemy, aby zaniechał on forsowania programu Polski Ład, na którym stracą samorządy, czyli pośrednio niestety stracimy my wszyscy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Oczywiście w trybie sprostowania, bo pan poseł Kamiński nie zrozumiał mojej wypowiedzi. Rzeczywiście ustawa kompensuje ubytki w podatku PIT i CIT dla samorządów. Natomiast po dokonaniu tej operacji, po dokonaniu kompensacji łącznie samorządy zyskują.

A więc rzeczywiście kompensacja jest z nawiązką, panie pośle.

Bardzo proszę, pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeżeli Polski Ład ma poprawić jakość życia, to nie powinien osłabiać samorządów, ale powinien je wzmacniać. Takie opinie dało się słyszeć podczas ostatniego forum ekonomicznego w Karpaczu i to są opinie, które wypowiadali doświadczeni samorządowcy, do których państwo również macie szacunek i często ten szacunek demonstrujecie. Jednak takich rozwiązań nie ma w tym projekcie. Próbujecie przykleić plaster na wielką ranę, którą zadajecie samorządom. Tradycyjnie walczycie z problemem, który sami stworzyliście.

Mówię o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na tej sali na ten temat rozmawialiśmy. Dlaczego nie można po prostu zwiększyć jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w PIT i w CIT proporcjonalnie do ich obniżki? Kolejny cytat: Projekt ustawy ze względu na jego pilny charakter nie został poddany procesowi uzgodnień oraz przedstawiony do zaopiniowania i konsultacji publicznych. Przecież Polski Ład ogłoszono 4 miesiące temu. Tak nie załatwia się kluczowych dla państwa spraw, a takimi sprawami są właśnie relacje pomiędzy władzami lokalnymi i centralnymi, jak również system podatkowy. Polska 2050, podobnie jak wszelkie inne siły polityczne działające w Polsce, docenia rolę samorządów lokalnych w naszym kraju. Będziemy przeciwni każdemu kolejnemu uszczupleniu budżetów tych samorządów. Uznajemy, że zgłaszanie tak głębokich zmian w systemie finansów publicznych na niecałe 4 miesiące przed terminem, od którego mają zacząć obowiązywać, jest po prostu niedopuszczalne. Oczywiście będziemy pracować nad treścią tej ustawy i zgłaszać poprawki, tak aby jak najmniej szkodziła ona polskim samorządom. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? To bardzo proszę. Zamykam listę.

Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na początku apeluję do szanownego pana posła, pana przewodniczącego Kowalczyka o to, aby nam ujawnił, która to gmina zyska ten milion więcej niż. Myślę, że wszyscy z przyjemnością tego wysłuchamy, a później sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest. Inni samorządowcy też wypytają tego włodarza, jak to dokładnie wygląda, jak to się dzieje, że on zyskał, a oni tracą. Czytam w uzasadnieniu projektu ustawy, że zaproponowane rozwiązania zapewniają dostosowanie do wyzwań, przed jakimi staną samorządy w konsekwencji wdrożenia ambitnych rozwiązań Polskiego Ładu.

Pozbawiacie tego de facto mieszkańców, bo to nie jakiś nie wiadomo jaki samorząd (Dzwonek), tylko mieszkańcy nie będą mieli na drogi, nie będą mieli na to, żeby zapewnić odpowiedni poziom edukacji itd. Pytanie jest takie: Kiedy wreszcie zrozumiecie, że potrzeby, które są najbliżej ludzi, czyli związane właśnie z edukacją, z zapewnieniem odpowiedniej jakości usług publicznych, które organizuje samorząd, to są te potrzeby, które trzeba finansować? Nie można zabierać tych środków. A wy konsekwentnie te środki zabieracie. Panie pośle, bardzo proszę o przestrzeganie czasu. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Wysoka Izbo! Z analizy finansowej projektów, które dotyczą Polskiego Ładu, wynika, że po wygaśnięciu tych 8 mld w roku 2022 w kolejnych latach samorządy stracą po 11 mld zł rocznie. Mam zatem pytanie: Jak to się ma do realizowanej od 1989 r. proeuropejskiej polityki Polski polegającej na rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej? Dlaczego Zjednoczona Prawica cofa Polskę w tej kwestii o prawie 30 lat?

To jedynie pogłębi różnice pomiędzy samorządami.

Ostatnia kwestia.

Bardzo proszę, pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. Pan poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo! Według oceny skutków regulacji przedstawionej przez rząd negatywne skutki tzw.

Muszę przyznać, że kiedy słuchałem pana przewodniczącego Kowalczyka i usłyszałem, że używa przykładu własnej gminy, żeby uzasadnić rzekomo nadzwyczajnie wysoką kompensatę, zacząłem się martwić. Jako żywo przypomniał mi się przykład Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. A więc pytanie, czy tak będzie i tym razem.

Mam nadzieję, że nie doprowadzicie państwo do tego, że samorząd stanie się fasadowy.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To nie jest tak, jak mówi pan premier, że samorządy są bogate i mają pieniądze na wszystko. W chwili obecnej wiele samorządów ma problem z dochodami bieżącymi, a co za tym idzie - z relacją, o której mowa właśnie w art. 242 w jego nowym brzmieniu, czyli z wyłączeniem wolnych środków bilansujących nierówność dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi.

Zmniejszone wpływy do tych budżetów z PIT-u, które są dochodami bieżącymi jednostek samorządu terytorialnego, to dodatkowy problem, dlatego że będzie wymuszone na samorządach ograniczanie wydatków bieżących, i to drastyczne w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zabraknie również pieniędzy na niezbędne wydatki (Dzwonek), np. na oświetlenie, utrzymanie infrastruktury, opiekę itd. Minuta minęła.

Wysoka Izbo! Tytuł ustawy to: ustawa o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład. O wsparciu? W ustach premiera, który na każdym kroku rzuca samorządom kłody pod nogi, to brzmi jak ironiczny żart. Od kilku lat dobijacie samorządy poprzez obciążanie ich bezsensownymi obowiązkami i kosztami związanymi z deformą edukacji. Polski Ład jest kolejnym krokiem w tę stronę. Na skutek proponowanych zmian podatkowych samorządy będą traciły miliardy złotych. Z obecnych szacunków wynika, że w ciągu najbliższej dekady ich dochody będą mniejsze o 132 mld zł. Teraz łaskawie proponujecie subwencję rozwojową, która rzekomo miałaby zniwelować częściowo te skutki i naprawić problem, który sami stworzyliście. Jak możemy mieć pewność, że to rzekome wsparcie nie będzie kroplą w morzu potrzeb? Czy tym razem znów będzie tak jak z funduszem inwestycji lokalnych (Dzwonek), który posłużył do tego, żeby karać regiony Polski, które głosują na opozycję? Wysoka Izbo! 1399, 1480, 1530, 1531, 1533, 1534 - numery druków z projektami ustaw, nad którymi dzisiaj procedowaliśmy. Każda z innej materii, ale mają jeden wspólny mianownik - wszystkie ograniczają wpływy samorządów, wszystkie zabierają pieniądze samorządom. Panowie i panie z PiS-u, przestańcie okradać samorządy, przecież samorządy nie mają możliwości zakombinowania pieniędzy. Przecież wójt czy burmistrz nie przepiszą działek na starostę czy na marszałka, jak robią to niektórzy posłowie z waszej strony. Wójt czy burmistrz nie zamienią się majątkiem z innym wójtem czy burmistrzem, żeby nie zapłacić waszych podatków. Panowie i panie, sprawy najważniejsze, woda, którą dostajecie w waszych domach, w waszych miastach. Tę wodę doprowadzają wam wójt i burmistrz, nie minister klimatu, on tylko weźmie za to swoją działkę. On tylko chce na nich położyć łapę. Pani poseł Katarzyna Lubnauer. Panie Marszałku! Od początku było wiadomo, że Nowy Polski Ład jest wprowadzany kosztem dwóch podmiotów: aktywnych, przedsiębiorczych Polaków i samorządów. Okradacie samorządy. Jako matematyk powiem jasno: jeżeli komuś się zabiera rocznie od 12 do 15 mld zł, a oddaje zamiast tego w pierwszym roku 8 mld zł, a w kolejnych latach - od 3 do 4 mld zł, to jest on okradany. Oznacza to, że jeżeli oddacie tę jedną trzecią, to będzie to znaczne uszczuplenie środków. On wyglądałby jak komputer, a służyłby jak cep. I ta ustawa dokładnie tak wygląda. Jeżeli spojrzymy na to, że Unia Metropolii Polskich i samorządy nie chcą zaakceptować waszej zmiany. Ta zmiana po prostu nie jest korzystna. Pani poseł Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wydaliście wyrok na samorządy, na całe społeczności lokalne, a ten wasz Polski Ład to jest taki finansowy, już naprawdę ostateczny wyrok.

A jednorazowa subwencja to będzie ok. 25%, czyli ci mieszkańcy cały czas tracą 75%. To jest 37 przychodni, 20 szkół z oddziałami przedszkolnymi, 125 żłobków, w których miejsce znalazłoby 18 tys. dzieci. Za co jest ta kara?

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nowy Ład uderza w ludzi najbardziej przedsiębiorczych, tych, którzy prowadzą własne firmy i biorą odpowiedzialność za prowadzenie swoich biznesów, i uderza w samorządy. Moje miasto Szczecin tylko w przyszłym roku według wstępnych szacunków straci ok. 80 mln zł. Za te pieniądze można by wybudować szkołę, cztery przedszkola, wyremontować drogi albo kupić 30 nowych elektrycznych autobusów. Nie będzie można tego zrobić, bo wy wprowadzacie rozwiązania, które dla samorządów są po prostu niekorzystne. Jedna kwestia, która jest zasadnicza: jeżeli tam są mechanizmy, które później macie wdrażać, które będą decydować o tym, ile pieniędzy popłynie do danych samorządów, to ja powiem szczerze: w żaden sposób wam nie ufam. Bo Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który wdrożyliście, był po prostu niesprawiedliwy. Wszystkie dokumenty pokazały, że te gminy, w których rządzili ludzie z PiS, dostawały ile? Taka jest prawda na temat waszego Nowego Ładu. To jest po prostu niesprawiedliwość. Pani poseł Barbara Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Szanowni Państwo!

Dziękuję, pani poseł. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wnosząc właściwy projekt ustawy, rząd sam potwierdza w uzasadnieniu, że tzw. Nowy Ład, albo raczej nieład, dobije finansowo samorządy. Jeśli osłabimy samorządy, to osłabimy również mieszkańców. Według wyliczeń samego resortu finansów samorządy co roku tracić będą kwotę prawie 15 mld zł. W ciągu dekady będzie to 145 mld zł. Różnica? Będzie brakować na sport, na edukację, transport, usługi, nie wspominając o kulturze. To jest niszczenie dorobku 30 lat polskiej demokratycznej samorządności. Moje rodzinne miasto Inowrocław straci prawie 20 mln zł.

Panie Ministrze!

Moje pytanie do ministra: Dlaczego państwo nie lubicie samorządów? Lubicie tylko niektórych samorządowców.

Jak pokazał pan poseł Kowalczyk, jego gmina może zyska. Proszę się przeprowadzić.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Prawda o tej ustawie jest taka, że w ogóle samorządów w niej nie wspieracie a fundusze im odbieracie. I gdybyśmy poszukali prostych analogii, to miliony złotych, które chcecie zabrać samorządom, po prostu przekażecie do samorządów, w których rządzą ludzie Prawa i Sprawiedliwości. Miasta w moim okręgu wyborczym na Kujawach: Inowrocław, Bydgoszcz, Żnin, Tuchola - one wszystkie stracą. Ale was to nie obchodzi, bo tam przecież nie rządzi nikt z Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby rządził, to i pieniądze byście szybko znaleźli. Od 2020 r. solą w waszym oku jest samorząd terytorialny, dlatego że nie pozwolił wam przeprowadzić nielegalnych wyborów i sprzeciwił się autokratycznej władzy, która chciała za wszelką cenę te wybory przeprowadzić. Samorząd terytorialny, który powinien być ostoją demokracji, takim pozostanie. Szybciej wy skończycie rządzić, niż samorząd rozbijecie.

Wysoka Izbo! Te, które pochodzą z dochodów podatkowych, bo one są przewidywalne. Wszystkie subwencje, wszystkie dotacje usztywniają budżety samorządowe.

W pierwszym roku to może być równowartość przychodów podatkowych, w kolejnych latach już nie. Mamy doświadczenie, że najlepszy budżet, który otrzymały samorządy, to był tzw. budżet Misiąga. Wtedy jeszcze były depozyty z przychodów budżetowych. Dlatego uważam, że wprowadzanie takiego usztywniającego (Dzwonek) instrumentu jest szkodliwe z punktu widzenia funkcjonowania samorządu. Dziękuję bardzo. Pani poseł Urszula Nowogórska, Koalicja Polska. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Mam takie pytanie, bo w zasadzie większość korporacji samorządowych mówi, że wprowadzenie w obieg prawny tego projektu ustawy spowoduje spadki finansowe w samorządach. Chciałam zapytać, czy rząd, ministerstwo rozważa możliwość całkowitej bądź częściowej możliwości odzyskiwania VAT-u z inwestycji - to, o czym wspomniałam w swoim wystąpieniu. I drugie moje pytanie, bo chciałabym usłyszeć od pana ministra stanowisko w odniesieniu do projektu ustawy, który był procedowany wcześniej, mianowicie o świadczeniu 500+. Te środki finansowe, które były przekazywane na świadczenie 500+ do samorządów, a wchodziły w dochody samorządów i podnosiły wskaźniki, jaki będą miały wpływ, jakie przełożenie, jeżeli chodzi o kondycję finansową samorządów w chwili obecnej po wprowadzeniu tego projektu ustawy? Bo jednoznacznie stanowiska pana ministra nie usłyszałam, dlatego bardzo o to proszę. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zaproponowany projekt ustawy wprowadza m.in. nową część subwencji ogólnej, część inwestycyjną dla gmin, powiatów i województw. To rozwiązanie oczywiście ma przede wszystkim wzmocnić potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego. Jak czytamy w projekcie ustawy, podział środków na poszczególne samorządy będzie dokonywany na podstawie określonego algorytmu. Stąd moje pytanie: Co będzie uwzględniał ten algorytm, jakie będzie zawierał parametry i czy zostanie tak skonstruowany, aby promować samorządy słabsze, żeby maksymalnie ograniczać nierówności pomiędzy poszczególnymi gminami i powiatami? Dziękuję bardzo. Pan poseł Henryk Kowalczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Ta ustawa mówi jasno o algorytmie i sposobie przeliczania. Naprawdę, proszę doczytać. Padały zarzuty, że art. 242 ustawy o finansach publicznych samorządy zaknebluje, jeśli chodzi o możliwość. Właśnie też są zmieniane założenia i lista przychodów, jeśli chodzi o art. 242, więc proszę to przeczytać. Poza tym subwencja, która będzie liczona, zalicza się do dochodów bieżących, nie inwestycyjnych, bieżących. Więc nie ma żadnej różnicy między tą subwencją a dochodami podatkowymi.

Pan poseł Tomasz Ławniczak, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo!

Natomiast generalnie dochody własne samorządów, bo to są inne dochody pochodzące również z podatków lokalnych, wzrosły, generalnie rzecz biorąc, włącznie z PIT-em i CIT-em, o 7%.

Wreszcie sam Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Dzwonek)

Panie Ministrze! Przecież, szanowni państwo, doskonale wiecie, z czym mamy do czynienia, z jaką manipulacją mamy do czynienia. Dzisiaj rozmawiamy o tej ustawie, a w piątek będziemy rozmawiali o ustawie regulującej kwestie dotyczące podatków dochodowych PIT. Mówiąc krótko, dzisiaj ładnie mówicie, że chcecie dać samorządom, a w piątek będziecie im zabierać. A pamiętajcie, że kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Więc prawda jest taka, że nie ma w tej ustawie ani w tych ustawach, które proponujecie, rzeczywistej koncepcji finansowania samorządów. Po prostu znowu zamiast decentralizacji państwa mamy do czynienia z centralizacją państwa, bo wprowadzacie kolejną subwencję, bo chcecie, mówiąc krótko, jako rząd podejmować decyzje, jak będą finansowane samorządy. Dlatego mam pytanie, panie ministrze: Czy planujecie reformę finansów samorządów w Polsce, zwiększenie wpływów i udziałów w podatku PIT, CIT, być może w podatku VAT, żeby (Dzwonek) wreszcie to uregulować? Dziękuję bardzo. Pani poseł Karolina Pawliczak, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Samorządy stracą na polskim bezładzie miliardy złotych. Będzie mniej inwestycji, mniej dróg, chodników i innych ważnych zadań, które mogłyby zostać zrealizowane, gdyby nie ta zabójcza dla polskich samorządów ustawa. Np. Kalisz straci rocznie ponad 49 mln zł, blisko 23 mln - Ostrów Wielkopolski, blisko 30 mln - Leszno, a ponad 13 mln - Jarocin i inne miasta i gminy Wielkopolski oraz całego kraju. To cios w niezależność jednostek samorządowych, który doprowadzi do ich finansowej ruiny. Odczują to mieszkańcy i wielkich metropolii, i małych gmin, i miasteczek. Rekompensaty i subwencje, które proponujecie, to kropla w morzu potrzeb, dlatego mówimy głośne „nie” dla centralizacji państwa i łupienia samorządów. Pytanie, kiedy wreszcie to zrozumiecie i kiedy to zrobicie. Pan poseł Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Pośle Kowalczyk!

Samorządy rzeczywiście zrekompensowałyby te straty, gdybyście zwiększyli udział w podatku PIT, panie ministrze. Dlaczego tak bronicie się i nie chcecie pomóc - rzeczywiście pomóc - samorządom? Jeżeli chodzi o mniejsze gminy, to rzeczywiście można by było dodatkowo wprowadzić tę subwencję rozwojową. Mówi pan, że samorządy nie stracą. Proszę, panie ministrze, powiedzieć mi, jak zrekompensujecie to mieszkańcom Białegostoku - bo to mieszkańcy stracą. Mieszkańcy nie będą mogli cieszyć się z nowych chodników, dróg rowerowych i innych inwestycji. Dziękuję. Teraz głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Sebastian Skuza. Bardzo proszę, panie ministrze.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Subwencja rozwojowa będzie mogła być przeznaczana również na wydatki bieżące. Nie traci ona przymiotu subwencji, to podkreślam. Jak będzie naliczana, czy będzie dbała o jednostki mniejsze? Jak najbardziej tak. W części podstawowej, 60-procentowej, algorytm będzie naliczany liczbą mieszkańców, ale z odpowiednią kwotą minimalną i maksymalną, chroniącą właśnie jednostki małe. Nie będzie tutaj żadnej uznaniowości. Wszystkie przepisy dotyczące subwencji rozwojowej będą przepisami natury ustawowej. Nie ma tutaj miejsca na jakąkolwiek dowolność. Jeszcze raz podkreślę, że gdyby się okazało, że kwota referencyjna, czyli ta, którą same jednostki samorządu terytorialnego wyprognozowały, zwaloryzowana, była niższa od łącznych dochodów z CIT-u i PIT-u, to subwencja rozwojowa będzie musiała ją w pełni uzupełnić.

Tak że mówię jednoznacznie: nie ma wpływu, będzie to neutralne. Padały tu również pytania dotyczące poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Wysoki Sejmie, chciałem zauważyć, że wraz z projektem ustawy do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu została przekazana szczegółowa ocena skutków regulacji.

Jakie tu jest porównanie?

Nie mogę również zgodzić się z twierdzeniem, że subwencja usztywnia budżety samorządowe. Myślę, że subwencja jest bardzo elastycznym, jeżeli nie najbardziej elastycznym dochodem jednostek samorządu terytorialnego.

Są np. modele skandynawskie, gdzie nawet jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość wprowadzenia dodatków do podatków, a nie tylko udziału sztywnego, ale również możliwość określenia pewnych stawek podatkowych. Są też modele z innych krajów, gdzie to transfery budżetowe są największym tego typu źródłem zasilania jednostek samorządu terytorialnego. Tak jak powiedziałem, nie przewidujemy zwiększenia udziału w podatkach i wyjaśniałem dlaczego. Mieliśmy dyskusję z gminami wiejskimi i tam nam jednoznacznie wskazywano na problem, że w gminach wiejskich, gdzie dochody są z podatku rolnego, z emerytur rolniczych czy też z niskich wynagrodzeń, zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych naprawdę nic by nie zmieniło.

Myślę, że niewiele.

Niemniej jednak, szanowni państwo, Wysoki Sejmie, chciałbym zauważyć, że to jest inwestycja rządu w jednostki samorządu terytorialnego.

Subwencja. Pojawiały się jeszcze kwestie związane z inflacją. Sugerowałbym jednak, żeby patrzeć na gospodarkę całościowo, nie tylko przez jeden wskaźnik, bo to naprawdę może być mylące. Teraz krajem, który stosunkowo dobrze radzi sobie z inflacją w Unii Europejskiej, jest, Wysoki Sejmie, Grecja. Myślę, że w całości nie zamienilibyśmy się na sytuację makroekonomiczną. Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład, zawarty w druku nr 1531, do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Marszałek Sejmu proponuje, aby Sejm na podstawie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu wyznaczył komisjom termin przedstawienia sprawozdania umożliwiający rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o pilnym rządowym projekcie ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (druki nr 1533 i 1552) Proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! W imieniu sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawiam sprawozdanie komisji gospodarki druk nr 1552 o pilnym rządowym projekcie ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., druk nr 1533. Marszałek Sejmu zgodnie z art. 73 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 9 września powyższy projekt ustawy do Komisji Gospodarki i Rozwoju do pierwszego czytania. Jednocześnie marszałek Sejmu na podstawie art. 73 ust. 2 regulaminu Sejmu wyznaczyła termin przedstawienia sprawozdania do dnia 15 września 2021 roku.

W trakcie posiedzenia komisji zgłoszonych zostało pięć poprawek.

Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jako pierwszy pan poseł Dariusz Stefaniuk, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wprowadzenie stanu wyjątkowego na części województwa podlaskiego oraz województwa lubelskiego było decyzją trudną, ale świadczyło o odpowiedzialności rządu za bezpieczeństwo obywateli naszego kraju. Stan wyjątkowy swoim obszarem objął 183 miejscowości znajdujące się na terenie ośmiu powiatów Polski Wschodniej. Wbrew narracji, jaką dzisiaj uprawia opozycja parlamentarna, stan wyjątkowy spotkał się z pełnym zrozumieniem okolicznych mieszkańców i przedstawicieli samorządów lokalnych. Osobiście rozmawiałem z wieloma z nich, ponieważ jest to region, w którym mieszkam. Potwierdza to słowa wypowiedziane przez pana ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, że restrykcje w najmniejszym stopniu nie będą ingerowały w życie zawodowe mieszkańców gmin przygranicznych. W przypadku działalności, które nie mogą być prowadzone, rząd proponuje rekompensaty i tej właśnie ustawy dotyczy stanowisko, jakie mam zaszczyt zaprezentować w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Proponujemy przedsiębiorcom oraz rolnikom świadczącym usługi hotelarskie, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także prowadzącym działalność pilota wycieczek czy przewodnika turystycznego rekompensatę. Jest to grupa usługodawców najbardziej dotkniętych wprowadzonymi ograniczeniami. Rekompensata będzie przyznawana przez właściwego wojewodę na wniosek przedsiębiorcy. Zależy nam na jak najszybszej pomocy ww. branżom, dlatego wojewodowie będą rozpatrywać wnioski niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich złożenia. Rekompensatę ustala się za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy w okresie obejmującym miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. Szanowni Państwo! Ta ustawa jest przykładem, że wspólnie jako rząd oraz parlament bierzemy odpowiedzialność za naszych mieszkańców. Nie zostawiamy ich samych sobie i chcemy, aby sytuacja na naszej wschodniej granicy jak najszybciej wróciła do normalności.

Dlatego jako przedstawiciel Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, poseł tej ziemi, ale również mieszkaniec tych terenów rekomenduję przyjęcie tego projektu ustawy, druki nr 1533 i 1552. Bardzo dziękuję. Teraz pan poseł Robert Tyszkiewicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Chyba, panie pośle, żyjemy w różnych rzeczywistościach, bo ja też jestem mieszkańcem tego regionu, też spotykam się, rozmawiam z przedsiębiorcami, z mieszkańcami i chcę panu powiedzieć, że fatalna decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego odcięła ten wspaniały region Rzeczypospolitej od reszty kraju, pozbawiła mieszkańców poczucia bezpieczeństwa, a co najważniejsze, z dnia na dzień odcięła od jednego z podstawowych źródeł dochodu, od dochodu z działalności turystycznej. Gdyby było tak, jak mówi pan poseł, że nie wywołało to żadnych istotnych skutków, nie dyskutowalibyśmy dzisiaj o specustawie o rekompensatach, która ma w pilnym trybie uratować od upadłości szereg przedsiębiorstw i działalności gospodarczych w tym regionie. Nie zgadzam się kategorycznie, nie wiem, skąd biorą się liczby mówiące o ok. 200 przedsiębiorstwach. Zapewniam pana ministra i Wysoką Izbę, że problem praktycznie ogłoszonego lockdownu gospodarczego na tym terenie dotyka znacznie większej liczby przedsiębiorstw. Dlatego dobrze się stało, że rozmawiamy w Sejmie o specjalnej ustawie o rekompensatach, ale aby ta ustawa mogła odegrać swoją rolę, aby rzeczywiście pomogła w potrzebie i uratowała dochody wielu przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i zwykłych obywateli prowadzących działalność i żyjących z turystyki, musi to być ustawa sprawiedliwa i kompletna. Co to znaczy sprawiedliwa? To znaczy taka, która rekompensuje poniesione straty i utracone korzyści na adekwatnym do tych strat poziomie. Nie satysfakcjonuje nas i zapewniam, że także nie satysfakcjonuje przedsiębiorców, adresatów tej pomocy proponowany przez rząd poziom 65%. Dlatego będziemy powtarzać i wnosić: Tylko 80-procentowa rekompensata jest sprawiedliwa i adekwatna, jeżeli chodzi o poniesione straty. Będę w tej kwestii w imieniu Koalicji Obywatelskiej przedstawiał poprawki. Ustawa kompletna to znaczy ustawa obejmująca rzeczywiście większość podmiotów i branż, które ponoszą straty z tytułu wprowadzenia stanu wyjątkowego. Dlatego wnoszę także dzisiaj poprawki dotyczące rozszerzenia prawa do rekompensaty dla branż przewozu turystów i transportu rekreacyjnego, kultury, rozrywki i rekreacji oraz sprzedaży detalicznej produktów spożywczych oraz pamiątek.

Zmiany, o których mówimy, podniosą ten koszt do ok. 10 mln. To jest w skali budżetu naprawdę maleńka kropla. Dlatego zwracam się i apeluję do strony rządowej w imieniu mieszkańców i przedsiębiorców z pogranicza wschodniego, Podlasia i Lubelszczyzny. Panie ministrze, warto z tej okazji skorzystać. Panie marszałku, chciałem na pana ręce przekazać poprawki do projektu ustawy, druki nr 1533 i 1552. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Grabczuk, również Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! nie są wystarczające. Absolutnie. Bardzo prosimy, byście państwo poparli nasze propozycje, tak by przepisy dotyczyły również szeroko rozumianego transportu, zwłaszcza transportu rekreacyjnego i przewozu turystów. Nie ma turystów - nie ma dochodów. We Włodawie miał się odbyć Festiwal Trzech Kultur. Nie odbył się. Zostały poniesione różnego rodzaju koszty. Nie ma turystów. Sklepy z pamiątkami, również sklepy spożywcze mają znacznie mniejsze obroty. Zrekompensujmy to również i sklepom. Cieszę się, że wczoraj nasze dwie propozycje zostały zaakceptowane, to dotyczy wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz (Dzwonek) kontroli wojewody. Ostatnie zdanie, panie marszałku, proszę państwa. Nie upierajmy się przy tych 65%.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jako Podlasianin mam przyjemność przedstawić w imieniu klubu Lewicy stanowisko dotyczące projektu ustawy o rekompensacie dla podmiotów gospodarczych w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. 2 tygodnie - na tyle miała zostać zamknięta branża gastronomiczna w czasie pandemii.

Największe straty poniósł wtedy sektor usługowy, w tym branża gastronomiczna, która została dotknięta najdłuższymi obostrzeniami. Branża ta notowała najgorsze wyniki w historii, spadek liczby klientów w ciągu roku przekroczył 90%. Ponad 200 tys. osób straciło pracę w gastronomii lub zmieniło formę zatrudnienia. Kolejne tarcze oparte na klasyfikacji PKD okazywały się dziurawym sitem niegwarantującym wszystkim takiej samej niezbędnej pomocy. W końcu w czerwcu 2021 r. po 16 miesiącach od pierwszego zamknięcia wróciliśmy do jako takiej normalności, choć jeszcze niepełnej wolności. Niestety ta normalność nie trwała długo. Dla 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim skończyła się ona właśnie 2 września, gdy do stanu pandemii dołączył stan wyjątkowy. W czasie stanu wyjątkowego na terenie tych miejscowości obowiązuje zakaz przebywania w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach oraz zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzenia w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych niebędących imprezami masowymi. Te ograniczenia już ponownie powodują straty w lokalnych firmach, m.in. właśnie w branży hotelarskiej czy gastronomicznej. W tej sytuacji przyjęty w minioną środę przez rząd projekt rekompensat o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności praw i obywatela to konieczne i oczekiwane wsparcie. Zgodnie z projektem rekompensatę będą mogli otrzymać przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako piloci wycieczek lub przewodnicy turystyczni, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii. Na razie na pieniądze mogą także liczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki. Czy i tym razem ta pomoc okaże się dziurawa? Zdaniem Lewicy nie. Proponowana w projekcie rekompensata w wysokości 60% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. to dla tak dotkniętych kolejnymi obostrzeniami sektora usług zdecydowanie za mało. Dlatego w imieniu klubu Lewicy składam poprawkę zwiększającą proponowane wsparcie do 80%. Klub Lewicy popiera wcześniejsze przedłożenie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, Koalicja Polska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zabierając głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści, chcę powiedzieć, że ta ustawa jest potrzebna. To jest pilna ustawa, dlatego że to państwo wprowadziło restrykcje, ograniczenia praw i wolności, ograniczyło działalność gospodarczą wielu podmiotom, wielu osobom fizycznym, dlatego należy im się pilna pomoc. Nie wnikam w to, czy wprowadzenie tych ograniczeń było słuszne czy niesłuszne. Nie powinno być tutaj dyskusji, czy 65% jest wystarczającym odsetkiem, dlatego że wszystkie udowodnione straty powinny być pokryte.

Składam również trzy poprawki do tego projektu ustawy, gdyż myślę, że ona jest niepełna i niedoskonała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Zdumienie mnie ogarnia, jak słyszę, kto nagle jest przeciwko ograniczeniom związanym ze stanem wyjątkowym.

To, co się tam działo, ten cyrk, który urządzali posłowie zarówno z Koalicji Obywatelskiej, jak i z Lewicy, którzy atakowali Straż Graniczną za to, że wykonuje swoje obowiązki, że broni granicy państwa. Wstydźcie się za to. Ludność miała dosyć tego, że im biegają po polach imigranci, a za tymi imigrantami biegają jeszcze oszalali posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy starają się ich wprowadzić do Polski. Tego miała dość ludność na Podlasiu. Naprawdę, trochę samokrytyki, trochę realizmu i wstydu. Szanowni Państwo! Oczywiście to było potrzebne. Potrzebne jest, panie ministrze, ogrodzenie z prawdziwego zdarzenia na granicy. Nie ma - jak na granicy zachodniej czy południowej - naturalnych przeszkód, cieków wodnych, nie ma gór.

Poprawki, które składamy jako Konfederacja, idą w dwóch kierunkach. Po pierwsze, mają na celu wykreślenie obligatoryjnego przeprowadzania kontroli w przypadku przyznania przedsiębiorcy rekompensaty przekraczającej 65 tys. zł.

Dziękuję. Pani poseł Joanna Mucha, Polska 2050. Panie Marszałku! Sprowokowana słowami mojego przedmówcy zacznę od czegoś innego, nie od tego, od czego miałam zacząć to wystąpienie. Otóż chciałabym powiedzieć, że pan poseł Winnicki i państwo z PiS cały czas nie rozumieją jednej rzeczy. Polacy są różni. W naszym przekonaniu tych drugich jest więcej. Z naszych rozmów, z naszych kontaktów wynika, że tych drugich jest więcej. Nie, Polacy są różni. To nie jest tak, panie ministrze, że stan wyjątkowy można sobie wprowadzać po to, żeby władzy było wygodnie.

Od tego jesteście, żeby ludziom było lepiej. Nawet jeśli wprowadzacie dzisiaj ustawę, która coś łata, która coś naprawia, to i tak krzywdzicie ludzi.

To nie jest tak, że wszystkim zrekompensujecie utracone zarobki. Ale ja bym prosiła, żeby pan mi nie przeszkadzał.

Mamy dwa hotele w Janowie Podlaskim. Do tego drugiego hotelu ludzie też nie przyjadą, bo stadnina jest zamknięta.

Nie uzyskają swoich dochodów, bo poniosły koszty w związku z organizacją różnego rodzaju imprez kulturalnych, które miały się odbyć, i nie dostaną od was rekompensaty.

Ważniejsze jest to, żebyście po prostu nie krzywdzili ludzi. Dziękuję. Przechodzimy do pytań. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Panie pośle, bardzo proszę.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Pytam o to dlatego, że to jest taki region, w którym szczyt przypada nie w czerwcu, lipcu, sierpniu, tylko właśnie we wrześniu.

Bo ta propozycja na pewno nie jest sprawiedliwa. Ona jest jakaś, ale na pewno nie jest sprawiedliwa. Dlaczego one nie są uwzględnione w tym projekcie ustawy?

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Kwestię roszczeń o odszkodowania z tytułu stanów nadzwyczajnych kompleksowo reguluje ustawa z 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Dodatkowo, co też jest bardzo istotne, każdy, kto otrzyma rekompensatę w wysokości 65%, nie będzie mógł zgodnie z ustawą dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania na zasadach ogólnych. Lewica zgłosiła wniosek: rekompensata powinna wynosić 80%. Pan poseł Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dlaczego tak karzecie podlaskich i lubelskich przedsiębiorców?

Z dnia na dzień ludzie stracili środki do życia. Panie ministrze, dlaczego to będzie rekompensata w wysokości tylko 65%? Dlaczego nie chcecie się przychylić do naszych poprawek? Proponujemy 80%. To nie tak wiele, a tym ludziom naprawdę może uratować biznesy.

Nie ma pana posła. Pan poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiedzialność za przedsiębiorców to też myślenie o tym, jak będą mogli wykonywać swoją działalność w sytuacjach kryzysowych. To, że wprowadziliśmy stan wyjątkowy, nie powinno być elementem, który wyłączy tę odpowiedzialność. Każdy projekt ustawy, który ma dać szansę na rekompensaty, wyrównanie strat, to projekt rozsądny. Tyle że tego rozsądku brakuje w całym podejściu do spraw związanych z sytuacją na granicy i dotyczących garstki uchodźców, którzy potrzebują pomocy.

Wysoka Izbo! Wprowadziliście ten stan wyjątkowy z dnia na dzień tylko po to, żeby odciąć nas wszystkich, społeczeństwo, od informacji, żeby wprowadzić strach wśród mieszkańców i wśród wszystkich obywateli i obywatelek Polski. Wprowadziliście stan wyjątkowy, całkowicie eliminując ruch turystyczny na tym terenie. Odcięto od dochodów branżę gastronomiczną, branżę turystyczną, ale także branżę usługową i branżę handlową, a rekompensaty wprowadzacie tylko dla hoteli, gastronomii i branży turystycznej. A co z ludźmi, którzy prowadzą na tym terenie sklepy? A co z ludźmi, którzy prowadzą na tym terenie inne usługi? Czy oni nie są godni tego, żeby także uzyskać rekompensatę? Pan poseł Wiesław Buż, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podzielam obawę, czy rekompensaty zostały właściwie adresowane do wszystkich podmiotów prawnych i fizycznych. Jest wiele firm, które nie prowadzą ewidencji uzyskanych przychodów. Na jakiej podstawie, panie ministrze, złożą wnioski o wypłatę rekompensaty, która ma wynieść 65% średniego miesięcznego przychodu? Często jest tak, że przewodnicy i inne osoby prowadzące działalność rozliczają się ryczałtowo i nie mają obowiązku rejestracji przychodów. Czy wystarczy, że złożą wniosek i deklarację, oświadczenie o wysokości miesięcznego przychodu, i to będzie podstawa do wypłaty rekompensaty? Ponadto również uważam, że 65-procentowa rekompensata jest zbyt niska i należy ją podwyższyć do minimum 80%. Kolejny problem.

Mam jedno zasadnicze pytanie. Uważam, że państwo osiągnęliście ten cel propagandowy, wprowadzając stan wyjątkowy. Pytam, dlatego że klient komercyjny nie decyduje się na rezerwacje w ostatnim czasie. Dobrze by było, gdyby ten sygnał przyszedł znacznie, znacznie wcześniej.

Wysoki Sejmie! Jak widzimy, największe kontrowersje budzi ustalenie kwoty rekompensaty. W ustawie zakłada się, że jest to 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy ze świadczonych usług prowadzonych w czerwcu, lipcu i sierpniu, a więc w okresie najlepszych miesięcy turystycznych.

I druga rzecz jest taka, że musimy pamiętać, że wprowadzenie stanu wyjątkowego to jest racja stanu. Wysoka Izbo! Rzeczywiście pomijamy ten aspekt wprowadzenia stanu wyjątkowego, bo to już się stało, natomiast ustawa ma uregulować kwestie rekompensat za poniesione straty za to, że w tym okresie nie jest prowadzona działalność gospodarcza przez różne podmioty działające na tym terenie. Po pierwsze, w projektowanej ustawie jest wyliczona kwota ok. 7 mln zł, w sumie dla ok. 200 przedsiębiorstw, więc moje pytanie jest takie, czy w tych wszystkich gminach jest tylko 200 podmiotów gospodarczych, które tam funkcjonują. Już nie chcę powtarzać tego pytania o sposób wyliczenia, że to akurat 65%, a nie 70%, 80% czy 100%. Czy szacowaliście również z tego powodu zmniejszenie wpływów do budżetów samorządów na tym terenie? Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Moi przedmówcy, pan poseł Grabczuk zgłaszał poprawkę dotyczącą transportu, w tym kajaków, które pływają po rzece Bug. Wydaje mi się, że to jest umiejscowione w ustawie i te firmy będą mogły uzyskać odszkodowanie i to jest moje pytanie do pana ministra. Chciałem się odnieść do wypowiedzi pani Muchy i pana Krawczyka, które moim zdaniem są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Nie wiem, czy państwo jako posłowie z Lublina w ogóle byliście na tej granicy, być może kiedyś Zapraszam, żebyście teraz przyjechali. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, bo ja tam byłem w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu, że sklepy działają, można spokojnie korzystać z kościołów, można spokojnie korzystać ze szkół, dzieci są dowożone do szkół, można dojechać na korepetycje, można wjechać i wyjechać z tej strefy, więc, szanowni państwo, opowiadacie bajki, nie znacie tej sytuacji, być może naczytaliście się w Internecie, a nie wiecie, jak tam jest, i opowiadacie to, szkalując tych ludzi.

Panie Ministrze!

I nieważne, czy wykonał usługę, czy nie. Druga rzecz. Dlaczego nie objęto wszystkich podmiotów zarejestrowanych w tych regionach, które prowadzą działalność gospodarczą, a są w stanie udowodnić, że poniosły stratę? To by było właściwe i rozsądne podejście.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Krutul, Lewica. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie Ministrze Wąsik! Mam nadzieję, że nie mniejsze niż 80% podlaskim i lubelskim przedsiębiorcom w pasie przygranicznym z Białorusią objętych stanem wyjątkowym. To nie wina przedsiębiorców, że 100-tysięczna armia żołnierzy zawodowych nie jest w stanie sobie poradzić z pasem granicznym z Białorusią. Pan poseł Robert Tyszkiewicz, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Najpierw chciałem się odnieść do wypowiedzi pana posła Winnickiego. Ale gdyby prawdą było to, co pan mówił, że stan wyjątkowy został wprowadzony z powodu pieszych wycieczek kilku posłów i aktywistów na naszą wschodnią granicę, to to by oznaczało, że jesteśmy państwem kabaretowym. Ja aż tak złego zdania o naszym państwie nie mam.

To znaczy, po pierwsze, czy będzie po zakończeniu stanu wyjątkowego specjalny program odbudowy wizerunku tej części województwa podlaskiego i lubelskiego, tej części turystycznej przygranicznej jako części bezpiecznej dla turystów?

Wysoka Izbo! Wprowadziliście stan wyjątkowy tylko po to, żeby media i organizacje pozarządowe nie mogły relacjonować tego, jak łamiecie prawo i w jak nieludzki sposób zachowujecie się na granicy. Od wielu tygodni grupa Afgańczyków i Afganek jest nielegalnie blokowana przez polskie i białoruskie służby. Zamiast szklanki wody otrzymali przemoc. Cały czas dowiadujemy się o kolejnych nielegalnych push-backach. Nie wprowadziliście stanu wyjątkowego jesienią i wiosną, gdy dziennie z powodu pandemii umierało kilkadziesiąt osób. Robicie to teraz, żeby ukryć swoją przemoc, ksenofobię i bezprawie. Cierpią na tym również mieszkańcy Podlasia i turystyka. Żadną rekompensatą nie zwrócicie im straconego czasu i nie zmażecie wizerunku frontu wojennego, który systematycznie tam budujecie. Ten stan wyjątkowy jest hańbą dla polskiego państwa, jest aktem tchórzostwa polskiego rządu. Żadnym manewrem prawdy nie ukryjecie. Pan poseł Robert Winnicki w trybie sprostowania. Wysoka Izbo! Panie pośle, pan sobie sam zaprzeczył w tej samej wypowiedzi, mówiąc o tym, że z jednej strony nie ma żadnego zagrożenia i że państwo polskie, ja się zgadzam, wykazuje się tutaj słabością.

Tak to wygląda. To wtedy to będzie ziemia bezpieczna, bo nie będą tam przechodzili nielegalni imigranci. Bardzo proste. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Teraz głos zabierze. sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Maciej Wąsik.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z uwagą przysłuchiwałem się wystąpieniom pań i panów posłów i przyznam się, że trochę zazdroszczę Litwinom i Łotyszom opozycji - opozycji, która wspiera rząd w momencie, kiedy pojawia się zagrożenie. Ale my dzisiaj mówimy o wsparciu tych, którzy ucierpieli w momencie, kiedy został wprowadzony stan wyjątkowy, który ograniczył dostęp do tych terenów przede wszystkim turystom. I chciałbym państwu odpowiedzieć na tę część pytań merytorycznych, które tu padły. Dlatego ustawa pilna, która daje rekompensatę utraconych dochodów, utraconych zysków i dochodów. Pan poseł Szopiński mówił, że jest ustawa z 2002 r., która mówi o wyrównywaniu szkód w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego.

Okazuje się, że rzeczywiście możemy wyrównywać szkody, jeżeli ktoś poniesie szkodę, czyli np. zawali się ściana po wjeździe samochodu Straży Granicznej. Ale my dajemy ludziom rekompensatę utraconych dochodów. Dlaczego 65%? Otóż przyczyny są dwie. Przede wszystkim porównujemy te 65% do wysokiego sezonu turystycznego, bo mówimy tu o szerokiej branży turystycznej - hotele, agroturystyka, gastronomia. Także dziękuję państwu posłom za zwrócenie uwagi, że ta ustawa była niepełna, ale rzeczywiście nie planowaliśmy tego stanu wyjątkowego od dawna, działaliśmy szybko i katalog tych branż w wyniku wspólnej pracy w komisji został uzupełniony. Ukłon dla posłów, którzy zwrócili na to uwagę. Dajemy 65% dochodów, przepraszam, przychodów, nie dochodów - przychody to więcej niż dochody - przychodów wysokiego sezonu turystycznego. Te pieniądze nie podlegają opodatkowaniu. Nie podlegają opodatkowaniu. Zdajemy też sobie sprawę, że jednak w branży gastronomicznej, turystycznej, w wypożyczalniach, jeżeli ktoś nie prowadzi działalności, to także zmniejsza sobie część kosztów, nie wszystkie oczywiście, bo pewne koszty są stałe, ale część kosztów zmniejsza.

Jestem o tym przekonany, szanowni państwo. Gdyby pani poseł mogła nie krzyczeć z sali do mnie, dobrze? Dziękuję bardzo. Kiedy rząd skierował wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego do prezydenta, natychmiast zrobiliśmy wideokonferencję ze wszystkimi samorządowcami tamtego regionu. A przypomnę, że ten stan wyjątkowy, szanowni państwo, nie jest w całym województwie lubelskim i podlaskim, nie jest nawet we wszystkich gminach przygranicznych, tylko w ich częściach. To kilka kilometrów, 3 w niektórych miejscach, w niektórych 5, w niektórych może trochę więcej, ale to jest mała część. Mało tego, wojewodowie zbadali, ilu jest przedsiębiorców danego rodzaju. Ale wiemy, że pomoc im się należy, bo rzeczywiście z dnia na dzień zakazano turystom korzystać z ich usług.

Granice.

Bardzo proszę, sprawozdawca komisji pan poseł Krzysztof Tchórzewski. Wysoki Sejmie! Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju poświęcone tej ustawie przebiegało bardzo dynamicznie, ale było w pełni merytoryczne, dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim posłom komisji za zaangażowanie się w prace nad tą ustawą.

Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Gospodarki i Rozwoju w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1507 i 1546) Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na dwóch posiedzeniach - co wymaga podkreślenia - w dniach 8 i 14 września br. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalił załączony projekt ustawy. Zgłoszone wnioski podlegały analizie.

Bardzo dziękuję. Sejm uchwalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Wydaje mi się, że pytanie kluczowe, jakie trzeba sobie zadać podczas procedowania nad tą ustawą - tą może najbardziej, ale także nad innymi ustawami - brzmi: Po co my tutaj jesteśmy, jaką rolę, jaką funkcję powinien pełnić polski parlamentarzysta, polski poseł, polski senator, zasiadając w Wysokiej Izbie? Zdawać by się mogło, że odpowiedź na to pytanie jest prosta, wręcz banalna. Jesteśmy tutaj po to, żeby Polakom, tym osobom, które powierzyły nam te zaszczytne funkcje posłów, senatorów, żyło się bezpiecznie i dobrze. A dzisiaj dotykamy materii, która dotyczy tego pierwszego elementu: żeby nam się żyło bezpiecznie.

I tu następuje pewne powiązanie, ponieważ przed chwilą rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy o kwestiach dotyczących rekompensaty dla przedsiębiorców, których dotknęło wprowadzenie stanu wyjątkowego, i wydaje mi się, że właśnie te dwa tematy, o których dyskutujemy, niejako się przenikają, są ze sobą powiązane. I może właśnie dlatego warto o nich powiedzieć, warto o nich wspomnieć, ponieważ mieliśmy okazję jako członkowie sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako prezydium, być na granicy polsko-białoruskiej, ale także uczestniczyć w niejawnych rozmowach, które ukazywały nam ten problem bardzo dogłębnie, konkretnie i bardzo merytorycznie.

Po tych wszystkich zdarzeniach, które miały miejsce, po tych wszystkich dyskusjach, które miały miejsce, myślałem, że nastąpi otrzeźwienie, że nastąpi zrozumienie tego, co tak na dobrą sprawę dzieje się na granicy. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Mieliśmy okazję wysłuchać bzdurnych wypowiedzi posłów dotyczących podejścia do bezpieczeństwa Polaków, podejścia do bezpieczeństwa ludzi, którzy tam mieszkają, którzy po prostu tego nie rozumieją.

To jest przerażające.

Bezpieczeństwo, proszę państwa, to jest coś, do czego jesteśmy tutaj powołani i zobowiązani - bezpieczeństwo pod każdym względem, sposób przewidywania tego, co się może złego wydarzyć na polskiej granicy, jakie mogą być efekty tego działania, także nieodpowiedzialnego działania państwa. W związku z tym, jeżeli nie trafiają do was argumenty osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo naszego kraju, to dlaczego nie trafiają do was argumenty waszych autorytetów z Unii Europejskiej, która jednoznacznie wypowiada się na ten temat, wskazując, żeby po prostu granicy polskiej, granicy Unii Europejskiej bronić i ją chronić. Proszę państwa, ta ustawa idzie właśnie w tym kierunku, idzie w kierunku obrony polskich obywateli przed niebezpieczeństwem, które - być może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę - jest bardzo duże, jest wręcz niewyobrażalne. Dlatego w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałbym zarekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy z prośbą - chodzi o to, co mówił pan minister w swoim poprzednim wystąpieniu dotyczącym poprzedniego punktu - abyście się państwo opamiętali i wzięli przykład z naszych przyjaciół z Litwy i z innych krajów (Dzwonek), które potrafią myśleć w kategoriach bezpieczeństwa. Pan poseł Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie mam wątpliwości co do tego, że działania podejmowane przez władzę, niezależnie oczywiście od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, powinny być rozsądne, odpowiedzialne, legalne, niebudzące wątpliwości, dążące do osiągnięcia porozumienia ponad politycznymi podziałami. W sytuacji zagrożenia, w sytuacji gdy wchodzi w grę kwestia bezpieczeństwa, niezwykle ważna jest solidarność, także zaufanie do rządzących, ale zaufanie powstaje, gdy władza nie pręży muskułów, ale tworzy i respektuje prawo, jest wiarygodna w tym, co czyni. Dlatego też odpowiedzialna władza powinna zapewnić bezpieczeństwo obywateli, strzegąc granic, pilnując porządku, ale w demokratycznym państwie prawa także podejmując działania na podstawie i w granicach tegoż prawa. Nie możemy pozwolić sobie na chaos prawny, a na taką sytuację właśnie czekają Łukaszenka, Putin i im podobni. Odpowiedzialna władza potrafi połączyć ochronę granic, bezpieczeństwo i porządek publiczny, przestrzeganie prawa, w tym przestrzeganie naszego polskiego prawa, prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego, ale także działania humanitarne związane z przestrzeganiem praw człowieka. Skoro potrzebne są dziś zmiany w przepisach prawa, aby dostosować je do aktualnej sytuacji, to dlaczego nie można przyjąć rozwiązań, które są zgodne z prawem i będą przy tym gwarantować bezpieczeństwo i stabilizację?

Projekt narusza przepisy tzw. dyrektywy proceduralnej.

A to wszystko odbywa się także w sytuacji, gdy Białoruś wypowiedziała umowę o readmisji przeciwdziałającej nielegalnej migracji. Wysoka Izbo! Negatywną opinię dotyczącą omawianego projektu przedstawiły m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, przedstawicielstwo wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych, jak również Biuro Analiz Sejmowych przygotowujące przecież opinie dla nas, dla posłów. Nie mówię o tym wszystkim tylko i wyłącznie po to, by wytykać państwu błędy, ale przede wszystkim po to, by zachęcić do dialogu i wypracowania bezpiecznych rozwiązań, tak w rozumieniu bezpieczeństwa granicznego, jak i bezpieczeństwa prawnego. Trzeba pokazać reżimom, że jesteśmy od nich mądrzejsi. Nie będziemy uczestniczyć w ich grze, to oni chcieliby destabilizacji naszego państwa. Dlatego władza nie może przygotowywać prawa, które jest niezgodne z podstawowymi zasadami demokratycznego państwa, w którym nie respektuje się praw człowieka i nie przestrzega norm prawnych, umów i zawartych konwencji. Oni na to czekają. Właśnie to jest ten kierunek, którego nie można obierać. Właśnie trzeba obierać przeciwny kierunek. Dlatego też w duchu odpowiedzialności za Polskę Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska składa poprawki do rządowego projektu ustawy, które pozwalają na uniknięcie naruszenia podstawowych standardów prawnych. Od ich przyjęcia uzależniamy nasze dalsze procedowanie. Jednocześnie, Wysoka Izbo, nie mamy wątpliwości, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, ale także przestrzeganie prawa oraz tzw. prawnoczłowieczego podejścia, które odpowiada konstytucyjnej zasadzie godności człowieka, a dodatkowo jest przejawem zwykłego humanitaryzmu.

Dziękuję. Pan poseł Maciej Konieczny, Lewica. Wysoka Izbo! Ogromna większość z nich przeżyje wojnę. Rok 1982 - podczas trwania stanu wojennego przez austriackie obozy przejściowe w Traiskirchen przewija się 30 tys. Polaków. Mimo że większości z nich nie grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo w ojczyźnie, otrzymują oni azyl w Austrii i innych krajach Zachodu. Początek lat dwutysięcznych - Polska przyjmuje 100 tys. uciekinierów przed wojną w Czeczenii, ratując życie wielu z nich. Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla stabilności i bezpieczeństwa kraju.

Statek zostaje zawrócony, ogromna większość pasażerów wkrótce potem ginie w komorach gazowych. Wielokrotnie w naszej historii Polacy uciekający przed wojną i prześladowaniami znajdowali schronienie w innych krajach. Po wielokroć to Polska stawała się bezpieczną przystanią dla uciekinierów. Prawo do azylu nie znalazło się w konwencji genewskiej, w prawie europejskim, w polskiej konstytucji przez przypadek. To podstawowe prawo każdego człowieka, tak jak podstawową potrzebą każdego człowieka jest bezpieczeństwo i szukanie schronienia dla siebie i swoich bliskich, często przed wojną, przed torturami, przed prześladowaniami. Mówimy o sprawach zupełnie podstawowych, głęboko zakorzenionych w europejskiej kulturze, w chrześcijańskiej tradycji, w polskiej tradycji gościnności. A jednak rządząca prawica chce wyrzucić to wszystko do kosza. Chce zrezygnować z respektowania podstawowego ludzkiego prawa do schronienia i czyni to przy okazji pierwszej lepszej prowokacji sąsiedniego reżimu, bo tym de facto jest ta ustawa. Jest porzuceniem prawa do azylu, próbą legalizacji tego, co już teraz dzieje się na naszej granicy, próbą legalizacji wywożenia ludzi do lasu, przerzucania ich siłą na białoruską stronę, próbą legalizacji praktyk, które być może przystoją białoruskiej dyktaturze, ale już nie demokratycznej Polsce. Obowiązkiem Polski jest zweryfikowanie wniosków azylowych także tych osób, które przekraczają zieloną granicę. To w świetle prawa międzynarodowego, w świetle prawa europejskiego, w świetle polskiej konstytucji nie pozostawia żadnych wątpliwości. Po prostu nie możemy wyrzucać tych ludzi z kraju bez sprawdzenia, czy nie grożą im z tego powodu śmierć, tortury czy prześladowanie. Nie możemy podejmować takich decyzji bez możliwości odwołania. Naprawdę szanujmy swoją inteligencję. Dochodzenie swoich praw przed polskim sądem z terenu Afganistanu, Somalii czy Syrii to jest czysta fikcja, i doskonale panowie o tym wiecie. Tą ustawą chcecie wyrzucić do kosza coś niezwykle cennego, coś, co towarzyszyło nam od dawna, otwartość na bliskiego w potrzebie, kawałek zwykłego człowieczeństwa. Niedawno jeszcze chodziła do szkoły w Kabulu. Teraz jest najmłodszą z grupy Afganek i Afgańczyków, która przez wiele tygodni koczowała w Polsce pod gołym niebem. Chcecie wyrzucić do kosza szanse 16-letniej Mariam na to, żeby chodziła do szkoły, bo ona powinna być w szkole, nie w rządzonym przez talibów Afganistanie, nie na łasce białoruskiego reżimu, dla którego jest tylko bezwolnym przedmiotem, ale jak każde dziecko - w szkole. I nad tym, drodzy państwo, będziemy głosować w piątek. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Przedstawicielstwo wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Polsce przekazało w dniu dzisiejszym do Sejmu stanowisko dotyczące tej ustawy. Jest w nim napisane, że zaproponowane rozwiązania są sprzeczne z konwencją genewską z 1951 r., Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także z dotychczasowym orzecznictwem Unii Europejskiej w tym zakresie. Napisane jest, że rozwiązania zaproponowane przez rząd są niezgodne z wiążącymi Polskę przepisami prawa międzynarodowego, ponieważ ustawa w takim kształcie może oznaczać zagrożenie dla wolności i życia ludzi zmuszonych do ucieczki. Przedstawicielstwo wysokiego komisarza skierowało zatem do Wysokiego Sejmu to stanowisko. Wysoki Sejmie! Kieruję ten apel i stanowisko wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców do rządu i proszę rząd o zajęcie stanowiska i opinię, gdyż nie można przejść do porządku dziennego nad opinią, że proponowane rozwiązania są niezgodne z wiążącymi Polskę przepisami prawa międzynarodowego.

Pan poseł Marek Biernacki, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sprawie jest bardzo istotny kontekst polityczny, który rozgrywa się cały czas na naszych oczach. To z jednej strony jest upadek Afganistanu, duży ruch migracyjny, polityka Łukaszenki, który objęty sankcjami działa w sposób szalony i chaotyczny. Mamy cały ten kontekst, który jest bardzo istotny i nakłada się na tę sytuację. Ustawa, o której mówimy, ma charakter ekstraordynaryjny.

A więc ta sytuacja narastała.

Polskie środowiska prawnicze krytycznie wypowiadały się o tej ustawie. Do tego też dochodzą takie instytucje jak fundacja helsińska, nasz BAS, ale też, co jest istotne, przedstawicielstwo wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych. Ta ustawa łamie prawo krajowe, prawo europejskie, prawo związane z Schengen, a przede wszystkim konwencję genewską.

Ale czy ta ustawa będzie też ustawą skuteczną?

Ale zakładamy, że będziemy chcieli uchodźców z Iraku skierować do Iraku.

Nie będziemy tworzyli obozów na lotnisku w Bagdadzie, ani nowych na granicy z Białorusią. Czy nie lepiej jest wykorzystać istniejące już narzędzia, które funkcjonują w Polsce, i je poprawić, żeby funkcjonowały lepiej?

I dobrze, że Polska ich przyjęła. Opozycja wspiera te działania rządu.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Szykuje się nam, jak mówią eksperci, kolejny kryzys migracyjny podobny do tego z 2015 r. PiS-owski rząd reaguje w sposób spóźniony, mało zdecydowany, ale trafny. Trafnym posunięciem było wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Nikt nie przewidział, że taka sytuacja się może wydarzyć. Tak że to jest taki mur chiński na miarę PiS-owskich możliwości, można rzec.

Szanowni Państwo! Pytam: Gdzie jest solidarność europejska? Było oświadczenie Komisji Europejskiej, ale gdzie jest konkretna pomoc?

Warto zajrzeć do statystyk przestępczości.

Wyszyńskiego, który naucza, jeżeli chodzi o porządek miłości, jak to wygląda. Kontekst koordynacyjny Łukaszenki, kontekst religijny, jeżeli chodzi o zagrożenie islamistyczne. Szanowni państwo, dlaczego kraje islamskie nie przyjmują islamskich uchodźców, ale są gotowe do tego, żeby sponsorować meczety w Polsce?

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W Sejmie jest takie powiedzenie, że złym projektom powinno wybijać się zęby poprawkami. Ale są takie projekty, które są złe, niedopracowane i którym nie pomogą nawet najlepsze poprawki. Tym projektom nie ma co wybijać. Prawa nie tworzy się szybko i doraźnie. W uzasadnieniu tego projektu czytamy o zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie porządku publicznego. Wszyscy chcemy i bezpieczeństwa, i porządku, ale niezależni obserwatorzy zwracają uwagę na to, że ustawę wprowadza się po to, by legalizować istniejące praktyki wywózek osób przekraczających polską granicę, a to łamie obowiązującą nasz kraj konwencję genewską, ale również europejską konwencję praw człowieka oraz orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przecież istnieją normy prawa międzynarodowego, panie ministrze, a tym projektem wybijacie, a nawet wyrywacie, zęby przepisom, które zapewniają prawa cudzoziemcom. Jeden z profesorów prawa, kiedy prosił studentów o rozwiązywanie kazusów, bardzo często pytał, czy ich stanowisko byłoby inne, gdyby rozwiązanie problemu dotyczyło konkretnie ich. Panie ministrze, czy gdyby to pan był na miejscu cudzoziemców, to chciałby pan przestrzegania wobec pana międzynarodowego prawa, międzynarodowych norm? Obrady komisji pokazały, że projektodawcy nie słuchają prawników, za nic mają fachowców od prawa międzynarodowego, a to niestety może być bardzo kosztowne dla Polski. Koło Parlamentarne Polska 2050 nie poprze tego projektu. Dziękuję. Do pytań zapisali się posłowie.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Oczywiście sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest poważna. Poza tym na Białorusi rządzi człowiek, o którym można powiedzieć wiele rzeczy, ale nie to, że jest stabilny i przewidywalny. W związku z tym ta sytuacja jest nieprzewidywalna.

A więc, panie ministrze, mówi pan o zaufaniu, a z pewnością po waszej stronie, po stronie rządu nie dajecie powodów do tego, żeby wam ufać. Po drugie, jeżeli sytuacja jest poważna, to zwołuje się Radę Bezpieczeństwa Narodowego i informuje się liderów partyjnych o tym, jakie są problemy, a nie straszy, tak jak jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który przyszedł (Dzwonek) i straszył, jakie to wielkie zagrożenia. Panie Ministrze! Przecież z Białorusią nie ma umowy o readmisji. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Mam pytanie dotyczące tak naprawdę sytuacji dzieci.

Pan poseł Jan Szopiński, Lewica.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Kryzys polsko-białoruski rzeczywiście wymaga podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa i porządku w naszym kraju. Natomiast czy ta ustawa musi zostać wprowadzona na stałe? Tak pisze o tym wysoki komisarz ONZ. Dlaczego ustawa z jednej strony chroni nasz kraj, a z drugiej strony narusza prawo międzynarodowe? Czy nie można, panie ministrze, wszystkich tych opinii, które zostały skierowane do rządu, tak ująć w tej ustawie, aby rzeczywiście, tak jak to jest na Litwie, nie była ona ustawą wprowadzoną na stałe, a była ustawą czasową? Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Każdy człowiek ma prawa - prawa naturalne, prawa chronione przez konwencje humanitarne. Jakie prawa mają ci ludzie? Pomijając wszystkie opowieści o tym, że są to przyjaciele Łukaszenki, nasi straszni wrogowie, trzeba powiedzieć, że to są to ludzie cierpiący, potrzebujący różnorodnej pomocy, a przede wszystkim ludzie mający prawo do tego, żeby ich zarejestrować, jeśli przekraczają granicę, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia.

Czy mają jakiekolwiek prawa?

Wysoka Izbo! 29 sierpnia trzech Afgańczyków - Hamidullah, Naqibullah i Ahmad - przekroczyło granicę i poprosiło Straż Graniczną o status uchodźcy. Uciekli z kraju, w którym panuje wojna, a władzę przejęli Talibowie. Łamiąc prawo, wywiozła tych chłopaków w nocy do ścisłego rezerwatu w Puszczy Białowieskiej i wypchnęła na terytorium Białorusi. Strażnicy grozili im bronią i mówili - idźcie, tam są Niemcy. Na szczęście wraz z grupą aktywistów i aktywistek udało nam się ich odnaleźć i pomóc im, więc teraz są bezpieczni. Ta ustawa ma legalizować bestialskie praktyki, które są niestety powszechne na naszej granicy. To łamanie prawa, to łamanie konstytucji i konwencji genewskiej. Prawa człowieka są święte, nie możecie ich łamać dla własnych chwilowych potrzeb politycznych. Nie ma zgody na zarządzanie strachem, nie ma zgody na przemoc.

Panie Przewodniczący Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Kaczyński! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt tej ustawy sankcjonuje bezprawie. Nielegalne zawracanie ludzi na granicy ogranicza ich prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, jest sprzeczne z konwencją genewską i z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, a co za tym idzie, jest niezgodne z naszą konstytucją. Cudzoziemcowi, który na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi. Wiem, że większość rządu uważa łamanie konstytucji za świetną zabawę, a nieprzestrzeganie umów międzynarodowych za patriotyczny obowiązek, jednak łamanie praw człowieka, w tym praw mniejszości i cudzoziemców, stało się dla was główną rozrywką.

Oto SMS-y znad granicy: Prosimy o pomoc. Strzelili do mnie, kilka centymetrów od mojej stopy, bardzo nas pobili.

Wysoka Izbo!

W ustawie wprowadzacie mechanizm, który de facto uniemożliwi odwoływanie się uchodźców od decyzji Straży Granicznej. Po pierwsze, chcecie, by odwoływać się oni mogli tylko do komendanta Straży Granicznej. Zupełnie ignorujecie prawo do odwołania się np. do sądu. To oznacza, że naruszona będzie zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, a proponowane zmiany są niezgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jako Lewica zgłaszamy poprawki dające możliwość odwołania się do sądu, a także możliwość oczekiwania na wyrok niezawisłego sądu na terytorium Polski.

Wysoka Izbo! Mam kilka pytań.

Dlaczego nie ufacie swoim własnym służbom?

Szczęść Boże służbie granicznej, policjantom i żołnierzom, którzy w tej sprawie robią to, co do nich należy. Czy ja dobrze słyszałem, że powiedział, że zajmuje się przeprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnych imigrantów? Proszę, panie ministrze, o wyciągnięcie wniosków operacyjnych i prawnych. Pytanie jest takie: Kiedy, a może już, zajmiecie się poważnie formatowaniem prawnym moratorium imigracyjnego? To dobrze.

Chciałem odpowiedzieć panu posłowi Braunowi na to, myślę, haniebne oskarżenie o pomoc w jakimś nielegalnym procederze. Nielegalne jest to, że ci ludzie, owszem, przekroczyli granicę, ale są skazywani bez sądu i wywożeni do lasu bez procedury. Nie można karać nikogo bez sądu.

Debatujemy dziś nad nowelizacją ustawy, która ma pozwolić na przyspieszoną deportację imigrantów za naszą wschodnią granicę. Oczywiście należy chronić nasze granice, co do tego nikt nie ma wątpliwości, zwłaszcza że oczywiste jest, co robi Łukaszenka i jakie ma zamierzenia. Ale dlaczego robicie to w tak nieudolny sposób? Gdzie humanitaryzm? Wprowadzacie stan wyjątkowy, pospiesznie dodajecie przepisy do ustawy o cudzoziemcach pozwalające na zawracanie emigrantów. Robicie pokazówkę w Usnarzu Górnym. Chciałam się zapytać, gdzie jest minister do spraw bezpieczeństwa pan Kaczyński. Przede wszystkim powinien tutaj dzisiaj siedzieć i słuchać naszej debaty. Drugie pytanie: Ilu nielegalnych imigrantów przekroczyło granicę Polski w tym roku?

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy, który procedujemy - myślę, że warto to przypomnieć - to próba dostosowania prawa krajowego do aktualnej, niezwykle trudnej sytuacji imigracyjnej, którą mamy na granicy z Białorusią. Państwo polskie mierzy się dziś z ogromnym problemem na naszej granicy i niestety - mówię to z ogromnym smutkiem - opozycja w znacznej części głosując przeciw temu projektowi, szkodzi bezpieczeństwu Polaków. Brak tych regulacji, które rząd proponuje, to ograniczenie skuteczności naszych służb, a przede wszystkim Straży Granicznej. Przypominam, że ten projekt ustawy zawiera rozwiązania mające służyć przeciwdziałaniu nadużywania instytucji ochrony międzynarodowej, która jest wykorzystywana przez ludzi, którzy naprawdę źle życzą Polsce i Polakom. I moje pytanie do pana ministra: Jak brak tej nowelizacji, tej zmiany przepisów wpłynąłby na bezpieczeństwo Polaków? Pan poseł Tomasz Szymański, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek przyszło się mierzyć Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji z tak kiepskim, z tak złym pomysłem, projektem. On jest tak zły, że nawet nazwa projektu nie jest zgodna z jego treścią. Na samym końcu zrobiliście państwo autopoprawkę, zmieniając całkowicie kształt ustawy, wprowadzając jakieś kolejne obostrzenia, kolejne rzeczy. Szanowni Państwo! Nie ma takiej możliwości, żebyście nie mogli państwo skorzystać z aktualnych norm i przepisów prawnych, które miałyby pełne zastosowanie do tego projektu i do tej sytuacji, jaką mamy na granicy. Ten projekt jest tak zły, że nie ma chyba żadnej instytucji, ani żadnej instytucji prawnej, która by powiedziała, że cokolwiek może być w nim dobrego. Biuro Legislacyjne Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych. Komisarz do spraw unijnych powiedział jednoznacznie, że łamiecie wszelkie standardy i procedury prawne powszechnie obowiązujące. Zastanówcie się państwo nad tym, ponieważ my również chcemy pomóc i doprowadzić wspólnie do takiej sytuacji, żeby naród polski i Polacy czuli się bezpiecznie. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Rzadko zdarza się, żeby jeden projekt ustawy łamał jednocześnie tyle traktatów międzynarodowych, dyrektyw prawa europejskiego, polską konstytucję - wszystko na dwóch stronach. On łamie zapisy konwencji genewskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, dwóch dyrektyw unijnych, polskiej konstytucji. Miażdżącą krytykę przedstawili do tego prawie wszyscy: Biuro Legislacyjne, prawnicy, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce. Te organizacje przedstawiły też rozwiązania, jak tę sytuację można rozwiązać dzisiaj w ramach prawa. W skrócie: ta ustawa to czyste bezprawie i dlatego nigdy nie będzie skuteczna. A przecież sytuacja na granicy jest paląca. Narastająca presja migracji dziś - przez wojnę hybrydową Białorusi i Rosji, a za chwilę, i w tle, przez kryzys klimatyczny. Ta sytuacja nie odejdzie.

Wysoka Izbo! Ochrona granic, bezpieczeństwo naszego kraju to nasza, polityków, odpowiedzialność. To nie budzi wątpliwości ani sporu. Pamiętajmy jednak, że stanowiąc prawo, nie możemy tego prawa łamać, a tak właśnie czyni polski rząd, proponując taką zmianę przepisów, o których wiemy już dziś na podstawie wcześniejszych dotychczasowych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że są z tym prawem niezgodne. Ile polskie państwo zapłaci w ramach przyszłych odszkodowań? Czy nie uważają państwo, że należałoby to uwzględnić w skutkach finansowych niniejszego projektu? Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wiele słów już padło na temat uchodźców, każda ze stron ma swoje racje i pewnie pozostaniemy przy swoich.

Apeluję, żeby ewentualnie, jeżeli pojawią się jakiekolwiek zarzuty, to żeby były kierowane do ministrów, do premiera, a nie do żołnierzy, nie do Straży Granicznej, którzy bronią naszego kraju, granicy Schengen, granicy europejskiej. Proszę o rozwagę i powstrzymywanie się przed jakimikolwiek powiedzeniami, które mogłyby obrazić pograniczników czy żołnierzy. Dziękuję, panie pośle. Wysoka Izbo! Rozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie naszego kraju. Miałem taką nadzieję, że posłucham czegoś mądrego od opozycji. Niestety ze smutkiem muszę powiedzieć, że państwo nas nie zawiedliście, nic mądrego żeście nie powiedzieli, nic dobrego dla naszego kraju. Ale to jest formuła pytań, w związku z tym mam takie pytanie. Panie ministrze, czy ta ustawa w ogóle by była potrzebna, gdybyśmy mieli inną opozycję, mądrzejszą? I jeszcze jedna kwestia, ponieważ mówiliśmy o łamaniu prawa, pan poseł Braun o tym mówił: Czy prawdą jest, że pan Konieczny wielokrotnie przekraczał nielegalnie granicę polsko-białoruską? Czy wobec niego zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje? Ponieważ mówiliśmy tutaj o działaniach innego posła, w związku z tym to jest właśnie to pytanie: Czy przez takie nieodpowiedzialne zachowanie chociażby Franka od Sterczewskich czy Klaudii od Jachirów można by było założyć taką sytuację, że to oni by dostali jakąś kolbą od białoruskiego (Dzwonek) pogranicznika w oczy? Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przywoływałem dzisiaj fakt wypowiedzenia umowy o readmisji przez Białoruś Unii Europejskiej, która przewiduje, że nielegalny imigrant i uchodźca zatrzymany w Polsce jest odsyłany do kraju, z którego przybył, w tym przypadku chodzi oczywiście o Białoruś. Stąd też moje pytanie: Skoro nie można zawrócić takich uchodźców na Białoruś, to gdzie państwo ich odeślecie? Na jakich zasadach? W jakim trybie? Jak ta procedura miałaby przebiegać, skoro też wielokrotnie wiemy, że takie osoby nie posiadają dokumentu tożsamości, a jednocześnie wiemy, że procedura związana z ustaleniem tożsamości musi chwilę potrwać. W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi: W jakim trybie, w jakim czasie państwo chcecie to przeprowadzić w nawiązaniu do ustawy, którą dzisiaj procedujemy? Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na pytania odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan minister Maciej Wąsik.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Padło tutaj wiele tez, wiele pytań, wiele zarzutów.

Otóż chciałem pani odpowiedzieć, że jeżeli są uchodźcami, to pierwszą granicę w myśl konwencji genewskiej mogą przekroczyć bezprawnie. Pierwszą z kraju, z którego grozi im niebezpieczeństwo. Każda następna granica powinna być przekraczana zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i prawa obowiązującego chociażby w Polsce. Czyli tych ludzi obowiązują polskie przepisy, jeżeli są uchodźcami. Ale czy są uchodźcami? Proszę mi odpowiedzieć, pani poseł. Co grozi Egipcjanom w Egipcie? Owszem, znajdują się tam także Afgańczycy albo ludzie, którzy podają się za Afgańczyków. Tylko proszę też pamiętać, że to nie są ludzie, którzy uciekali przed talibami na lotnisku w Kabulu. To nie są ludzie, którzy stanowili trzon państwa afgańskiego, którym grozi w Afganistanie niebezpieczeństwo. Pytanie czy uciekli, czy wyemigrowali w celach zarobkowych albo socjalnych. I powiem jeszcze pani tak, że my, Straż Graniczna widzimy ich drogę do Polski samolotami białoruskich linii lotniczych z Bagdadu, z Turcji, ale także często przez Moskwę. Doskonale widzimy tę drogę, widzimy zdjęcia w ich telefonach i wiele innych rzeczy. Jakie mają prawo? Mają prawo przebywać na terenie Białorusi, bo mają białoruskie wizy, bo przybyli jako turyści na Białoruś. Czy są nieszczęśliwi? Tak, są nieszczęśliwi.

Szanowni państwo, tak, to są ludzie nieszczęśliwi, ale to nie są uchodźcy, to są ludzie oszukani przez Łukaszenkę, bo to są ludzie, którzy często sprzedali majątki albo wzięli oszczędności swoich klanów po to, żeby kupić za wiele tysięcy dolarów bilet do Mińska. I oni teraz mówią do naszych pograniczników: Odwieźcie nas do Bagdadu. My się policzymy z tymi, którzy sprzedali nam te bilety. Szanowni Państwo! Polska wielokrotnie udzielała pomocy uchodźcom: i tym, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebowali, i tym, którzy uciekali z krajów, gdzie groziło im niebezpieczeństwo. Wszyscy pamiętamy rządy, które pomagały Czeczeńcom. Tak że teraz czuliśmy się w obowiązku moralnym pomóc wszystkim Afgańczykom, którzy współpracowali z polską dyplomacją, z polskim kontyngentem wojskowym, w przypadku których pozostanie w Kabulu groziło śmiercią, torturami, więzieniem. Przywieźliśmy ich do Polski.

Oni to wszystko dostaną w Polsce, ale to są uchodźcy.

I powiedziała tak: Spójrzmy na sytuację na granicy Unii Europejskiej z Białorusią. Reżim w Mińsku użył ludzi do swych celów, załadował ich do samolotów i dosłownie wypchnął na granicę z Unią. Nie możemy tego tolerować. Stąd szybka reakcja Unii na tę sytuację. Zapewniamy państwa, że będziemy nadal wspierać Litwę, Łotwę i Polskę. Nazwijmy to po imieniu. Jest to hybrydowy atak mający na celu destabilizację Europy. To są słowa szefowej Komisji Europejskiej.

Zakończyło się to klęską tej polityki. Szanowni Państwo! Ustawa, o której mówimy, w przypadku gdy cudzoziemiec został zatrzymany niezwłocznie po przekroczeniu granicy wbrew przepisom, daje możliwość komendantowi Straży Granicznej sporządzenia protokołu przekroczenia granicy oraz wydania zarządzenia o przekroczeniu granicy wbrew przepisom prawa. W postanowieniu zostanie określony nakaz opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zakaz, wraz z określeniem okresu obowiązywania, ponownego wjazdu na teren, na terytorium Rzeczypospolitej i innych obszarów Schengen. I chciałem państwu powiedzieć, że zastosowanie powyższego rozwiązania umożliwia przepis art. 2 ust. 2 lit. a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/115/WR z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawach wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, która przewiduje, że państwo członkowskie może jej nie stosować do obywateli państw trzecich, którzy zostali zatrzymani lub ujęci przez właściwe organy w związku z nielegalnym przekroczeniem lądowej, morskiej lub powietrznej zewnętrznej granicy tego państwa członkowskiego oraz którzy nie otrzymali następnie zezwolenia na pobyt lub prawa do pobytu w tym państwie członkowskim.

To nie jest uzasadnienie.

Szanowni Państwo! Jeżeli cudzoziemiec przekracza - muszą tu być spełnione dwa warunki równocześnie - granicę Polski w sposób nielegalny, czyli zieloną granicę, a jednocześnie jest to granica z państwem, w którym nie grożą mu śmierć, tortury, więzienie, wówczas szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który rozpatruje wniosek o udzielenie pomocy, może - nie musi, ale może - pozostawić ten wniosek nierozpatrzony, bez rozpatrzenia, właśnie dlatego, że jest to notorycznie nadużywana procedura. Jeżeli uzna, że są jednak przesłanki udzielenia pomocy tej osobie, taka pomoc może być udzielona. Chciałem powiedzieć tak. Usłyszałem tutaj wiele słów o łamaniu różnych wyroków, traktatów, przepisów, o łamaniu praw obywateli obcych państw, którzy gdzieś się tam nagle znajdują. Dlaczego nie słyszę od was żalu, że ktoś łamie polskie prawo, że ktoś przekracza polskie granice, polską granicę? Nie widzicie prawa Polaków do spokojnego życia na swojej ziemi, do ochrony granic? My jako rząd będziemy to prawo realizować konsekwentnie, ale także będziemy udzielać pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują, mądrze i rozsądnie. Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Odpowiedzi na pytania udzieli również sprawozdawca komisji pan poseł Zdzisław Sipiera. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Jeden to jest aspekt humanitarny. Tu, proszę państwa, nie ma zagrożenia, że Polska nie przestrzega elementów humanitarnych i tego nigdzie, w żadnym elemencie nie ma, natomiast jest to, co dzisiaj dokładnie, a państwo często powołujecie się na te aspekty, które wypowiada Komisja Europejska. Słowa, które cytował dzisiaj minister Wąsik, są adekwatne. To właśnie te słowa mówią w ten sposób: to Polska jest w tym momencie na tym etapie, w tym miejscu i w tej sytuacji formalnoprawnej, że trzeba jej pomóc. To właśnie Komisja Europejska nam mówi. Jak mamy to zrobić? Jeszcze otwierając bardziej granicę? Jeszcze stosując te przepisy, które będą zabawą w kotka i myszkę? I to, co było podkreślane, już eliminując aspekty personalne, ale pytania pana posła Brauna, czy poseł nie przekracza granicy. Czy to są rzeczy poważne, czy niepoważne? Proszę państwa, od tego nie jest poseł, od tego jest Straż Graniczna. Panie Pośle! Jeżeli my nie przestrzegamy jako posłowie prawa, które jest w Polsce, to o czym mamy mówić. Bardzo proszę, jutro będą dalsze prace i te wnioski, które, widzę, otrzymałem jako sprawozdawca, które mówią w ogóle o odrzuceniu w drugim czytaniu tej ustawy, to absolutnie nie idzie w tym kierunku, żeby zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa Polski, a raczej odwrotnie - zmniejszenie.

Żeby opozycja pokazała, że jest to jednak interes państwa polskiego i interes Unii Europejskiej, tak żebyśmy mogli nad tą ustawą procedować i ją przegłosować, żeby weszła w życie. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, by Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych celem przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia świętego Maksymiliana Kolbe w 80. rocznicę śmierci (druki nr 1452 i 1500) Uprzejmie proszę panią poseł Dominikę Chorosińską o przedstawienie sprawozdania komisji.

Pani Marszałek! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Kultury i Środków przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia świętego Maksymiliana Kolbe w 80. rocznicę śmierci. Posłem wnioskodawcą był już w tej chwili minister Tomasz Rzymkowski. Marszałek Sejmu skierowała ten projekt do komisji kultury. Komisja kultury w dniu 11 sierpnia przeprowadziła pierwsze czytanie oraz rozpatrzenie tego projektu uchwały. Projekt został uchwalony przez komisję bez głosu sprzeciwu i w finale uzyskał on następującą treść: „Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w 80. rocznicę śmierci.

Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli. Pochodził z rodziny, która zajmowała się tkactwem, a jego przodkowie byli emigrantami z Czech. W kościele w Pabianicach odnalazł powołanie do służby Bogu i człowiekowi. Po uzyskaniu doktoratu w Rzymie potrafił odnaleźć modus vivendi z władzami Japonii, by z wielkim sukcesem prowadzić działalność duszpasterską i misyjną w Nagasaki. Był założycielem ruchu Rycerstwo Niepokalanej, miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” oraz Radia Niepokalanów. Wyprzedził swoje czasy, doceniając rosnącą rolę mediów w kształtowaniu zasad życia społecznego opartego na wartościach chrześcijańskich. Od pierwszych dni II wojny światowej ten święty Kościoła katolickiego zgodnie z duchem franciszkańskim otworzył bramy klasztoru w Niepokalanowie dla uciekinierów, chorych i głodnych, zarówno dla chrześcijan, jak i Żydów. Ratując ojca rodziny - Franciszka Gajowniczka, złożył w ofierze swoje życie w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. W 80. rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając jego zasługi dla narodu polskiego oraz świadectwo miłości bliźniego, oddaje hołd męczennikowi oraz składa cześć jego pamięci” Komisja wnosi o uchwalenie powyższej uchwały. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Tomasz Rzymkowski. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym odnieść się do projektu uchwały. Jest mi trochę niezręcznie, gdyż jestem autorem tej uchwały. Św. Maksymilian Maria Kolbe jest nam wszystkim doskonale znany.

Był osobą duchowną, franciszkaninem, założycielem i twórcą największego klasztoru franciszkańskiego na świecie. Był również misjonarzem. Osiągnął to, co wielu franciszkanom się nie udało, czyli na stałe stworzył klasztor w słynnym z zupełnie innej przyczyny japońskim Nagasaki. Był również, co jest mało znane, autorem słowa, które pojawiło się za jego sprawą w języku japońskim, słowa: miłosierdzie. Ale oprócz tego, że był człowiekiem oddanym Bogu i drugiemu człowiekowi, był również, co z tego wynika, człowiekiem niezwykle oddanym bliźniemu. To piękne serce, które okazywał przez całe życie bliźnim poprzez troskę o ład moralny, troskę o rodzinę, najlepiej uzewnętrznia jego działanie podczas II wojny światowej, kiedy otworzył, tak jak to w uchwale zostało zawarte, bramy klasztoru w Niepokalanowie dla prześladowanych Polaków, ale również dla naszych współobywateli, naszych braci Żydów, za co został aresztowany i wysłany do symbolu niemieckiego totalitaryzmu, niemieckiego narodowego socjalizmu, do obozu zagłady Auschwitz, gdzie oddał życie za współwięźnia. Znaczy, dał to, co dla nas ludzi jest najcenniejsze, czyli oddał własne życie.

Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo, panie ministrze. W imieniu Koalicji Obywatelskiej głos zabierze pan poseł Wojciech Król. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zacznę od przypomnienia papieskich wizyt w byłym niemieckim obozie masowej zagłady Auschwitz-Birkenau, gdzie męczeńską śmiercią zmarł 80 lat temu o. Maksymilian Kolbe.

Karol Wojtyła wychował się i dorastał niedaleko Oświęcimia, był świadkiem wojny i niemieckich zbrodni. Wojna i jej okrucieństwa stały się czymś w rodzaju fundamentu jego późniejszego pontyfikatu.

Zdjęcia, kiedy przechodzi przez słynną bramę, obiegły świat. W miejscu takim jak to brakuje słów, a w przerażającej ciszy serce woła do Boga: Panie, dlaczego milczałeś? Dlaczego na to przyzwoliłeś?” - mówił niemiecki papież. 29 lipca 2016 r. papież Franciszek szedł samotnie drogą, którą przemierzyli jego dwaj poprzednicy. Papież, który ma niesamowity dar rozmowy, wybrał milczenie. Modlił się w ciszy. Milcząc, powiedział wszystko. W milczeniu Franciszek modlił się w celi śmierci o. Maksymiliana Kolbego. Ta wizyta odbyła się w dniu, w którym przypadła 75. rocznica apelu, kiedy o. Kolbe ofiarował swoje życie za współwięźnia.

Ojciec Maksymilian Kolbe, człowiek, który z otwartymi rękami witał uciekinierów, ewangelicznych głodnych i spragnionych, który z troską pochylił się nad ich losem, który przyjmował po bratersku chrześcijan i Żydów, umierał w ciszy śmiercią głodową, bo na taką śmierć skazali go oprawcy. Umierał w największej fabryce śmierci stworzonej przez ludzką nienawiść, w miejscu otoczonym ogrodzeniem z drutu kolczastego. W naszym kraju drut kolczasty jest wyjątkowym symbolem, symbolem okrucieństwa, opresji i cierpienia. Koalicja Obywatelska opowiada się (Dzwonek) za przyjęciem uchwały upamiętniającej 80. rocznicę śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Na koniec dodam, że mój syn 3 lata temu właśnie otrzymał imię Maksymilian. Dziękuję bardzo, panie pośle. Wysoka Izbo! Maksymilian Kolbe, a właściwie Rajmund Kolbe, to polski duchowny, którego znamy przede wszystkim z jego bohaterskiego czynu, czyli oddania życia za współwięźnia z obozu Auschwitz, skazanego na śmierć głodową Franciszka Gajowniczka, co oznaczało, że to Kolbe zginął w bunkrze głodowym dobity zastrzykiem z fenolu. Wielki heroiczny czyn, na który stać niewielu, niewątpliwie godny upamiętnienia. Rajmund Kolbe pochodził z ziemi łódzkiej. W 1910 r. wstąpił do zakonu franciszkanów i wtedy przyjął imię Maksymilian. Studiował m.in. w Rzymie, gdzie założył Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej. Po powrocie do Polski założył klasztor, wydawnictwo Niepokalanów i radio Niepokalanów.

Niestety oba te pisma pełne były antysemickich treści. Żydom zarzucano światowy spisek, demoralizację Polaków, propagowanie rozwodów i pornografii, postulowano ograniczenie im edukacji wyższej, wysyłano do Palestyny. Dla Kościoła katolickiego Kolbe miał oczywiście wielkie zasługi. Został beatyfikowany, a potem uznany za świętego. Dziś w Sejmie debatujemy nad uchwałą upamiętniającą, jak to sformułował wnioskodawca, 80. rocznicę śmierci św. Maksymiliana Kolbego. Język, którym uchwała jest napisana, tak jak jej tytuł, jest językiem Episkopatu Polski. Wnioskodawca, minister w rządzie PiS-u pomylił porządki i instytucje. Bo Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który reprezentuje nie tylko Polaków katolików, powinien honorować nie kościelnego świętego, tylko obywatela Rajmunda Maksymiliana Kolbego za to, że uratował życie innemu człowiekowi. A posłowie polskiego Sejmu powinni pytać, jaki wpływ miały antysemickie treści, które docierały do milionów Polek i Polaków przez media, którymi kierował zakonnik Maksymilian Kolbe. Czy te nienawistne treści nie przyczyniły się do takich tragedii jak wojenne denuncjacje lub powojenne pogromy nie tylko w Jedwabnem, których dokonali Polacy katolicy na Polakach wyznania mojżeszowego?

Dziękuję bardzo. Pani poseł, pani już skończyła. Pani poseł, proszę opuścić mównicę. Pani poseł, dość tego. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pozwólcie państwo, że rozpocznę od słów, które wszyscy katolicy pewnie znają: bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Urodził się, tak jak było powiedziane, szanowni państwo, 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W wieku 16 lat wstąpił do zakonu franciszkanów we Lwowie i otrzymał imię Maksymilian. Następnie pojechał do Rzymu, gdzie uzyskał doktoraty z filozofii, teologii. W 1917 r. założył tam Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Polski w 1919 r. założył pod Warszawą klasztor w Niepokalanowie oraz zaczął wydawać pismo „Rycerz Niepokalanej” Sukcesy odniesione w Polsce nie zadowoliły zakonnika. Chcąc zdobyć cały świat dla Niepokalanej, wyjechał w 1930 r. na misję do Chin, a potem do Japonii. Mimo że nawet niektórzy jego bracia uważali, że wyprawa na Daleki Wschód to szaleństwo, ojciec Kolbe stworzył w Nagasaki drugi Niepokalanów. Wydawał japoński odpowiednik „Rycerza Niepokalanej” oraz założył nowicjat i seminarium. W 1936 r. zakonnik wrócił do Polski, gdzie później zastała go II wojna światowa. Został aresztowany przez gestapo, był przesłuchiwany na Pawiaku.

Chciał w nich wzbudzić wolę życia i przetrwania, wspominał jeden z ocalonych więźniów. Do swoich towarzyszy mówił: ufajcie Niepokalanej, wy, młodzi, żyć będziecie, ja obozu nie przeżyję, ale wy będziecie uratowani.

Swoją decyzję uzasadniał wtedy tak: Mam już blisko 50 lat, życie moje przeżyłem, a ten ma życie przed sobą, ma żonę i dzieci. Zaskoczonemu Niemcowi, który pytał, dlaczego chce pójść na śmierć za obcego człowieka, odpowiedział: Chcę innym dodać odwagi do życia.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Krzysztof Tuduj w imieniu koła Konfederacja.

Wysoka Izbo! Św. Maksymilian Maria Kolbe to postać wybitna, wielki wzór do naśladowania. Człowiek, który pokazał, jak wielką siłę można czerpać z wiary i wierności zasadom katolickim. Św. Maksymilian chciał podbić świat dla Maryi, chciał podbić świat miłosierdziem, wyrugować z ludzkich serc nienawiść oraz wszelkie zło. Dzięki swojej determinacji założył największy w historii Polski religijny miesięcznik, stworzył też największy klasztor na świecie, klasztor w Niepokalanowie. Nigdy jednak nie opływał w bogactwa i prowadził bardzo skromne, ascetyczne życie. Pieniądze przeznaczał na rozwój medialnego imperium miłosierdzia. Swoim zasadom pozostał wierny do końca i nie odrzucił ich nawet w obliczu tortur i upokorzeń. Nieustannie pocieszał innych osadzonych i zachęcał do modlitwy. Gdy esesmani wybierali więźniów, którzy mieli trafić do celi i umrzeć śmiercią głodową, św. Maksymilian, choć nie został wybrany, wstawił się za innego więźnia i oddał za niego życie. Wspomniany więzień był bowiem żonaty, a Maksymilian nie chciał, żeby osierocił dzieci. Wolał sam oddać życie w męczarniach, by uratować obcego człowieka. Jestem księdzem katolickim, jestem stary, chcę umrzeć za niego, on ma żonę i dzieci - powiedział do niemieckiego esesmana, który przystał na jego prośbę. Maksymilian Kolbe do samego końca w celi głodowej pocieszał umierających wraz z nim więźniów. Do końca służył im, wyspowiadał wszystkich chętnych oraz podnosił na duchu w taki sposób, że ci byli jeszcze zdolni śpiewać radośnie katolickie pieśni.

Przychylamy się do uczczenia św. Maksymiliana Kolbego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Tu, w Sejmie, w kaplicy, która - no cóż, taka to była epoka kompromisu dziejowego - ma rozmiar nieco tylko większy od składziku na szczotki, pojawiły się z końcem ubiegłego roku relikwie św. Maksymiliana. Informuję o tym koleżanki i kolegów. Cieszę się, że jest jakiś kamień węgielny polskiego parlamentaryzmu, który na co dzień, rzecz jasna, nie dorasta do takich wzorców. Tak bardzo nie dorasta, że zdaje się to aż wręcz świętokradcze, że w ogóle przyzywamy tutaj imienia tego świętego. Oby taki moment mimo wszystko, mimo pewnych ekscesów (Dzwonek) i popisów ignorancji i pewnego zjednoczenia w tej sali, zostawił jakiś trwały ślad w naszej pracy. Oby to była nowa karta odkryta w historii tej kadencji, a zatem może zwiastująca jakąś lepszą przyszłość dla nas niegodnych i dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysoka Izbo! Bardzo proszę, panie pośle, bo koleżanki zajmują pana czas, a czas płynie. W chwili obecnej jest to jeden z kilku polskich profili z liczbą obserwujących większą niż 1 mln. Ten profil publikuje tylko zdjęcia. To są zdjęcia więźniów obozu w Oświęcimiu. Każde z tych zdjęć jest dowodem na tragedię tych ludzi, na tragedię każdego bohatera tych zdjęć. Maksymilian Kolbe, patron ziemi oświęcimskiej, jest dla mnie symbolem. Był jednym z wielu, którzy odnieśli zwycięstwo w miejscu, w którym miłość nie miała szans wobec nienawiści. A nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Pragniemy ogarnąć uczuciem najgłębszej czci każde z tych zwycięstw, każdy przejaw człowieczeństwa (...) na miejscu tak straszliwego podeptania człowieczeństwa, godności ludzkiej - zwycięstwo człowieka.

Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Oczywiście Maksymilian Maria Kolbe był postacią, która wykazała się wielkim heroizmem, i co do tego, że jest osobą godną naśladowania, nie mamy, jak myślę, wątpliwości.

Otóż kiedy czytam tę uchwałę, to mam takie poczucie, że ona stoi w swoim przesłaniu bardzo daleko od tego, co na co dzień widzimy w działaniach wnioskodawców. Przed chwilą omawialiśmy też projekt takiej ustawy, która może nawiązywać do tej uchwały.

Bardzo proszę.

i wykrzykują inwektywy, insynuacje pod adresem człowieka, który dobrotliwie pewnie mimo wszystko popatruje na to z nieba i wstawia się także i za swoimi potwarcami. Ale pytanie jest takie: Czyście czytały, czcigodne panie, którykolwiek z tekstów pomieszczonych na łamach czasopism wydawanych, publikowanych przez św. Maksymiliana?

Pani poseł, pani poseł, pani poseł. Lista posłów zapisanych. Ale dlaczego pani krzyczy, pani poseł? Dlaczego pani krzyczy?

Zamykam dyskusję. Do głosowania nad projektem uchwały przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Przemysława Krycha reprezentowanego przez adwokatów Karinę Aust-Niewiadomską oraz Krzysztofa Sajchtę z dnia 3 stycznia 2019 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Marty Golbik (druk nr 1421) Uprzejmie proszę pana posła Kazimierza Smolińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Przemysława Krycha reprezentowanego przez adwokatów Karinę Aust-Niewiadomską oraz Krzysztofa Sajchtę z dnia 3 stycznia 2019 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Marty Golbik. Marszałek Sejmu na podstawie art. 7c ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora skierowała w dniu 30 stycznia 2019 r. powyższy wniosek do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w celu rozpatrzenia. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, po rozpatrzeniu tego wniosku na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2021 r., na podstawie art. 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora przedkłada propozycję odrzucenia wniosku oskarżyciela prywatnego Przemysława Krycha z dnia 3 stycznia 2019 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Marty Golbik. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przypominam, że Sejm, zgodnie z art. 133 ust. 6 regulaminu Sejmu, rozpatruje sprawozdanie komisji, wysłuchując jedynie sprawozdawcy. Prawo do zabrania głosu przysługuje również posłowi, którego wniosek dotyczy. Nad sprawozdaniem tym nie przeprowadza się dyskusji. Ponieważ pani poseł nie wyraziła zainteresowania zabraniem głosu, do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Przemysława Krycha reprezentowanego przez adwokatów Karinę Aust-Niewiadomską oraz Krzysztofa Sajchtę z dnia 3 stycznia 2019 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Urbaniaka (druk nr 1422) Uprzejmie proszę pana posła Kazimierza Smolińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Przemysława Krycha reprezentowanego przez adwokatów Karinę Aust-Niewiadomską oraz Krzysztofa Sajchtę z dnia 3 stycznia 2019 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Urbaniaka.

Komisja po rozpatrzeniu tego wniosku na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2021 r. na podstawie art. 7c ust. 5 ww. ustawy przedkłada propozycję odrzucenia wniosku oskarżyciela prywatnego Przemysława Krycha z dnia 3 stycznia 2019 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Urbaniaka. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przypominam, podobnie jak w poprzednim punkcie, że Sejm, zgodnie z art. 133 st. 6 regulaminu Sejmu, rozpatruje sprawozdanie komisji, wysłuchując jedynie sprawozdawcy. Prawo do zabrania głosu przysługuje również posłowi, którego wniosek dotyczy. Nad sprawozdaniem tym nie przeprowadza się dyskusji. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 15 września br. Informuję, że zgłosili się posłowie celem wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Skoro nikt się nie zgłasza, listę posłów zgłoszonych do oświadczenia uważam za zamkniętą. Bardzo proszę, panie pośle.

Bardzo dziękuję, naprawdę wzruszona jestem do łez. Nie ma. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Światowy Dzień Sybiraka. Co roku 17 września w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Obchody zostały zorganizowane przez Związek Sybiraków, czyli polską organizację grupującą byłych zesłańców, którzy nazywają siebie sybirakami. Od 2013 r. Światowy Dzień Sybiraka ma status święta państwowego. W 2013 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie podjęto przez aklamację. Najważniejsze w tym dniu jest przypominanie prawdziwych losów zesłańców, spisywanie przekazów żyjących osób i przekazywanie ich dalej. Jest to współczesny hymn Związku Sybiraków. Autorem tekstu jest Marian Jonkajtys, sybirak, a kompozytorem Czesław Majewski. Tylko minuta? Tekst opiewa historię i męczeństwo Polaków, którzy przymusowo zostali zesłani na Syberię. Przytoczę jego tekst: „Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, Z rezydencji, białych dworków i chat Myśmy wciąż do Niepodległej szli, Szli z uporem, ponad dwieście lat!

I nam w marszu do Polski przewodził.

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, Szkół, urzędów i kamienic i chat: Myśmy znów do Niepodległej szli, Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat. Bo od września, od siedemnastego, Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas: Przez lód spod bieguna północnego, Przez łubiankę, przez Katyński Las! Na nieludzkiej ziemi znów polski trakt Wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat. Bo przed nami Polska - coraz bliżej! I myśmy szli i szli - dziesiątkowani! Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez Ludową przeszliśmy - niepokonani Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg! Pamiętajmy o sybirakach nie tylko w tym dniu. Wspominajmy tych, których nie ma już wśród nas. Wszystkim sybirakom już dzisiaj życzę zdrowia, radości i wielu pomocnych dłoni każdego dnia. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeszcze niedawno, bo w ubiegłym roku, w składzie Rady Ministrów funkcjonowało samodzielne ministerstwo sportu z ministrem sportu równym rangą innym ministrom. Niestety z historii naszej państwowości wynika, że jeżeli coś dobrze działa, ale nie da się do końca tym czymś sterować, to nie przetrwa to długo i skończy tak, jak np. skończyły polskie stadniny albo tak jak skończyła się kluczowa pozycja Polski w Unii Europejskiej.

Ministerstwo sportu było dla pana premiera za mało narodowe. Co może bardziej cieszyć każdego narodowego premiera niż kolejna narodowa reorganizacja? Narodowa reorganizacja dla narodowej reorganizacji tak bardzo wciągnęła pana premiera, że do dzisiaj polscy sportowcy nie mają ani własnego ministerstwa, ani żadnego narodowego centrum, a sprawy sportu wciśnięto na siłę ministrowi kultury, który najzwyczajniej w świecie się po prostu na tym nie zna. Spraw sportu musi bronić minister sportu. Dobrze radziła sobie z Ministerstwem Sportu pani minister Danuta Dmowska-Andrzejuk. Dlaczego ktoś wpadł na pomysł, żeby ją z tej funkcji zwolnić, a ministerstwo rozwalić? Nie wiem, ale wiem, że nie było to dobre rozwiązanie. Dlatego z tego miejsca apeluję do pana premiera Mateusza Morawieckiego i do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego: Polskiemu sportowi potrzebny jest minister sportu, a nie wieczny sportowy chaos narodowy, w którym jesteśmy w czołówce. Macie, panowie premierzy, kadry menadżerskie, macie pieniądze, zróbcie panowie w tej kwestii to, co się polskiemu sportowi należy. Dziękuję bardzo. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Pan poseł Władysław Kurowski, Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chciałbym z tego miejsca przedstawić jedną z wielu historii mojego regionu z okresu niemieckiej okupacji, historię, która już na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców, rodzin i całej społeczności lokalnej, a jej upamiętnienie to także mój obowiązek. W tej miejscowości powiatu myślenickiego w 1943 r. odbyła się krwawa i okrutna pacyfikacja, w wyniku której na tzw. bydlęcym rynku i w plebańskiej stodole zamordowano 26 osób - mieszkańców Sułkowic i Harbutowic. Akcja pacyfikacyjna została starannie zaplanowana i przygotowana przez okupanta niemieckiego. Według świadków na terenie Sułkowic było wówczas od 2 do 3 tys. żołnierzy. Duża liczba żołnierzy mogła świadczyć o tym, że Niemcy bali się interwencji oddziałów partyzanckich, które były rozlokowane w pobliskich lasach.

Oddziały pacyfikacyjne nadjechały do Sułkowic równocześnie ze wszystkich stron. Około godz. 4 rano zaczęto wypędzać ludzi z domów. Po odszukaniu osób z tzw. czarnej listy dokonywano ich aresztowań. Na rynku hitlerowcy rozpoczęli przygotowania do przesłuchań. Z całej wsi grupami prowadzono mieszkańców w stronę centrum, na rynek bydlęcy. Pełną szerokością drogi przesuwał się tłum ludzi otoczony szczelnym kordonem uzbrojonej żandarmerii. Przez cały czas ludzie byli popychani, bici i wyśmiewani. Widzieli, jak ich sąsiedzi są wyciągani z domów i przygotowywani do przemarszu. Żołnierze podsycali strach mieszkańców, mówiąc im z uśmiechem, że czeka ich śmierć, a cała wieś zostanie spalona, jak znajdą broń chociażby w jednym domu lub obejściu. Spędzonym na bydlęcy rynek mężczyznom kazano leżeć głową do ziemi z wyciągniętymi przed siebie rękami. Nieposłusznym groziły kary cielesne, a nawet śmierć przez rozstrzelanie. Cały bydlęcy plac zaścielony był ludźmi. Było tam ok. 3 tys. osób. Słońce paliło niemiłosiernie, ciężarne kobiety mdlały z wyczerpania. Dla nikogo nie było litości. Ludzi znajdujących się na tzw. czarnej liście gestapo prowadziło pod plebańską stodołę. Na rozkaz gestapowców wstawali i wchodzili po kolei przed niby-sąd, który zlokalizowany był w środku stodoły. Tam odbywały się bestialskie przesłuchania. Ludzie byli bici i torturowani. Później za stodołą plebańską odbyła się egzekucja osób konających i już nieżyjących. Na ofiarach wykonywano wyrok śmierci przez strzał w tył głowy.

Gestapowcy zakazali pogrzebu pomordowanych. Dopiero po wojnie, w 1945 r. ekshumowano ich ciała i uroczyście pochowano na cmentarzu parafialnym. Jego celem było wzniesienie w miejscu tragedii pomnika upamiętniającego ofiary tamtych wydarzeń, a także wszystkich mieszkańców Sułkowic, którzy zostali zabici przez gestapo, zginęli w obozach hitlerowskich lub podczas walki z okupantem. Odsłonięcie pomnika odbyło się 7 maja 1975 r., w przededniu 30. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Jakie były przyczyny pacyfikacji? Główną jednak była chęć zastraszenia mieszkańców, by pokazać, że nie warto pomagać partyzantom i walczyć o wolność. Nie można jednak traktować Sułkowic jako odosobnionego przykładu takiego bestialstwa. Pacyfikacji wsi i miasteczek w 1943 r. i w 1944 r. w Małopolsce było bardzo dużo, a wojsko niemieckie niemal wyspecjalizowało się w przeprowadzaniu takich akcji. Niech tamte wydarzenia na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pomimo wieloletniej tradycji w zakresie opieki nad zabytkami wciąż istnieje w Polsce problem niszczenia obiektów o walorach historycznych, artystycznych, a także sentymentalnych. Brak zainteresowania nimi powoduje, że ważny element naszej kultury odchodzi w zapomnienie i z roku na rok maleje szansa na ich ratunek. Trudno podać jedną przyczynę tego zjawiska. Kwestia środków finansowych nie zawsze jest tutaj kluczowa. Rodzimym przykładem takiego obiektu jest wiatrak typu holender w Krasocinie, który jest jedynym zachowanym młynem wietrznym w powiecie włoszczowskim. W województwie świętokrzyskim zachowały się dwa murowane wiatraki: jeden krasociński, drugi położony w Szwarszowicach, powiat ostrowiecki. Murowany wiatrak w Krasocinie zbudowano około 1920 r. w miejsce jego XIX-wiecznego poprzednika wykonanego z drewna, który już w czasie I wojny światowej stanowił punkt obserwacji dla wojsk austriackich i rosyjskich. W styczniu 1945 r. w trakcie ofensywy obiekt omal nie został zniszczony przez Rosjan i od tamtego czasu z roku na rok popadał w coraz większą ruinę. Taki stan był do roku 1980, w którym dzięki staraniom władz gminy Krasocin wyremontowano wiatrak, i rok później utworzono w nim Muzeum Chleba, którego pomysłodawcą był Feliks Rak. 20 lat później na skutek wichury wiatrak stracił swoje skrzydła, a regulacja jego stanu prawnego sprawiła, że przeszedł w prywatne ręce. Dopiero pod koniec 2017 r. gmina Krasocin ponownie stała się jego właścicielem, a dzięki wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków” wiatrak został zrewitalizowany. Obecnie, podobnie jak w latach 80., stanowi atrakcję turystyczną, w której mieści się Krasockie Muzeum Chleba. Obiekt w swych murach gromadzi wiele eksponatów związanych w wypiekiem chleba. Organizowane tutaj warsztaty stanowią ważny element kulturalno-edukacyjny dla najmłodszych, uczą szacunku do chleba i pracy rolników, zaś dla całych rodzin są wielopokoleniową wycieczką. Wiatrak jest swoistą wizytówką gminy Krasocin i jej symbolem. Długoletnia walka o jego ratunek przyniosła oczekiwany skutek - został ocalony od zapomnienia. Od nas zależy, jaki będzie ich los. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia obiektu, nie tylko w tym dniu. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica. Nie ma. Pan poseł Maciej Górski, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma.

Szczęść Boże wszystkim, którzy o tej późnej porze jeszcze znajdują się w tej sali, w Wysokiej Izbie! 5 minut w trybie oświadczenia poselskiego. To jedyny od miesięcy, od kwartałów moment, w którym tu czy w ogóle w przestrzeni publicznej mogę szerzej, na miarę tych skromnych możliwości, wypowiedzieć się na temat tragicznej sytuacji, w jakiej znalazły się naród polski i państwo Rzeczpospolita na skutek działań nie zaborców, nie okupantów, o których wspominał tu jeden z kolegów, przypominając tragiczne zdarzenia lat II wojny światowej. To nie agresorzy zewnętrzni, nie jakiś desant z kosmosu, to rząd, rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, władza pod flagą biało-czerwoną - bez hakenkreuza, bez sierpa i młota. Ta władza sprowadza na naród polski powszechne niebezpieczeństwo. Praktykuje to od 1,5 roku pod pretekstem walki z mniemaną pandemią, zamykając i otwierając przestrzeń publiczną, dokręcając i odkręcając śrubę, ale zawsze ze skutkami niszczącymi dla polskiego życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, także politycznego, ponieważ stopień zakłamania i hipokryzji, jaki osiągnęła Wysoka Izba w tym okresie, myślę, że równać się może tylko z najmroczniejszymi czasami poprzednich reżimów. Tym gorzej dla was, bo dzisiaj, jak sądzę, nikt nie przystawia wam lufy rewolweru do skroni - mówię do posłów dziś rządzącej większości - nikt wam nie grozi wywózką na Sybir, nikt was nie wysyła do Oświęcimia, a jednak realizujecie misję zagłady wobec własnego narodu. Dzieci i wojsko to dwa probierze waszej polityki. To są zjawiska o charakterze wojennym. To wy wydaliście wojnę narodowi, wy, rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, ze wsparciem, kontrasygnatą Wysokiej Izby, a także urzędu prezydenckiego. Dzieci poddane kwarantannie, szkoły, w których zaprowadzono reżim skutkujący obniżeniem kondycji psychofizycznej, to jasne, także skutkujący pomieszaniem serc i umysłów, dezinformacją, która jeśli jej celem staje się najmłodsze pokolenie, jest czymś szczególnie strasznym. Kto może robić dzieciom takie rzeczy? Jakieś bestie, ludzkie bestie, Niedzielski i spółka. Tak, to są ci ludzie, którzy niszczą naród polski i niszczą jego nadzieję - najmłodsze pokolenie. I druga tragedia, która powinna dotykać każdego polskiego państwowca - to, co robicie z wojskiem i służbami. To jest bowiem rdzeń państwowości. I właśnie Wojsko Polskie zostało zawirusowane, nomen omen, wirusem uznaniowości w postępowaniu, wirusem nieformalnych nacisków. Nie przyjmujecie do wojska ochotników, bo nie legitymują się papierami, których nielegalnie od nich wymagacie. Relegujecie z wojska dobrych żołnierzy, którzy nie podporządkowują się tej tresurze, którą sami przyjęliście, Bóg z wami, ale którą staracie się też narzucać innym. A zatem wojsko i dzieci. Kogo inne argumenty nie przekonują, niechaj przynajmniej drgnienie sumienia zreflektuje na tej drodze. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo!

W tej sytuacji rząd powinien podjąć zdecydowane działania zmierzające do obniżek podatków, tak żeby ta cena paliwa mogła spaść. Wysokie ceny paliw zagrażają generalnie gospodarce i utrzymywanie ich na tym poziomie jest kontrskuteczne, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. I to jest kolejne uderzenie w kierowców, bo przecież rząd szykuje dzisiaj absurdalny wzrost, jeśli chodzi o mandaty za różne wykroczenia drogowe.

Oni są chyba najbardziej obciążani, jeżeli chodzi o podatki w różnej wysokości, w różnej formule i różnie się nazywające. Ale, jak mówię, tu nie chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo gdyby chodziło o bezpieczeństwo, to rząd podejmowałby zupełnie inne działania. I o jednym z takich działań chcę dzisiaj powiedzieć.

Te bardzo często stosowane przez zarządców dróg minimalne wartości nie pozwalają na swobodne i przede wszystkim bezpieczne przejście przez drogę osób, które mają ograniczoną możliwość poruszania się, bądź też rodzin lub seniorów.

W związku z tym dzisiaj zwracam się do rządu, w szczególności do ministra infrastruktury, o podjęcie działań zmierzających do wydłużenia tych minimalnych czasów przejść.

I to będzie o wiele bardziej skuteczne i o wiele bardziej rozsądne niż karanie kierowców w szerokim zakresie podnoszeniem stawek mandatów do wartości niespotykanych w innych państwach europejskich.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Jesteście bezpieczni, nie zaprzątacie sobie głowy sprawami, które jeszcze parę dni wcześniej polaryzowały i emocjonowały świadków wydarzeń z pogranicza polsko-białoruskiego. Dziś emocje nieco opadły. Spektakularne i, można by powiedzieć, proporcjonalne w nieodpowiedzialności zachowania niektórych polityków i ich akolitów zeszły z wokandy publicznej debaty, ale przecież służba i trud ochrony integralności granic państwa i bezpieczeństwa ojczyzny nie zbladł, stale jest wyzwaniem. Dlatego też zwracam się do wszystkich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz waszych przełożonych, pana komendanta głównego Straży Granicznej gen. dywizji Tomasza Pragi, czy też do bliskich mi funkcjonariuszy, m.in. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. Straży Granicznej Tomasza Michalskiego, z wyrazami uznania i wsparcia za wierność służbie ochrony granic naszej ojczyzny. Jako mieszkaniec Krosna Odrzańskiego, gdzie zlokalizowana jest komendantura Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, z natury rzeczy znam specyfikę waszej służby. Doceniam ją i analizuję od lat także jako socjolog pogranicza. Nie mogę wobec tego, co dokonuje się obecnie w przestrzeni publicznej, czyli wobec próby zdyskredytowania waszej formacji i służby etosu pograniczników, pozostawać biernym. Zbyt ważna jest wasza służba, zbyt obciążająca także w sensie miru domowego rozumianego szeroko zarówno w kontekście wspólnoty ojczyzny i jej bezpieczeństwa, jak i w sensie bardzo osobistym, prywatnym, perspektywy prywatnej, domu własnego, by w momencie gdy plwa się w twarz polskim żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej, nie stanąć w waszej obronie. Wiem, że i bez moich słów wsparcia doskonale dajecie sobie radę. Napawa mnie dumą obserwowanie profesjonalizmu i sprawności działań Straży Granicznej oraz maksymalnej cierpliwości w znoszeniu medialnych manipulacji oraz groteskowych, acz mających swoje znaczenie w urabianiu nastrojów społecznych wybryków niektórych polityków opozycji. Wstyd mi, że zasiadam w tej samej Izbie parlamentarnej z osobami, których czyny, szczególnie te wynikające ze świadomej intencji, godzą w bezpieczeństwo Polski. Bo jeżeli chodzi o tych, którzy robią to z głupoty czy cynicznej kalkulacji: żeby o mnie mówili, to efekt społecznych wyborów. Takich mamy posłów, jakich sobie wybraliśmy. Nie zmienia to postaci rzeczy, że właśnie ci groteskowi, określani także jako pożyteczni idioci, mogą być uznawani jako reprezentatywni dla wspólnoty parlamentarzystów, tylko dlatego że jest o nich głośno, a są jak ślepe narzędzie w rękach sił, które uruchamiają niepożądane działania wobec Polski, której powinni służyć. Współczesność wysoko stawia poprzeczkę zarówno Wojsku Polskiemu, jak i Straży Granicznej. Ufam, że w każdym z możliwych doświadczeń, w jakich się znajdują, najlepiej i najskuteczniej jak to możliwe, chronią integralność i bezpieczeństwo Polski. Niech Pan Bóg was strzeże, a wy strzeżcie nas. Dziękuję bardzo. Pani poseł Monika Falej, klub Lewica. Nie widzę. Pan poseł Piotr Adamowicz. Nie widzę. Pan poseł Fryderyk Kapinos, Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W dniu 3 września br. społeczność miasta Mielca oraz powiatu mieleckiego przeżywała piękną uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Był to wielki i wyjątkowy dzień dla wszystkich obecnych oraz byłych zawodowych strażaków, którzy pełnili swą służbę na ziemi mieleckiej. Przekazany sztandar jest symbolicznym wyrazem uznania ich zasług i trudu włożonego w zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności na przestrzeni lat, gdyż mielecka komenda jest spadkobierczynią i kontynuatorką chlubnych tradycji pożarniczych tego terenu. O tym, jak szczególnym wyróżnieniem dla każdej jednostki służb mundurowych jest sztandar, nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to symbol honoru, wierności i męstwa, będący wielkim powodem do dumy. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu został on przekazany w obecności fundatorów oraz przedstawicieli polskiego parlamentu, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, władz województwa podkarpackiego, władz samorządowych miasta i powiatu mieleckiego oraz wszystkich znamienitych gości i lokalnej społeczności. Miałem zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Nadanie sztandaru miało miejsce w obecnym roku, w 75. rocznicę zawodowego pożarnictwa na ziemi mieleckiej. Jego historia to czas rozpoczęty powołaniem przez zarząd miasta w dniu 26 stycznia 1946 r. Pogotowia Straży Pożarnej w Mielcu.

Warto pamiętać i przypominać o tych wszystkich zdarzeniach, gdzie zwykle jako jedni z pierwszych meldowali się na akcjach ratunkowych, spiesząc ze wspomnianą pomocą w obliczu pożarów, wypadków i klęsk żywiołowych. Lokalnej społeczności strażacy dali poczucie bezpieczeństwa, cieszą się szacunkiem i zaufaniem. Realizując swoją zawodową misję, w piękny sposób pokazują etos strażackiej pracy, prawdziwą solidarność i pomoc drugiemu człowiekowi. Za to wszystko pragnę serdecznie podziękować obecnym oraz byłym strażakom zawodowym pracującym na ziemi mieleckiej. Na kolejne lata życzę również bezpiecznej służby - Panu Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Pani poseł Joanna Fabisiak. Nie ma. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Zapraszam, pani poseł.

Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Pan poseł Fryderyk Kapinos wygłosił oświadczenie w sprawie 75-lecia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, będąc przewodniczącym społecznego komitety ufundowania sztandaru. Jako członek społecznego komitetu ufundowania sztandaru, chciałabym się do tych życzeń przyłączyć, przyłączyć się do gratulacji z okazji 75. rocznicy powstania i ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, okazując szacunek dla wszystkich druhen i druhów, którzy przez te lata służyli społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że zawsze będziemy pamiętać o tych, którzy odeszli i którzy zasługują na najwyższe uznanie. Po tym świętowaniu chciałabym wygłosić dwa oświadczenia.

Doskonale wiemy, że nie wszyscy spokojnie śpią. Doskonale wiemy, że niektórzy nie śpią w swoich domach, dlatego że upominają się o ważne sprawy dla nas, pacjentów, o to, żeby ochrona zdrowia funkcjonowała poprawnie. Tekst naszego dezyderatu był następujący: Komisja Zdrowia, dostrzegając znaczenie prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, niniejszym wnosi o pilne podjęcie rozmów przez pana premiera z protestującymi przedstawicielami zawodów medycznych. Z uwagi na upływające kolejne dni strajku oraz nieudolne działania ministra zdrowia rozpoczęcie dialogu osobiście przez pana premiera wydaje się konieczne do zażegnania poważnego kryzysu w systemie opieki zdrowotnej, z którym mamy obecnie do czynienia. W ocenie Komisji Zdrowia podjęcie przez prezesa Rady Ministrów dialogu z przedstawicielami zawodów medycznych uznać należy jako niezbędny środek do zapewnienia lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym warunków pracy gwarantujących bezpieczne i niczym niezakłócone realizowanie świadczeń medycznych. Komisja Zdrowia wyraża głębokie zaniepokojenie aktualną sytuacją w systemie ochrony zdrowia oraz problemami, z którymi borykają się pracownicy podmiotów leczniczych. Wobec powyższego podjęcie przez pana premiera pilnych działań w tym zakresie wydaje się wysoce uzasadnione. Jest mi wstyd, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Komisji Zdrowia głosowali przeciwko przyjęciu tego Jednak nie wszyscy mogą spokojnie spać. Mój drugi apel do premiera, prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego jest w sprawie walki z ASF i pomocy rolnikom z powiatu mieleckiego.

Takich ognisk obecnie jest ponad 30. Rolnicy mają problem ze zbyciem zdrowych sztuk ze strefy czerwonej. Nie ma odpowiedniego wsparcia w tej sprawie ze strony rządu. Apelują do premiera Morawieckiego o podjęcie pilnych działań wszystkich służb, które mogą pomóc rolnikom. Sprawa jest niezwykle ważna, sprawa jest niezwykle pilna. Rolnicy czekają, panie premierze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Teresa Hałas, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z wielkim żalem informuję, że w dniu 12 września br. odeszła od nas pani Janina Kalinowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, ocalała ze zbrodni wołyńskiej, wielka wojowniczka o prawdę rzezi wołyńskiej i Kresów Wschodnich. Zawsze walczyła o pamięć o Polakach pomordowanych na Wołyniu oraz o nazwanie ten bestialskiej zbrodni ludobójstwem. Pani Janina Kalinowska była nam niezwykle bliska. Od lat Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” aktywnie wspiera działania stowarzyszenia w upamiętnianiu ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach pomordowanych na Wołyniu i osób, które przeżyły tę straszną tragedię. Janina Kalinowska urodziła się prawdopodobnie w 1935 r. Data je urodzin została ustalona przez sąd, ona sama jej nie znała. Wychowywała się w kolonii Funduma, wsi polskiej wojskowych osadników w powiecie włodzimierskim, gdzie mieszkała z rodziną. 11 lipca 1943 r. ukraińscy nacjonaliści, frakcja Stepana Bandery oraz jej zbrojne ramię - Ukraińska Powstańcza Armia, napadli na tę miejscowość, mordując w okrutny sposób niemal wszystkich mieszkańców w liczbie 260 osób. Zamordowali również jej rodziców i 2-letniego brata. Jak później podkreślała: miałam szczęście, bo moi rodzice i brat nie zginęli od siekiery, wideł ani innych narzędziach zbrodni, tylko zostali rozstrzelani. Niewiele z tego pamiętam. Kiedy padły strzały, mama, upadając, musiała pociągnąć mnie za sobą. Później ukrył ją sąsiad, znajomy jej ojca zaprowadził ją do Włodzimierza, gdzie zaopiekowała się nią polska rodzina, z którą pani Janina została zesłana na roboty do Niemiec. Od maja 1945 r. jako sierota po wojnie przebywała w obozie przejściowym w Niemczech. W 1948 r. rodzina, u której przebywała, przywiozła ją do Polski. Trafiła do domu dziecka w Zamościu prowadzonego przez Polski Komitet Opieki Społecznej. Życiowym mottem pani Janiny Kalinowskiej była pamięć i prawda o Wołyniu. Przekazywała świadectwo smutnej i tragicznej prawdy o Polakach zamordowanych z największym okrucieństwem, jakie poznał świat. W ramach Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu organizowała szereg wyjazdów na Wołyń, aby przy symbolicznych krzyżach ustawionych na miejscach masowych mordów były zapalane znicze i składane kwiaty. Podejmowała również szereg inicjatyw, aby uczcić pamięć Polaków pomordowanych na Wołyniu. Prowadzone przez panią Janinę Kalinowską Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu zostało uhonorowane dwoma niezwykle ważnymi tytułami: Kustosza Pamięci Narodowej w 2013 r. oraz Strażnika Pamięci w 2019 r. Jej świadectwo było inspiracją do powstania wielu książek, artykułów prasowych, felietonów i filmów. Wierzę, że jej życiowa droga pomoże przyszłym pokoleniom pójść w jej ślady i kontynuować dzieło pamięci, a także spojrzeć na Wołyń naszych przodków jako na piękną krainę w dorzeczu Bugu, gdzie tylko krzyże, opuszczone cmentarze i miejsca przypominają o polskich gospodarzach. Ona zaś sama pozostanie na zawsze w naszej życzliwej pamięci jako ambasador ziemi wołyńskiej i Kresów Wschodnich. Pani poseł Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W Lubaczowie 17 września odbywają się uroczystości związane z 50. rocznicą istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie.

Obecny patron, którego mural zostanie właśnie odsłonięty, zapisał się chwalebną kartą w historii polskiej jako obrońca Lubaczowa przed Ukraińcami w 1918 r., a przede wszystkim jako dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża w kampanii wrześniowej w 1939 r. Za zasługi bojowe podczas I wojny światowej został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Był to przede wszystkim wielki człowiek, stawiany do dzisiaj przez wielu przez swoje czyny za wzór żołnierza, obywatela i dowódcy. Dzięki nim zapisał się na zawsze w pamięci potomnych i zajął jakże zasłużone miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Lądowa Obrona Wybrzeża pod dowództwem płk. Stanisława Dąbka należy do zaszczytnych tradycji Wojska Polskiego. Wieczorem 19 września 1939 r. w rejonie Babich Dołów w obliczu nieuchronnej klęski odebrał sobie życie strzałem w głowę, nakazując zarazem niezwłoczne zaprzestanie walki po jego śmierci. Dąbka na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Redłowie została odsłonięta płyta nagrobna z wyrytymi słowami „Pokażę Wam jak Polak walczy i umiera” W 1964 r. otrzymał pośmiertnie awans na stopień generała brygady nadany mu przez gen. Władysława Andersa, a w 1969 r. przez prezydenta na uchodźstwie Augusta Zalewskiego. Uroczystość 50-lecia szkoły jest dla kierownictwa szkoły, grona pedagogicznego, rodziców, uczniów i całej społeczności miasta Lubaczowa wydarzeniem wyjątkowym. Na przestrzeni tych 50 lat ta szkoła wydała wielu znakomitych wychowanków, odgrywających dziś ważną rolę w regionie, w kraju i za granicą. Jest to okres na tyle długi, by przywołać wspomnienia o pięknych kartach historii tej szkoły, w którą na trwale wpisała się osoba jej patrona. W dobie ciągłych poszukiwań autorytetów moralnych niech stanie się ona wzorem do naśladowania dla wszystkich pokoleń. W tym szczególnym dniu chciałabym złożyć słowa uznania dla pana dyrektora, wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi za dotychczasową działalność, za wytrwałość, serce i oddanie, z jakim wykonujecie państwo swoją codzienną pracę. Życzę jednocześnie satysfakcji z wykonywania codziennej pracy. Bądźcie dla swoich uczniów autorytetami, niech każdy dzień przynosi wam radość i zadowolenie. Życzę dalszych wspaniałych osiągnięć, a uczniom sukcesów i wytrwałości w rozwijaniu zainteresowań. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Wysoka Izbo! Wytrwali Parlamentarzyści! Pozwólcie, szanowni państwo, że opowiem dzisiaj o pewnym fenomenie, którym jest susza w Polsce.

Co to spowodowało, szanowni państwo?

Jeden powiat w województwie zachodniopomorskim. Ale co się stało, szanowni państwo? Rolnik musi złożyć wniosek do agencji restrukturyzacji.

Można więc powiedzieć, że w Polsce można zlikwidować suszę aplikacją. To nie była pierwsza susza. To była kolejna susza na Pomorzu Zachodnim, dokładnie czwarta, a 5 lat temu były nawalne deszcze. I jest pytanie, jak długo będziemy jeszcze udawać, że tego problemu nie ma, bo on jest. Tylko kiedyś było o tyle lepiej, szanowni państwo, że wojewoda wysyłał komisje z ośrodków doradztwa rolniczego wraz z przedstawicielami gmin i rolników i oni szacowali.

Dlatego, panie ministrze, panie niemy ministrze - bo, jak państwo wiecie, już prawie rok pan minister jest, ale tu, w tym miejscu go jeszcze nie było - może wreszcie trzeba wziąć się za tę aplikację, wyrzucić ją do kosza, posłuchać tych ludzi, którzy dzisiaj mówią o realnych stratach. Panie ministrze, apeluję do pana, żeby naprawdę zastanowić się nad zmianą systemu szacowania, być może nad powrotem do starego systemu szacowania strat suszowych, bo to, co wprowadziliście państwo, nie działa i jest szkodliwe dla polskiego rolnictwa.

Wyglądało to na początku dobrze, później wyglądało fatalnie. Nie mówię o jakości, nie mówię o innych parametrach tego zboża.

Tu jeszcze raz, szanowni państwo, być może też za państwa pośrednictwem, proszę, by pozbyć się tego, a też pomóc tym rolnikom, którym można jeszcze w jakikolwiek sposób pomóc.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.